W zeszłym tygodniu na tajnym posiedzeniu Sejmu doszło do bezpodstawnego zawyżenia klauzuli tajności. Dlatego na podstawie ustawy o informacji niejawnej, art. 9, żądamy ujawnienia stenogramu z tego posiedzenia po to, żeby wszyscy obywatele mogli usłyszeć i zobaczyć, przeczytać ten bełkot, który mieliśmy okazję usłyszeć w zeszłym tygodniu. Oprócz tego wnoszę o przerwę i - po tej przerwie - pełną informację jawną premiera Morawieckiego o aferze mailowej, informację o tym, czy ABW wszczęła kontrolę poświadczenia bezpieczeństwa ministra Dworczyka. Wszyscy doskonale wiecie, że to jest afera, która paraliżuje funkcjonowanie państwa. że dysponenci tych maili będą. codziennie terroryzować prace rządu kolejnymi informacjami z waszych prywatnych maili. Nie ma innego wyjścia niż dymisja [[Oklaski]] osób zamieszanych w tę aferę. A poza wszystkim odwołajcie dzisiaj ministra Kamińskiego, to przestaniecie się bać korzystać.

Nie ma podstawy prawnej do odtajnienia obrad, panie pośle. Dziękuję. To nie dotyczy tego wniosku o utajnienie obrad, panie pośle. Proszę przeczytać sobie konstytucję, panie pośle. Wysoka Izbo! Dzisiaj związki zawodowe PGE z OPZZ zaapelowały do nas, do 460 posłów, żebyśmy mówili jednym głosem w sprawie Turowa. Jest rzeczywiście tak, że jeżeli pan wicepremier Jacek Sasin jedzie i rozwiązuje sprawę Turowa, to na pewno wniosek o jego odwołanie nie pomaga Rzeczypospolitej. I to jest wilcze prawo opozycji składać taki wniosek, ale apeluję do pana przewodniczącego Borysa Budki, aby ten wniosek dzisiaj wycofał do czasu zakończenia sprawy w Turowie, ponieważ pana argumentacja niestety zostanie. To nie jest czas na debaty polityczne na ten temat, porozmawiajmy o tym po zakończeniu sprawy w Turowie. Dlatego wspieram zdecydowanie związki zawodowe z OPZZ i apeluję jednak o lojalność wobec Rzeczypospolitej. Wtedy kiedy atakowane jest polskie państwo, mówmy jednym głosem. Panie przewodniczący, ja panu dzisiaj.

Proszę bardzo, pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Pani Marszałek! Składam wniosek formalny o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i włączenie do porządku obrad informacji ministra edukacji i nauki i wyjaśnień, które należą się Wysokiej Izbie. Wyjaśnień, dlaczego po raz kolejny w dniu dzisiejszym minister edukacji dopuścił się szczucia i obrażania obywateli legalnie realizujących swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń, [[Oklaski]] dlaczego nazwał osoby uczestniczące w sobotniej paradzie równości. osobami nienormalnymi, dlaczego minister edukacji szczuje także na uczniów, także na uczniów LGBT+, którzy również uczestniczyli w tej paradzie. Wyjaśnień wymagają także. informacje, które docierają do Wysokiej Izby, że minister Przemysław Czarnek próbuje podporządkować sobie w sposób radykalny i totalny funkcjonowanie każdej szkoły. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł, dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! do normalności. Ale do normalności nie wraca Lewica ani pani poseł. Pani poseł, ja mam wniosek formalny, żeby pani raz jeszcze wysłuchała mojej wypowiedzi i przestała kłamać bezczelnie. Polacy widzą. Polacy widzą waszą narrację, pełną. chamstwa, pełną kłamstwa, fałszowania rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ dwa razy padł ten sam wniosek, a nie ma takiej możliwości, przegłosujemy wniosek o przerwę. Bardzo proszę. pani zgłosiła go po raz kolejny. pani go zgłosiła po raz kolejny niezgodnie z regulaminem, więc. przegłosujemy wniosek o przerwę, żeby nie było kolejnych wniosków o to samo. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za chwileczkę, najpierw przegłosujemy wniosek formalny, panie pośle. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wniosek nie uzyskał większości. Z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Panie Ministrze! Powiedział pan słowa następujące: Przecież wszyscy Polacy widzą, co się dzieje na ulicach, i wiedzą, na czym polega tolerancja. Przecież to, co się tam działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i równością. Polacy widzą, kto jest normalny, a kto nie. Panie Ministrze! Panie ministrze, nie jest pana prawem, nie jest pana kompetencją odmawianie uczniom, młodzieży, nauczycielom ani żadnej [[Oklaski]] mniejszości korzystania, prawa do korzystania. z konstytucyjnego prawa do gromadzenia się i wyrażania własnych poglądów.

Pani poseł, dziękuję. Proszę, z wnioskiem formalnym pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja.

Przypominam, panie pośle, że wniosek o przerwę już przegłosowaliśmy. Może mam trochę poważniejszy wniosek niż poprzedni. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Ja zgłaszam też wniosek o przerwę w celu zwołania Konwentu Seniorów. w bardzo konkretnej sprawie, w celu uzupełnienia porządku obrad o informację ministra obrony narodowej w sprawie rozporządzenia z 21 maja, którym to rozporządzeniem de facto zabrał jedyne źródło utrzymania setkom polskich rybaków z Wybrzeża i Zalewu Wiślanego. Chciałbym, żeby pan minister odpowiedział nam, jak teraz ci rybacy mają żyć, skoro nie było dla nich nawet odszkodowania, a łowiska są zamknięte. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Wysoka Izbo! Składam wniosek o odroczenie obrad do jutra, do godz. 9, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego informacji pana premiera na temat tego, dlaczego dwie skrajne organizacje związane z panem Robertem Bąkiewiczem, czyli stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, otrzymały w sumie 3 mln publicznych pieniędzy na swoją działalność. Szanowna Pani Marszałek! Nie może być tak, że Polacy chcą rozwiązania Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” a państwo z Funduszu Patriotycznego, o który wnioskował pan premier i pan wicepremier Gliński, po prostu sponsorujecie zwykłych chuliganów. Tak po prostu nie może być. Dziękuję, pani poseł. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przypominam, że Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni złożył wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek - obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat decyzji rządu w sprawie przyjęcia 2050 roku jako daty granicznej osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Proszę dać mi powiedzieć, jakie są wyniki posiedzenia. Konwentu i moich decyzji. Mamy nowy system, wróciliśmy do normalnego, stacjonarnego głosowania, w związku z tym ja też muszę wiedzieć, czy od razu mogę powiedzieć „dziękuję” i są wyniki, czy musimy chwilę czekać. Uznaję to głosowanie. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie neutralności klimatycznej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy u wszystkich państwa działa? Nikt nie zgłasza problemów, tak?

Sejm wniosek odrzucił. Proszę panią poseł sekretarz o odczytanie komunikatów.

Proszę państwa, tylko krótki komunikat. Ten punkt, który przegłosowaliśmy w poprzednim głosowaniu, będzie rozpatrywany jutro na koniec posiedzenia Sejmu. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1188 i 1212) Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1188. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, w dniu 19 maja 2021 r. powyższy projekt ustawy. Bardzo proszę państwa posłów, którzy nie biorą udziału w tej części posiedzenia, o opuszczenie sali i pozwolenie pani sprawozdawcy na przedstawienie uzasadnienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani marszałek.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych i jego racjonalizacja, w tym wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje. Chodzi o ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty. I tak: ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej - w aktualnym stanie prawnym powstają wątpliwości interpretacyjne w stosunku do osób prowadzących działalność będących wspólnikami spółek: jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.; proponuje się uzależnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych od statusu wspólnika; ujednolicenie zasad wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w systemie ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia tzw. służb mundurowych; ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego; uproszczenie zasad podlegania ubezpieczeniom dobrowolnym; zrównanie form wypłaty świadczeń długoterminowych; prawo do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez zakład i do potrącania świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych zasiłków oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń; uproszczenie procedury przy dokumentowaniu prawa do rodzicielskich świadczeń uzupełniających; elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczeń A1. Ustawa obejmuje również zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń. I tak, inny sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które występują o emeryturę w czerwcu. To bardzo oczekiwana zmiana. Proponuje się, by na stałe wprowadzić rozwiązanie przyjęte na 2020 r. dotyczące zasad ustalania wysokości nowych emerytur przyznawanych w czerwcu, począwszy od roku 2021, w tym waloryzacji kapitału początkowego i składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju br., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Proponuje się zwiększenie zakresu ochrony rentowej osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna bądź po ustaniu prawa do tych świadczeń. Proponuje się ujednolicenie przepisów m.in. w zakresie przeliczania emerytur z tzw. starego i nowego systemu emerytów kontynuujących aktywność zawodową; zmianę zasad zawieszenia renty socjalnej w przypadku wykonywania aktywności zawodowej; zmianę w zakresie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Przepisy, które zawarte są w ustawie, mają usprawnić obsługę i uporządkować działania płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych. Proponuje się ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczonych do lat 5; zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek nienaliczania odsetek z tytułu składek z przyczyn leżących po stronie zakładu i wydawania zaświadczeń o niezaleganiu spadkobiercom. Proponuje się modyfikację pojęcia „rodzaj działalności według PKD”, a także obowiązek założenia PUE przez wszystkich płatników składek. Jeżeli chodzi o usprawnienie obsługi prowadzonych rozliczeń z płatnikami składek, proponuje się wprowadzenie przepisu jednoznacznie definiującego, jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy, a zatem jakie wypadki pracodawca powinien ujmować w informacji ZUS IWA. Brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadkach przekształceń, łączenia lub podziału płatników składek. Proponuje się doprecyzowanie sposobu ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez płatnika w okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania z urzędu statystycznego zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD.

I tak, proponuje się likwidację funduszu rezerwowego. Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów FUS. Tryb dokonywania i zatwierdzania zmian w planie finansowym zakładu. Proponuje się wprowadzenie możliwości umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje się nowe zasady powoływania Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalił załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1188 i 1212. Teraz przekażę główne zmiany. Projekt ustawy zawiera m.in. następujące propozycje. Ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie od dnia wpisania spółek do KRS-u albo od dnia nabycia udziału w spółce, natomiast ustanie z dniem wykreślenia spółki z KRS-u albo zbycia wszystkich udziałów w spółce z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności spółki. Następna propozycja zmiany to uproszczenie zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom. Podleganie ubezpieczeniom dobrowolnym następować będzie od dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia do dnia wskazanego w formularzu wyrejestrowania. Przy czym objęcie lub ustanie ubezpieczenia dobrowolnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż odpowiednie zgłoszenie, wyrejestrowanie zostanie złożone w ZUS. Zgłoszona osoba będzie podlegać temu ubezpieczeniu nawet w przypadku opłacenia składki po terminie lub nieopłacenia jej wcale. Będzie istniała możliwość ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie, a w przypadku osób, których niezdolność do pracy zaistnieje w okresie, w którym będą miały one zaległości z tytułu składek, nowo wprowadzone regulacje umożliwią ubieganie się o świadczenie po spłacie zadłużenia na zasadach analogicznych jak w przypadku świadczeń z ubezpieczeń wypadkowych. Potrącenie z opłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłaconych przez ZUS będzie prowadzone przez zminimalizowanie kosztów dochodzenia. Doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia zachodzą przesłanki do uznania świadczeń za nienależnie pobrane, ZUS wydaje decyzje odmawiające prawa do zasiłku i zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku.

Będą nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed przerwą i po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Nie zmieni się długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia - wynosi on nadal co do zasady 182 dni i 270 dni w przypadku niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy. Skróceniu ulegnie natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia - przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni. Nowe zasady będą dotyczyły powoływania Rady Nadzorczej ZUS.

Obecnie zwolnieni z obowiązku zakładania profilu informacyjnego ZUS są pracodawcy zatrudniający do pięciu osób.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie m.in.: zasad przyznawania emerytur czerwcowych, zasad wypłacania zasiłków chorobowych, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób będących wspólnikami spółek jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o., zasad przeliczania emerytur z tzw. starego i nowego systemu emerytów kontynuujących aktywność zawodową oraz likwidacji funduszu rezerwowego. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. Pani Marszałek! Przedmiotowa ustawa zakłada skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia ze 182 dni do 91 dni. Czy projektodawcy konsultowali ten przepis ze służbami medycznymi? Czy w okresie 3 miesięcy jest możliwość wyleczenia depresji, która powstała na skutek rozwiązania stosunku pracy? Ustawa przewiduje również w stosunku do okresów niezdolności do pracy powstałej po przerwie nieprzekraczającej 60 dni od ostatniej niezdolności do pracy zaliczanie tych okresów do jednego okresu zasiłkowego, nawet wtedy gdy niezdolność do pracy przed przerwą i po przerwie była spowodowana inną jednostką chorobową. Wyobraźmy sobie teraz sytuację: pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu złamania kości udowej - skomplikowana choroba - wykorzystał pełny okres zasiłkowy 182 dni, po miesiącu okazało się, że wykryto u niego nowotwór. Drodzy państwo, taka osoba nie skorzysta już z prawa do zasiłku chorobowego, bo rząd dzisiaj chce przepchnąć ograniczenia skracające okresy zasiłkowe. Przepis ten jest wyjątkowo nieprzemyślany i ukierunkowany jedynie na oszczędności. W imieniu klubu Koalicja Obywatelska złożę w tej sprawie poprawkę. Kolejna zmiana.

Czy rząd zastanawiał się nad tym, że w czasie po pandemii wiele firm odbija się po kryzysie, a wy chcecie obciążyć je dodatkowymi kosztami? Jak będzie wyglądać składka zdrowotna, gdy wprowadzony zostanie Nowy Ład? Coraz częściej mówicie o emeryturze obywatelskiej, w Krajowym Planie Odbudowy mówicie o dłuższej aktywności zawodowej. Szanowni państwo, niech rząd podejmie wreszcie debatę, niech zaprosi ekspertów, skorzysta z nauki i badań naukowych i zaproponuje coś jasnego i czytelnego dla obywatela. W tym miejscu również składam poprawkę. W odniesieniu do nowych zasad przyznawania emerytur dla osób, których wnioski zostały złożone w ZUS w czerwcu, jest to dobre rozwiązanie.

W związku z czym składam poprawkę dotyczącą możliwości przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad dla osób, które nabyły prawo do emerytury w czerwcu od 2009 r. do 2019 r. Poprawka ta wyjdzie naprzeciw zasadzie równego traktowania, a emeryci będą mieć poczucie sprawiedliwości. Projektowane zmiany przewidują ujednolicenie możliwości przeliczania emerytur przyznanych ze starego systemu i nowego systemu. Zmiany te spowodują, że pracujący emeryt, który pobiera emeryturę ze starego systemu, będzie mógł przeliczyć swoje świadczenie raz w roku, a nie, jak do tej pory, raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. Zmiany te są niekorzystne dla aktywnych emerytów. W tym miejscu nasuwa się pytanie: Czy rząd dąży do podwyższania emerytur dla aktywnych zawodowo emerytów, czy zablokuje im tym samym możliwość podwyższania świadczeń? Tym samym zniechęca ich do aktywności i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Tutaj również złożymy poprawkę. Proponowany projekt ustawy przewiduje likwidację funduszu rezerwowego. Fundusz ten jest stworzony jako fundusz rezerwowy dla funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego, a tworzony jest przez ZUS ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku bankowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W uzasadnieniu tej zmiany czytamy, że występuje ciągły niedobór środków w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i istnieje konieczność dotowania tego funduszu ze środków z budżetu państwa. W mojej ocenie likwidacja tego funduszu spowoduje zaciemnienie przejrzystości. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska poprze przedmiotowy projekt ustawy, ale pod warunkiem że zostaną przyjęte nasze poprawki. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica.

Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rząd po raz pierwszy otwarcie mówi, że trzeba oszczędzać na tych, którym zdrowie szwankuje. Przepisy zaproponowane w tej ustawie nie uzyskają poparcia klubu parlamentarnego Lewicy. Stoimy tutaj na stanowisku wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Myślę, że rząd nie wsłuchuje się w opinie partnerów społecznych, którzy w sposób jednoznaczny odrzucają próbę ograniczenia właśnie świadczeń chorobowych. To, co państwo proponujecie, oznacza również ograniczenie, skrócenie okresu ochronnego przed rozwiązaniem stosunku pracy w kontekście art. 53 Kodeksu pracy. Mamy w tej sprawie poprawki. Jeśli chcemy przyjąć tę ustawę - to prawda: ważną, porządkującą pewne kwestie, regulującą, doprecyzowującą - powinniśmy jednak szukać porozumienia. Czy w okresie pandemii, tak trudnym okresie wychodzenia z niej - mam na myśli teraz kryzys gospodarczy - trzeba również wprowadzać tak restrykcyjne zmiany, tak niekorzystne dla ubezpieczonych, tych, którzy korzystają z zasiłków chorobowych? Uważamy, że nie jest to dobry okres. Rozwiązania zawarte w ustawie, dotyczące chociażby kwestii ujednolicenia przepisów w zakresie przeliczania emerytur z tzw. starego i nowego systemu emerytalnego dla tych, którzy kontynuują aktywność zawodową i rozliczają świadczenia, są też proponowane w dół, czyli będzie gorzej. W tej chwili mają oni możliwość po zakończeniu każdego kwartału, cztery razy w roku, złożyć wniosek o rozliczenie. Rząd mówi: ujednolićmy te dwa systemy, stary i nowy, i zróbmy to raz w roku. To odbędzie się po raz kolejny z niekorzyścią dla tych, którzy kontynuują aktywność zawodową.

Dziś według danych ZUS-u 81% świadczeniobiorców korzysta z systemu bankowego, czyli można powiedzieć: dokonywane są przelewy. W uzasadnieniu projektu rządowego pokazywane są rodzaje tych świadczeń, np. te wprowadzone dla matek 4+, niecałe 37% z nich korzysta z systemu bankowego. Musimy brać pod uwagę, że wielu świadczeniobiorców jest niesamodzielnych, mieszka w środowiskach małych, wiejskich, gdzie nie ma dostępu do Internetu. Dzisiaj mówienie o tym, że trzeba ich przymusić do tego, aby swoje konstytucyjne prawo do emerytury mogli odebrać przez posiadanie właśnie tego konta i takie rozliczanie, uważamy za niewłaściwe.

Ale kiedy mamy jednorazowe świadczenie, tzw. czternastą emeryturę, zróżnicowaną, wówczas powinniśmy dostarczać tę decyzję również na wniosek samego ubezpieczonego.

Tutaj mówi się o dwóch służbach, mianowicie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To też uważamy za nieuzasadnione. Konkludując, przedstawiam stosowne poprawki do projektu ustawy. Jednoznacznie mówimy o tym, że nie wolno oszczędzać na osobach, które są w trudnej sytuacji i korzystają z chorobowego. Jeśli poprawki nie uzyskają akceptacji Wysokiego Sejmu, klub będzie głosował przeciw tej ustawie. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Państwo Parlamentarzyści! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam przyjemność przedstawić państwu stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1188. Po analizie tej ustawy i konsultacjach zarówno z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jak i z przedsiębiorcami, uważamy, że proponowane rozwiązania w większości są do zaakceptowania. Jest jednak wiele przepisów projektowanej ustawy, które budzą poważne wątpliwości. Chodzi np. o przepis dotyczący wypłat świadczeń długoterminowych w formie bezgotówkowej oraz o tzw. emerytury czerwcowe. Propozycja wprowadzenia obligatoryjności bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych jest co do zasady oczywiście słuszna - jest bezpieczniejsza dla świadczeniobiorców i tańsza. Należy jednak zauważyć, że w grupie świadczeniobiorców są osoby, które z różnych przyczyn wolą jednak tradycyjną formę dostarczania świadczeń. Są osoby, które nie miały, nie mają i nie będą miały konta.

Tutaj rodzi się pytanie: Jakie kryteria i jakie okoliczności ustawodawca ma na myśli? Uważam, że należy pozostawić możliwość wyboru samym zainteresowanym.

Proponowany projekt przewiduje wprowadzenie powyższej zasady na stałe, jednak tylko w stosunku do emerytur przyznawanych od czerwca br. Rozwiązanie to nie uwzględnia sytuacji osób pobierających emerytury czerwcowe z lat ubiegłych, które pozostaną trwale obniżone. Jest to krzywdzące dla tej grupy osób i budzi wątpliwości konstytucyjne. Przedmiotowa ustawa zakłada zmniejszenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia ze 182 dni do 91 dni.

Czytając te zapisy, nasuwa się nieodparte wrażenie, że rząd nerwowo szuka pieniędzy, ponieważ nijak nie spina się budżet funduszu ZUS. Ustawa ma ułatwić ZUS ściągalność składek z tytułu nienależności pobranych świadczeń. Stracą na tym oczywiście Polacy. Pamiętajmy, że mamy już drugi rok pandemii. W tym czasie wiele polskich firm upadło. Polacy starają się jak mogą wiązać koniec z końcem. Przypominam, że w zamrażarce sejmowej od kilku lat leżą projekty naszych ustaw zgłoszonych przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej również nie miała maseczki.

Chciałbym skupić się na kilku najważniejszych. Po pierwsze, zdążyliście już zabić spółki komandytowe.

Doprowadziliście do tego. Jakąś formą ucieczki od tego było prowadzenie spółki. Właśnie wprowadzacie opodatkowanie, ozusowanie wspólników, więc jest to działanie jednoznacznie przeciwko ludziom, którzy prowadzą jakąkolwiek własną działalność. Jak każdy rząd, jak wasi poprzednicy po prostu nienawidzicie ludzi, którzy potrafią coś zrobić samemu i nie muszą pracować ani w spółce Skarbu Państwa, ani w jakimś urzędzie. Druga rzecz.

Wiele osób z tej formy nie korzysta.

Będzie to więc wielka operacja zmuszania ludzi do tego, żeby rejestrowali się w systemie, w którym ich w tym momencie nie ma i nie byłoby, gdybyście ich do tego nie zmusili. Kolejna rzecz to skrócenie okresu ubezpieczenia w przypadku niezdolności do pracy z 6 do 3 miesięcy.

Tak że brawo dla was.

Kolejna rzecz to zmiana sposobu naliczania składek. Chciałbym powiedzieć: jest taka święta zasada - prawo nie działa wstecz.

Umowę, która oczywiście nie jest pisana, nie jest w żaden sposób zakontraktowana; tak sobie po prostu ten ZUS nielegalnie działa, w taki właśnie sposób, bo w prywatnym sektorze trzeba jednak coś podpisać, na coś się zgodzić.

Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby coś takiego robić, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas do tego, że robi takie rzeczy, na które żaden inny rząd by sobie nie pozwolił.

Po prostu nie mielibyście po takim ruchu klientów, ponieważ gdyby prywatna firma, w której się ubezpieczam, w której składam swoje pieniądze na dodatkowe ubezpieczenia, poinformowała mnie, że z dnia na dzień zmieniają się, skrajnie źle, warunki przetrzymywania moich pieniędzy na ich kontach, to bym te pieniądze po prostu odebrał. Wy natomiast Polakom na to nie pozwalacie. Dziękuję bardzo. Przypominam: wszyscy na sali muszą mieć maseczki.

Panie i Panowie Posłowie! Ustawa przewiduje pewien rodzaj udogodnień, ujednolicenia zasad, ale z drugiej strony wprowadza też wiele dość kontrowersyjnych zapisów; o niektórych mówili moi poprzednicy. W projekcie proponuje się m.in. objęcie ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, niezależnie od okoliczności, w których funkcjonują. Rozumiem, że to jest sposób Prawa i Sprawiedliwości na uzupełnienie kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie, w starym systemie emerytalnym, emeryt i rencista wykonujący pracę zarobkową i z tego tytułu podlegający ubezpieczeniu może zgłosić cztery razy w roku wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych. Modyfikujecie te przepisy i proponujecie, by taki wniosek można było złożyć raz w roku, co spowoduje zrównanie przepisów w starym i nowym systemie emerytalnym.

I najbardziej kontrowersyjny przepis. Projektowane zmiany przewidują też nowe zasady zaliczania okresów niezdolności do pracy. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed przerwą i po przerwie, jeżeli ta przerwa nie jest dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność nie występuje w okresie ciąży. Nie zmieni się długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia i on dalej będzie wynosić 182 dni, ale już skróceniu ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. To chyba nie są czasy na wprowadzenie tego typu zmian. Jak rozpoznać chorego w trakcie ubezpieczenia i chorego po upływie okresu ubezpieczenia.

Tego typu rozwiązania budzą wątpliwości dotyczące ich wpływu na osoby uprawnione, zarówno w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. W uzasadnieniu nie ma odniesienia w tym zakresie. W projekcie wprowadza się także potrącenie, a polega to na tym, że składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata nieopłacone w terminie będą potrącane ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To też budzi nasze wątpliwości. Po wprowadzeniu tej zmiany nie będzie ważne, czy płatnik składek zapłacił je czy też nie, ale to czy płatnik składek wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych.

Mam kilka poprawek i oczywiście od przyjęcia tych poprawek, ale także tych zmian, o których mówili poprzednicy, będziemy uzależniać nasze poparcie dla tej ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Określam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Pierwszy pan poseł Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W świetle prac prowadzonych nad zmianą przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym pragnę zapytać, i prosić o wyjaśnienie, czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzająca składki ubezpieczeniowe do ZUS-u, a jednocześnie posiadająca dużą działkę na terenach wiejskich, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, nadal ma obowiązek opłacać składki ubezpieczeniowe w obu firmach, to znaczy w ZUS-ie i w KRUS-ie. Czy w przypadku odprowadzania składek do obu firm ubezpieczeń społecznych, do ZUS-u i do KRUS-u, ubezpieczony może w przyszłości liczyć na wypłatę świadczeń emerytalnych pochodzących z obu firm czy tylko z jednej?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Znam pana jako działacza związkowego prezentującego swe poglądy tutaj, w tej Wysokiej Izbie, który w jednoznaczny sposób opowiadał się za tym, aby ochrona pracowników wynikająca z Kodeksu pracy była na odpowiednim poziomie. Natomiast tutaj państwo proponujecie rozwiązania dotyczące jednolitego liczenia czasu, 60 dni, co jest związane z ochroną wynikającą z Kodeksu pracy oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czyli to rozwiązanie pogorszy sytuację, jeśli chodzi o ochronę stosunku pracy. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Hanajczyk, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dla mnie osobiście to dość zaskakujący projekt, ale zaskakujący w wydaniu autora, czyli PiS, partii, która jest bardzo populistyczna, bardzo prosocjalna. Rozumiem, że te rozwiązania muszą wybrzmieć również w środkach publicznych, bo pewno dla wielu Polaków będą dość zaskakujące. Są rozwiązania, które należy pochwalić, natomiast zupełnie dla mnie niezrozumiały jest czas wprowadzania tych rozwiązań. Osobiście znam wiele osób, które po pandemii, po przejściu choroby COVID-owej z jednej strony bardzo się obawiają utraty zatrudnienia, a z drugiej strony potrzebują bardzo wiele czasu, by dojść do siebie - ze stanem zdrowia, z depresją. W związku z tym chcę zadać takie pytanie, chociaż wydaje mi się, że ono jest retoryczne, bo te rozwiązania (Dzwonek) wynikają z faktu, że w systemie nie ma pieniędzy i być może prędzej czy później zaczniemy również rozmawiać o wieku emerytalnym. Dlaczego chcecie państwo ograniczyć możliwość przeliczenia emerytury dla osób z tzw. starego systemu emerytalnego sprzed 1999 r., dla osób, które nadal pracują?

Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Jakim uszczelnieniem systemu jest planowana zmiana Rady Nadzorczej ZUS?

Sobie również zmniejszacie, tylko tutaj o 50%, a tutaj o 25%.

Wydaje mi się, że (Dzwonek) ta zmiana to kara dla przedsiębiorców za to, że mieli odwagę protestować i głośno wskazywać wasze niekompetencje i złe decyzje, brak realnej pomocy dla nich. Niestety, ale z e-maili prawdy również dowiadujemy się, że centra handlowe i galerie były zamknięte właśnie w wyniku protestów przedsiębiorców, a nie w wyniku sytuacji epidemiologicznej i COVID-owej w kraju.

Zacznijcie kochać Polskę i Polaków i przestańcie ich traktować w sposób feudalny. I bardzo proszę o dyscyplinę, bo nie chcę nikomu przerywać. Bardzo proszę, pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na trzy kwestie, które według mnie są bardzo niepokojące w tej ustawie. Chodzi przede wszystkim o zmiany dotyczące dorabiających emerytów i rencistów, zmiany, które nie premiują aktywności zawodowej, do której powinniśmy zachęcać osoby starsze. Druga kwestia to emerytury czerwcowe.

Chcę się dzisiaj o te osoby upomnieć, ponieważ te przepisy, które proponujecie. Niezauważanie tej grupy osób przypomina mi tak naprawdę tę sprawę, której nie potrafiliście załatwić przez długi okres, czyli sprawę kobiet z rocznika 1953. Proszę kończyć, panie pośle. I trzecia sprawa, która bulwersuje, to rada nadzorcza ZUS, która będzie powołana na nowo w 2022 r.

Bardzo proszę, pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze!

Ustawa ta jest z października 1998 r., była wielokrotnie nowelizowana i teraz jest kolejna, duża nowelizacja. Myślenie, jeśli chodzi o system ubezpieczeń społecznych, też od tego roku wielokrotnie się zmieniało.

Czy nie należy stworzyć nowego aktu prawnego, który ureguluje ten dzisiejszy system ubezpieczeń społecznych na nowo, w pełni?

Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. To pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam dwa pytania. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że przepis ten miał charakter przejściowy i osoby, które chciały z niego skorzystać, już to zrobiły. Czy mają państwo jakieś dane, z których to wynika? Skąd państwo wiedzą, że wszyscy, którzy chcieli skorzystać z tego przepisu, rzeczywiście to zrobili? To jest bardzo ciekawe. I druga sprawa dotycząca zmian w prawie do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Piszą państwo w uzasadnieniu projektu, że taka regulacja ograniczy ewentualne nadużycia. Mam pytanie: Dlaczego traktują państwo wszystkich obywateli, obywateli, którzy chorują, którzy chorują przewlekle, jak potencjalnych oszustów? To po stronie państwa leży kontrola prawidłowości i przestrzegania prawa. Zresztą obserwujemy to również na rynku pracy: pomimo kolejnych apeli Lewicy nie decydują się państwo na wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie. Tutaj rzecz należy do ZUS-u. Dlaczego traktują państwo obywateli jak oszustów? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście przedmiotowy projekt ustawy zawiera takie rozwiązania, które trudno uznać za sprzyjające ludziom aktywnym, ludziom przedsiębiorczym. To jest zastanawiające, bo powstaje takie wrażenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niezbyt sprzyja tym ludziom, którzy chcą pracować, panie ministrze. Warto się jeszcze nad tym zastanowić. Natomiast mam też pytanie dotyczące trochę innego projektu, ale ważnego dla przyszłych emerytów. Chodzi o projekt, który przewiduje defraudację 15% środków, które Polacy zgromadzili na otwartych funduszach emerytalnych. Przypomnę, że cały czas ten projekt leży w parlamencie.

Teraz państwo de facto wprowadzają rozwiązanie, które spowoduje, że emerytury będą zwolnione z opodatkowania. Panie Ministrze! Mam jedno pytanie: Czy i kiedy rząd wycofa się z tego projektu, który ma za zadanie zdefraudować środki zgromadzone przez Polaków w OFE, i kiedy wprowadzicie przepisy, które zlikwidują tę szkodliwą prowizję z tytułu przekształcenia OFE w nowe OFE? Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę o założenie maseczki. Dziękuję. Bardzo proszę. Z całą pewnością te rozwiązania nie są korzystne dla pracowników i z całą pewnością nie jest to właściwy czas na ich wprowadzanie, ale uchwalanie ustaw to jest jedno, a praktyka to drugie. Chciałbym zapytać pana ministra: Czy pan minister dysponuje takimi danymi, a jeśli pan minister nie dysponuje takimi danymi, to prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w ilu przypadkach w 2020 r. decyzjami ZUS-owskimi odmówiono przyznania prawa do emerytury i ile z tych odmów było skutecznie zaskarżonych do sądu? Pytam dlatego, że bardzo często zwracają się do mnie, do mojego biura mieszkańcy, którym ZUS odmówił prawa do emerytury, a następnie na drodze postępowania sądowego tę emeryturę przyznano. Bardzo często powstaje takie wrażenie, że ZUS przez tę praktykę próbuje ograniczyć wypłatę emerytur. Pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Powiem wprost: PiS chce obciąć zasiłki chorobowe o połowę. Ten szkodliwy PiS-owski projekt po 31 latach ogranicza zasiłek chorobowy ze 182 dni do 91. Nadal jesteśmy w trakcie ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. Wiele osób, które przechorowały COVID-19, walczy o powrót do zdrowia, mierząc się ze skutkami i powikłaniami ten poważnej choroby. Jedną z chorób, na którą cierpią ludzie po pandemii, jest także depresja, z której nie da się wyleczyć w ciągu 91 dni. Wiele osób, również przewlekle chorych, w trakcie szczytu pandemii było kompletnie odciętych od możliwości leczenia w normalnym trybie. Oni też potrzebują czasu, aby wrócić do zdrowia. Dlatego mam pytanie: Panie ministrze, dlaczego rząd PiS tak okrutnie traktuje obywateli? Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak to jest, że zawsze robicie tak, że jedną ręką dajecie, a drugą ręką zabieracie? Z jednej strony dajecie możliwość przeliczenia czy też ustalenia wysokości emerytury na podstawie miesiąca korzystniejszego, maja, ale z drugiej strony zabieracie możliwość waloryzacji tej emerytury czy też zwiększenia wskaźnika raz na 3 miesiące w sytuacji, kiedy ktoś pobiera emeryturę i pracuje, zabieracie możliwość właśnie tego kwartalnego przeliczenia, dajecie tylko taką jednorazową możliwość. Ale to, co jest najbardziej skandaliczne, to to, że rzeczywiście skracacie okres zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudniania ze 182 dni do 91. Przecież już od 1990 r. była taka możliwość, kiedy było bezrobocie strukturalne (Dzwonek), kiedy były kryzysy gospodarcze, ale żaden rząd do tej pory nie podniósł ręki na to, aby zmniejszyć ten zasiłek, i to o połowę, a wy to robicie. Pytanie jest jedno: Panie ministrze, ile na tym zaoszczędzicie? Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Skrócenie zasiłku chorobowego ze 181 dni do 91 to jest po pierwsze. Ale po drugie, szanowni państwo, wszyscy wiemy, jak dzisiaj działa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Działa źle. Jest mnóstwo skarg, jest mnóstwo spraw sądowych, które są spowodowane złym orzecznictwem w ZUS-ach. Stanie się tak, ponieważ ktoś, kto jest przewlekle chory i nie ma prawa do świadczenia chorobowego, oczywiście skieruje sprawę do sądu.

Ostatnie pytanie zadaje pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Wysoka Izbo! To, że ta ustawa oczywiście jest jakimś kolejnym skokiem na kasę ludzi prowadzących działalności, ale też ubezpieczonych w przyszłości i ubezpieczonych obecnie, i emerytów, to już sobie ustaliliśmy, to już wybrzmiało tutaj w wystąpieniach wszystkich moich poprzedników, a i ja też o tym mówiłem w swoim wystąpieniu. Ale w związku z tym, że to już sobie ustaliliśmy i że to dosyć jasno wybrzmiewa z tej ustawy, z zapisów mówiących o dodatkowym opodatkowaniu, o skróceniu okresu ubezpieczenia itd., mam jedno bardzo konkretne pytanie: Jaki jest w tym momencie stan ZUS-u, jaka jest kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jakie są braki, jak wielka jest kwota, którą w tym momencie państwo musi gdzieś uciułać, żeby załatać dziurę, która jest od państwa wymagana, którą państwo musi wpłacić, ponieważ się zobowiązało? Dziękuję bardzo. Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana ministra Stanisława Szweda. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję za dyskusję dotyczącą zmiany ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która popularnie zwana jest ustawą o racjonalizacji, gdyż taki jest cel tej ustawy.

Głównym celem jest to, abyśmy ten system spróbowali uporządkować.

Nie ma w ustawie zmian, jeśli chodzi o wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych.

To są dane, które wskazują, że musimy w tym systemie dokonywać zmian.

Jeśli chodzi o kwestię spółek komandytowych, to tutaj nie dokonujemy zmian. Te zmiany są podyktowane też orzecznictwem Sądu Najwyższego i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w swoim orzecznictwie mówi, że musimy doprecyzować przepisy, żeby były jasne przy rozstrzyganiu różnego rodzaju sporów. Takie rozwiązania tutaj w tym zakresie są.

Sytuacja z przechodzeniem na emeryturę jest taka, że jeżeli ktoś spełnia dzisiaj w Polsce warunki, czyli gdy kobieta ma skończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat, to w obecnym systemie emerytalno-rentowym jest tak, że nie ma możliwości odmówienia przydzielenia emerytury i renty.

Jeśli chodzi o kwestie związane z radą nadzorczą, to tu nie ma żadnego zamachu na stronę pracodawców.

Taki był układ rady nadzorczej. Ale przez te lata w Polsce powstały już cztery dodatkowo spełniające warunki reprezentatywne organizacje pracodawców, stąd również zgodnie z ustawą organizacje pracodawcy mają swojego przedstawiciela, organizacje związkowe są na tym samym poziomie, czyli organizacje związkowe są reprezentatywne.

Nie zabieramy, tylko racjonalizujemy ten system.

Corocznie przy okazji omawiania budżetu państwa te dane są podawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

To tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę dyskusję i proszę o uchwalenie ustawy.

Bardzo proszę, pani poseł. Chciałam bardzo podziękować, szczególnie panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi i zespołowi, za pracę nad tą ustawą.

Wiele przepisów wynika, tak jak już powiedział pan minister, z orzecznictwa Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym bardzo proszę, żeby państwo - zwracam się tutaj do posłów opozycji - w swoim zacietrzewieniu nie uprawiali demagogii, tylko naprawdę czytali ze zrozumieniem to, co jest w ustawie, jakie zmiany są wprowadzane.

Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie ministrze, i proszę o uchwalenie przedmiotowej ustawy. Bardzo dziękuję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1018 i 1248) Proszę panią poseł Annę Dąbrowską-Banaszek o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 1018.

Projekt dotyczy przedłużenia kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. wnosi o przyjęcie ww. projektu. Bardzo dziękuję, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Pierwsza głos zabierze pani poseł Danuta Nowicka, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 1018. Przedstawiony projekt przewiduje przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy, jeżeli kadencja tych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. O kwestii przedłużenia kadencji organów statutowych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców dyskutowano z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców oraz reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych. Akceptację na wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych wyraziły m.in.: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Pracodawców Business Centre Club, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” Przedłożony projekt został pozytywnie oceniony przez Radę Ministrów. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. wnosi o uchwalenie go przez Wysoki Sejm. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie omawianego projektu ustawy. Bardzo proszę, pani poseł Ewa Kołodziej, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druki nr 1018 oraz 1248. Ze względu na stan epidemii utrzymujący się ponad rok organy statutowe wielu organizacji, tj. związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, ale również jeśli chodzi o społecznych inspektorów pracy, nie mogły przeprowadzić planowo wyborów statutowych nowych organów w swoich organizacjach. Sytuacja ta wymaga zatem uregulowania prawnego, stąd omawiany projekt przewiduje przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy. Przedłużenie kadencji trwać będzie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po jego odwołaniu do momentu wyboru organu statutowego, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia. W procedowanym projekcie ustawy nie został uwzględniony organ samorządu zawodowego, a zatem proponujemy rozszerzenie brzmienia art. 14i poprzez dodanie po słowach „społecznego inspektora pracy” słów „lub organu samorządu zawodowego” Jest to kolejna grupa przedstawicieli konkretnego środowiska, która ze względu na pandemię nie jest w stanie przeprowadzić planowo wyborów nowych organów statutowych zgodnie ze swoimi statutami. W związku z powyższym składam dzisiaj stosowną poprawkę i w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska po moim wystąpieniu pozwolę sobie przekazać pani marszałek stosowną poprawkę.

Prezentowane rozwiązania legislacyjne uzyskały pozytywną opinię rządu oraz następujących organizacji: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, głównego inspektora pracy, NSZZ „Solidarność”, jak również Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Pracodawców Business Centre Club, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Dodam, że rozwiązanie, którego do tej pory brakowało, jest w obecnej sytuacji konieczne i bardzo wyczekiwane przez zainteresowane strony. Z danych GUS wynika, że w Polsce działa 12,5 tys. związków zawodowych i ok. 400 organizacji pracodawców. Jak słusznie zauważają wnioskodawcy, ich statuty w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości przeprowadzania wyborów czy podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pragnę przy tej okazji przypomnieć, iż uniknęlibyśmy nie tylko dzisiejszej debaty, ale z pewnością moglibyśmy zapobiec chaosowi w wielu organizacjach, których istnienie jest tak ważne dla dialogu społecznego w Polsce, gdyby większość sejmowa rozpatrzyła jeszcze w ubiegłym roku jedną z naszych, Koalicji Obywatelskiej, poprawek zgłaszanych do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Myśmy taką sytuację, szanowni państwo, przewidzieli i już wcześniej, już w zeszłym roku takie propozycje składaliśmy. Jednak ta propozycja nie znalazła uznania większości parlamentarnej. Reasumując, przedstawiając niniejsze stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, chciałabym wyrazić pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu ustawy.

Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska.

Wysoka Izbo! Projekt ustawy, który stworzył klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów jest oczywistą odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych organizacji i związków zawodowych, które w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i następujących w tym czasie obostrzeń nie mogą wybrać swoich ciał statutowych. Dlatego zaproponowaliśmy wydłużenie tych kadencji do czasu odwołania tego stanu i określonego czasu po nim.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w opiniowaniu tego projektu ustawy, na czele z Forum Związku Zawodowych, OPZZ, głównym inspektorem pracy, NSZZ „Solidarność” i wieloma, wieloma innymi organizacjami pracodawców, przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy zainteresowali się tą kwestią. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować także państwu legislatorom sejmowym, którzy wspierali nas we właściwym procedowaniu nad tą ustawą i w stworzeniu poprawek, które wynikają z konsultacji. Dziękuję stronie rządowej za przychylenie się i współpracę.

Druga, która wynika z zainteresowania innych podmiotów - tutaj uzupełniamy - związków pracodawców, ich federacji i konfederacji, oraz zmieniamy jedno słowo, przy stanie epidemii zamieniamy „lub” na „albo” Chciałbym powiedzieć, że w trakcie procedowania nad tą ustawą oczywiście odzywały się inne organizacje, które dowiedziały się o tym procedowaniu. Wiem, że jeden z klubów parlamentarnych także zgłasza stosowną poprawkę. Jeżeli będzie taka możliwość, na pewno się przychylimy do jej poparcia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych po przedstawieniu sprawozdania komisji odnośnie do tego projektu. Wysoka Izbo! Sam projekt dotyczy przedłużenia kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oczywiście jest to pomysł, projekt, który nawiązuje do praktyki legislacyjnej utrwalonej w czasie stanu epidemii, z czym mieliśmy do czynienia w okresie ostatniego półtora roku. Można się zastanawiać, na ile jest to aktualny problem, jednak pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zarówno sytuacja w zakresie szczepień, jak i, powiedziałbym, pewnego ogłoszenia sukcesu w walce z epidemią może spowodować, że np. w okresie jesieni będziemy mieli do czynienia z niejako nawrotem sytuacji, która będzie uniemożliwiała normalne funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji, w tym organizacji związkowych, tych, o których mowa w tym projekcie. W związku z tym, że jest to możliwe, sam pomysł oceniamy pozytywnie. Jako Koło Parlamentarne Polska 2050 będziemy ten pomysł wspierać i sam projekt popierać. Myślę, że na uwagę zasługuje fakt, iż jest to w pewien sposób projekt wyjątkowy. Jest to projekt klubu opozycyjnego. W ostatnich latach takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Jeżeli powiem, że jest to jeden pewnie z dwóch, może trzech projektów w ciągu ostatnich 6 lat, które zostały czy są procedowane przez parlament jako projekty autonomiczne i których autorami są posłowie opozycji, to będzie pokazywało, jak wyjątkowa to sytuacja. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, jest to oczywiście projekt idący w dobrym kierunku. W związku z powyższym, tak jak już zaznaczyłem, Polska 2050 będzie ten projekt wspierać na dalszej ścieżce legislacyjnej. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. Panie Pośle, maseczki, maseczki. Nie, panie pośle, nie oszukujmy się. Dajemy Polakom przykład, jak się zachowujemy na sali. Panie pośle, bardzo proszę. Obowiązuje zarządzenie pani marszałek Sejmu. My dajemy przykład Polakom. Bardzo proszę założyć maseczkę albo wyjść z sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo! Szkoda, że zdecydowano się włączyć go do porządku obrad tak późno. Jest to inicjatywa, która odpowiada na potrzeby związków zawodowych. Podobne rozwiązanie udało się wprowadzić w ustawach COVID-owych w przypadku organizacji społecznych, nie było więc żadnego powodu, żeby pomijać związki zawodowe w tej regulacji. Ona umożliwia rzeczywiście wydłużenie kadencji organów tam, gdzie regulamin nie przewiduje możliwości zdalnego obradowania i zdalnego podejmowania decyzji.

Nie mamy żadnej pewności, że będziemy na pewno, w 100% bezpieczni, co udowadniał przed chwilą swoją postawą jeden z kolegów posłów. A więc zdecydowanie będziemy za tą ustawą, będziemy ją wspierać. Mamy nadzieję, że pojawią się dyskutowane na posiedzeniu komisji w tej sprawie konieczne poprawki, bo pewne poprawki są potrzebne. Mam nadzieję również, że uda się ją jak najszybciej wprowadzić w życie, żeby ułatwić organizacjom społecznym i zawodowym funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów posłów chce się jeszcze zgłosić do zadania pytania? Jeżeli nikt, zamykam.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Niezliczona była liczba przypadków, kiedy nowelizowane były specustawy COVID-owe. Dziś kolejny taki przypadek w sprawie szczegółowej, natomiast ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat spraw ogólnych. Przez Polskę w tej chwili przelewa się fala bezprawia, bezprawia związanego z nadużyciami prawnymi dokonywanymi pod pretekstem specjalnych regulacji prawnych czy sanitarnych dokonywanych w związku z chorobą COVID-19. Konfederacja w ostatnich dniach przedstawiła remedium na te nadużycia. To ustawa: stop segregacji sanitarnej. Zapraszam wszystkich posłów do podpisywania tego projektu. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście za tym, żeby bezpodstawnie łamać prawo obywatelskie, żeby popierać segregację sanitarną, to powinien się z imienia i nazwiska w tej Izbie ujawnić, pokazać wyborcom i powiedzieć: to ja chcę łamać wasze prawa obywatelskie, Polacy, to ja stoję za tym, żeby rząd mógł naruszać prawa tych, którzy pracują dla naszego państwa - żołnierzy, funkcjonariuszy służb, grozić wstrzymywaniem awansów, grozić usunięciem ze służby tylko za to, że np. ktoś korzysta z praw, które nawet rząd teoretycznie popiera, czyli z dobrowolności przyjęcia lub nieprzyjęcia szczepienia na COVID-19. Długo by można było mówić o absurdach związanych z niszczeniem działalności gospodarczej w Polsce. W tej chwili, mimo rekordowo niskiej liczby zachorowań, ciągle utrzymywany jest kuriozalny stan epidemii. Drogi rządzie, uchylcie ten stan epidemii. Drogi rządzie, pójdźcie po rozum do głowy i zacznijcie stosować jednakowe zasady dla wszystkich. Dlaczego w tej chwili rzekomo obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, a przez Warszawę właśnie przeszła wielka parada równości? Okazuje się, że jak ktoś wywiesi tęczową flagę, to dla tego rządu, rzekomo prawicowego, jak tutaj mówiła pani Biejat, że to rząd Prawicy, podobno nawet Zjednoczonej, mimo że wzajemnie próbują się zniszczyć w tej chwili z Gowinem i Bielanem, manifestacje pod tęczową flagą są nietykalne. Stan epidemii? A gdzie tam. A niech idzie i 15 tys., byle pod tęczową flagą, bo mają ochronę ambasady amerykańskiej, bo wywiesili tęczową flagę. To jest dla was punkt odniesienia.

Byli partyjni, którzy mieli co innego do powiedzenia na okoliczności publiczne i co innego na okoliczności prywatne. Dzisiaj mamy partyjnych z rządu, partyjnych z opozycji. Podwójna moralność w każdej kwestii. Uchylmy stan epidemii, skończmy z tym absurdem. Zamiast specustawami COVID-owymi wydłużać w tej chwili kadencje w różnych organizacjach, zajmijmy się rzeczywistym bezprawiem. Parki rozrywki na świeżym powietrzu maksymalnie do 50% obłożenia. Dlaczego? Ile jeszcze miesięcy będziemy niszczyć ludzi, którzy zainwestowali prywatny majątek, żeby innym sprawić trochę radości? Następna sprawa. Obiekty sportowe, nawet te na świeżym powietrzu, do 50%. Co to za bzdury? W Sejmie 100%, a na świeżym powietrzu 50%? Na poprzednim posiedzeniu w tych ławach opozycyjnych widziałem byłego szefa Platformy bez maseczki, jednego z liderów Lewicy bez maseczki, a do mediów ganiacie w maseczkach. Kim jesteście? Opozycją? Czy wspieracie rząd w bezprawiu? Następna sprawa. W części pozostałych obostrzeń już występuje segregacja sanitarna. W kościołach rzekomo ma być 75% osób, ale nie dotyczy to osób w pełni zaszczepionych. Policjantów postawicie przy wejściu do kościoła, żeby sprawdzali, czy ludzie są zaszczepieni czy nie? Będą musieli sobie na czoło przykleić te certyfikaty szczepienne? Następna sprawa. Zadzwonił do mnie obywatel w ostatnich dniach, że był szczepiony w Stanach Zjednoczonych, gdzie przechorował COVID. I okazuje się, że on się do waszego systemu nie jest w stanie zapisać. Nieprzewidziany przypadek. Nic z tego nie wynika. Stworzyliście system iście kafkowskiego absurdu, w który wprzęgnięci są obywatele. Dopóki dziennikarze będą to wszystko traktować poważnie, wy będziecie to traktować poważnie. Retorycznie jesteście przeciwko rządowi, walicie w pulpity, jak coś przez przypadek uda wam się przegłosować, a nie potraficie postawić się w sprawach elementarnych. Stop segregacji sanitarnej - nasz projekt ustawy. Zapraszam, panie pośle, do podpisywania. Pokażcie czynami, a nie słowami. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pytań. Pierwsze pytanie zadaje pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Panie Pośle Bosak! I bardzo dobrze, bo Polska musi być otwarta, tolerancyjna i włączająca, a nie wykluczająca. Szanowni państwo, poza tym, że wspieramy ten postulat, który się pojawił, dotyczący przedłużenia kadencji, to zwracamy również uwagę na patologię tej ustawy. I to będzie konkretne pytanie do panów ministrów. To jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówi o tym, że w Ministerstwie Zdrowia, wykorzystując ustawę COVID-ową, omijaliście Prawo o zamówieniach publicznych. Jaki to ma związek z przeciwdziałaniem COVID-owi? Kiedy zostanie zmieniony - to jest konkretne pytanie - art. 6a ustawy COVID-owej, zgodnie z którym do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-owi nie stosuje się prawa zamówień publicznych? Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Dlatego z całą pewnością poprzemy to, aby przedłużać kadencje podmiotów społecznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, szeregu instytucji, które zgłaszają się do nas i proszą również o to, aby przesunąć wszystkie wymagania statutowe, wymagania przewidziane prawem. To jest oczywistość, żeby w pandemii dać na to szansę, i będziemy popierać projekt ustawy zgłoszony przez kolegów z Koalicji Polskiej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo proszę, pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Kolejna nowelizacja ustawy COVID-owej - potrzebna, wskazana i oczekiwana. Niestety, ustawa nie zawiera i nie obejmuje wszystkich organizacji, jeśli chodzi o możliwość przedłużenia kadencji. Nie obejmuje bowiem związków zawodowych organizacji przedsiębiorców, a także nie ma słowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ale nim przejdziecie państwo do kolejnej nowelizacji, która będzie dotyczyła ustawy COVID-owej, moje pytanie brzmi: Co z projektem ustawy COVID-owej dotyczącym przedsiębiorców, art. 15ze, czyli najemców w galeriach handlowych, i czterech lockdownów, które ich wykańczają i narzucają zobowiązania finansowe, przez co tracone są miejsca pracy i zamykane firmy? Projekt trafił do komisji i leży w zamrażarce. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Pomijam już fakt - bo tutaj akurat jest jeden z nielicznych przykładów, gdzie mogę zgodzić się z panem posłem Bosakiem - że w moim przekonaniu wprowadzenie tego stanu i na jego podstawie ograniczenie chociażby wolności działalności gospodarczej czy wolności zgromadzeń jest absolutnie niezgodne z konstytucją i prawdopodobnie w najbliższym czasie, w najbliższych latach będziemy mieli mnóstwo pozwów sądowych, myślę, że wygranych w tym zakresie.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Moje pytania będą szły w tym samym kierunku, bowiem pandemia jest czasem przejściowym i taki charakter powinna mieć ta ustawa. To powinna być ustawa o charakterze przejściowym, a nie stałym. Pierwsze pytanie powtórzę za panem posłem: Kiedy nastąpi usunięcie tego stanu? Przecież wszystkie wskaźniki są pozytywne, pan minister mówi, że jesteśmy na dobrej drodze, ale może być kolejna fala czy jeszcze kolejna. Tymczasem w tej ustawie jest tylko mowa o tym, że do 90 dni po usunięciu, po likwidacji, po ogłoszeniu, iż zakończony jest stan pandemiczny. Ale kiedy? Bo w przeciwnym wypadku powstaje jednak takie poczucie i niebezpieczeństwo, że te kadencje będą przedłużane właściwie nie wiadomo jak długo. Czerwiec to czas, kiedy w spółdzielniach mieszkaniowych są walne zgromadzenia.

Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Pierwotnie ten projekt ustawy obejmował tylko związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców i społecznego inspektora pracy. W trakcie oficjalnych konsultacji i zgłaszania opinii doszły uwagi przedsiębiorców, ich federacji i konfederacji, i postanowiliśmy jako klub taką poprawkę zgłosić poprzez uzgodnienia z rządem i z legislatorami.

Druga sprawa. Obiecałem, że nie będę narzekał w oficjalnej wypowiedzi, ale też uważam, że można było to zrobić szybciej. Mam nadzieję, że za chwilę nie będziemy mieć stanu zagrożenia epidemicznego. Rzeczywiście, jak przejrzymy pisma naukowe, [[Dzwonek]] najbardziej prestiżowe typu brytyjski „Lancet”, to tam jest napisane, że jeżeli mamy podwójne szczepienie, nie ma szans się zakazić, więc mam nadzieję i apeluję do Prezydium Sejmu, żebyśmy tutaj, w ramach wykonywania obowiązków - jesteśmy w pracy - ci, którzy się zaszczepią, nie musieli nosić maseczek, bo jak idziemy do telewizji czy gdziekolwiek indziej, to tam nikt od nas nie wymaga maseczek, a jesteśmy w identycznym gronie jak tutaj. Szanowny panie pośle, nie ma nigdzie stwierdzenia, że nawet po dwóch szczepieniach nie można zachorować na tę chorobę. Można, tylko lżej się ją przechodzi. To nie jest tak, że jak jesteśmy zaszczepieni, to już nigdy nie zachorujemy. Możemy zachorować, tylko przechodzimy tę chorobę lekko i nie musimy iść do szpitala. Nawet w naszym Sejmie są osoby, które były dwukrotnie szczepione i przechodziły tę chorobę. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Mówimy o związkach zawodowych i innych rzeczach, a czy myślimy o stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach, partiach politycznych, walnych zgromadzeniach w spółkach? Dlaczego tak wybiórczo?

Czy to w jakichś innych przepisach jest uregulowane? Ostatnie pytanie zadaje pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Z ustawy COVID-owej w dalszym ciągu wynika obowiązek instalowania specjalnej aplikacji przez osoby, które zostaną skierowane na kwarantannę. Nie jest tajemnicą, że ta aplikacja gromadzi dane o użytkowniku, w tym dane lokalizacyjne.

Ich oświadczenie jest składane pod odpowiedzialnością karną, państwo grożą odpowiedzialnością karną za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

Jak długo te dane są przechowywane? Kiedy zostaną zniszczone? Po co wam te dane? Dziękuję bardzo. Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pana Marka Niedużaka o udzielenie odpowiedzi. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Tak na moje oko mamy tutaj w dużej mierze pytania z właściwości ministra zdrowia, ale również ministra sprawiedliwości, chyba ministra cyfryzacji i być może całej Rady Ministrów, szczególnie jeśli chodzi o pytania dotyczące stanu epidemii.

Właśnie niektórym pytającym chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest przedłożenie rządowe.

Chociaż, tak jak mówię, tutaj jednomyślności po stronie pracodawców akurat nie było.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druki nr 1236 i 1304) Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedłożenia sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z druku nr 1304 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe z druku nr 1236.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i wielki honor przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość co do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. To sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych zostało zawarte w druku sejmowym nr 1304. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera te rozwiązania, popiera te bardzo dobre pomysły, które zostały przedstawione przez przedsiębiorców, przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i poparte właśnie przez Ministerstwo Finansów oraz zaproponowane w tym projekcie ustawy.

Podczas prac w komisji miałem zaszczyt zgłosić dwie poprawki, które uzyskały akceptację wysokiej komisji i znajdują się w tym przedłożeniu.

Te uwagi, te propozycje zostały przyjęte przez wysoką komisję, jak wspomniałem.

Tak jak wspomniałem, ten projekt ustawy był szczegółowo omawiany podczas pierwszego czytania.

Przede wszystkim zwracam jednak uwagę na to, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę do Wysokiej Izby o to, aby ten projekt ustawy przyjąć. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, pani marszałek.

Mamy wrażenie, że trochę na kolanie to jest pisane, więc nie zgadzam się tu z przedmówcą, że to super było przygotowane. Jeżeli przedsiębiorcy oczekują, że przepisy prawa będą proste i stabilne, a główną wadą jest komplikacja właśnie tych przepisów i problemy z ich interpretacją, to może trzeba sobie dawać więcej czasu na takie przygotowywanie projektów ustaw, żeby chociażby legislatorzy aż tylu błędów nie wytykali. To jest często powtarzane - to, że polski system podatkowy zniechęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, a te przepisy nie są dla ludzi, dla zwykłych ludzi, choć to zwykli ludzie prowadzą przedsiębiorstwa, ale często dla prawników z korporacji, doradców podatkowych bądź samych urzędników, którzy te przepisy interpretują.

Mówię: chcemy wierzyć, bo potem niejednokrotnie życie nas przekonuje, że kłopoty właśnie z interpretacją przepisów, ze zrozumieniem prawa są czasami, mimo dobrych chęci, jeszcze gorsze niż przed jakimikolwiek nowelami. Wpłynęło też stanowisko Związku Banków Polskich. Rząd wczoraj nie umiał się do tego stanowiska odnieść, bo go nie znał. Pytanie: Czy już dzisiaj pan minister to stanowisko poznał? Związek Banków Polskich zwraca uwagę na niedociągnięcia tej ustawy, na coś, co może przeszkadzać, jak chociażby to, że trzeba systemy informatyczne przygotować do tego, żeby rozpoznawały przelewy z KRUS, więc Związek Banków Polskich mówi o przedłużeniu terminu wejścia w życie przepisów tej ustawy z tym związanych. Pyta też o kurs walut, według którego trzeba przeliczać korekty transakcji w przypadku transakcji międzynarodowych, czy też o sposób dostarczania i zakres informacji, jeśli chodzi o powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, które ma być wysyłane odnośnie do byłych klientów banku.

Czy jest to problem, czy tylko „wydumany” problem? Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, jeżeli ktoś zwraca uwagę, to po co się tak spieszymy?

Jeszcze raz: chcemy wierzyć, że to jest dobrze napisane i że przedsiębiorcy z tego naprawdę skorzystają. Dlatego zamierzamy poprzeć te rozwiązania, zwracając uwagę na ten tryb prowadzenia legislacji, żeby nie spieszyć się, nie pisać na kolanie i na tyle konsultować, reagować, badać, żeby wygładzać te przepisy, żeby one były przyjazne przedsiębiorcom, żeby przedsiębiorcy przestali mówić, że w prowadzeniu działalności gospodarczej przeszkadzają im przepisy obowiązujące w Polsce. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Trela, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko w imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Tak jak mówiłem podczas pierwszego czytania, każdy projekt ustawy, który ulepsza, poprawia czy ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorców, jest godny poparcia. Lewica go poprze. Poprze oczywiście te poprawki, które były wczoraj zgłaszane na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. On może fundamentalnych wątpliwości nie budzi, natomiast pytań na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych było bardzo wiele, przedstawiciela Ministerstwa Finansów czy ministra finansów nie było, na te pytania nie miał kto odpowiedzieć. Na to też nie było żadnej odpowiedzi. A więc z tym pośpiechem co do oceny jakości przedkładanych projektów ustaw pozwoliłbym sobie się nie zgodzić. Również niespecjalnie zgadzam się z nadmiernym pośpiechem, dlatego że nawet ustawy techniczne, które doprecyzowują pewne rzeczy czy wskazują bardziej szczegółowy ich zakres, powinny być opracowywane i powinny być dyskutowane zdecydowanie dłużej, nawet jeżeli nie budzą wątpliwości sprawy ich fundamentu. Natomiast co do zakresu przedmiotu i kierunku działań w takich sprawach należy to poprzeć. Oczywiście bezsporną kwestią jest to, że projekt ustawy też dostosowuje pewne rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie Unii Europejskiej, sprawy wspólnotowe, chociażby te, które dotyczą wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. Jeszcze raz w imieniu koalicyjnego klubu parlamentarnego deklaruję poparcie dla tego projektu ustawy wraz ze złożonymi poprawkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe po przedstawieniu sprawozdania komisji. Szanowni Państwo! Jak już tu wielokrotnie zostało zauważone, w przedstawionym projekcie rząd wskazał, iż celem tych rozwiązań są zmiany w rozliczaniu przez podatników podatku od towarów i usług. Przedstawione Wysokiej Izbie rozwiązania nazwano pakietem Slim VAT 2 i rzeczywiście wypada się zgodzić, że zawartość tego pakietu jest w wersji slim. Oczekiwalibyśmy od rządu zdecydowanie bardziej odważnych działań, jeżeli chodzi o upraszczanie, o likwidowanie zbędnej biurokracji, o wdrażanie takich mechanizmów, które sprzyjają prowadzeniu działalności. Bo dzisiaj wydaje się, że jednym z najważniejszych problemów, ale też i wyzwań po stronie przedsiębiorców, po stronie pracowników jest uczynienie zadość tym wszystkim obowiązkom biurokratycznym, które są codziennie nakładane przez rząd i kolejne urzędy, urzędy skarbowe i inne urzędy, które wymyślają coraz to nowe ścieżki biurokratyczne, które muszą zostać pokonane, żeby osiągnąć jakiś efekt dotyczący relacji z urzędem. W związku z tym, panie ministrze, oczywiście to dobrze, że powstają takie rozwiązania sprzyjające przedsiębiorcom. Niestety w parlamentarnej zamrażarce, w komisjach parlamentarnych jest bardzo wiele projektów autorstwa również rządu Prawa i Sprawiedliwości, które komplikują tę gospodarczą rzeczywistość. I mam taki apel do pana ministra, aby jednak spróbować te działania w jakiś sposób omówić w ramach prac rządu, tak aby charakter tych zmian był zawsze jednoznacznie upraszczający, jednoznacznie ułatwiający działanie polskim firmom, polskim przedsiębiorcom, pracownikom. Z jednej strony dzisiaj widzimy, że jest projekt, który niejako idzie w tym kierunku, ale tak jak powiedziałem, jest wiele innych projektów, które wprost przeciwnie, te warunki prowadzenia działalności komplikują, a tak być nie powinno, i tamte projekty oceniamy pod tym względem jako negatywne. Zresztą nawet dzisiaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w projekcie ustawy, który dotyczył systemu ubezpieczeń społecznych, postulowane tam przez rząd zmiany nasuwały refleksję, że rząd nie lubi ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy ciężko pracują, którzy wykonują swoją pracę codziennie z myślą o swoich rodzinach, o swojej przyszłości, więc warto by było, aby zdecydował, czy jest za przedsiębiorczością, za ludźmi pracy, za tymi, którzy codziennie ciężko pracują, czy wprost przeciwnie - woli urzędników, którzy komplikują życie tym ciężko pracującym ludziom. Natomiast sam projekt, tak jak zostało już wspomniane, rodzi pewne wątpliwości, które najszerzej zostały wyartykułowane w stanowisku Związku Banków Polskich. Dotyczą one m.in. kwestii dostosowania systemów teleinformatycznych do wymagań przepisów zaproponowanych w tym projekcie. I, panie ministrze, wczoraj te wątpliwości, które podniósł Związek Banków Polskich, nie zostały rozwiane i to jest bardzo poważny element, który oczekujemy, że pan minister tutaj wyjaśni. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówią banki, że w tym terminie, który jest zapisany w ustawie, te systemy informatyczne nie będą dostosowane do tych wymagań. Bo jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to - szczerze mówiąc - te zmiany na nic, ponieważ, jak słusznie wskazuje Związek Banków Polskich, żeby można było w sposób jasny, oczywisty i czytelny je wprowadzić i aby one mogły działać, musi zostać wykonana jakaś praca. Nie wiadomo, czy jest to możliwe. Drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że Polska 2050 składa poprawkę do tej ustawy. Jej ratio legis jest ułatwienie dokonania pewnych operacji związanych z uwalnianiem środków właśnie na rzecz przedsiębiorców.

Bardzo proszę, pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja.

Otóż zwracam uwagę, że w Polsce już od dłuższego czasu Polacy siedzą legalnie w restauracjach bez maseczek. Tutaj jesteśmy w wielkiej, klimatyzowanej sali plenarnej, w której obecnie znajduje się może kilkanaście osób, ale mimo to pani marszałek mnie wyprosiła, kiedy pojawiłem się tu bez maseczki, i zastanawiam się, czy to jest zwykła hipokryzja, bo poza kamerami już wszyscy nieco inaczej się zachowują, czy to jest po prostu stawianie bezpieczeństwa posłów wyżej niż bezpieczeństwa zwykłych Polaków. Natomiast co do VAT-u i podatków VAT. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć o rzeczy podstawowej do zwykłych ludzi, którzy nie siedzą w szczegółach legislacji, żebyśmy dobrze zrozumieli, co to jest podatek VAT. To nie jest jakiś specjalistyczny podatek nakładany na przedsiębiorców. To jest zwykły, powszechny haracz nakładany na wszystkich, bo na konsumentów.

Przedsiębiorcy, usługodawcy, handlarze są tylko przymusowo poborcami tego podatku VAT, a wy za każdym razem ten VAT płacicie. U nas stara się to ukryć, tak że, szanowni państwo, pamiętajcie: jak dostajecie 500+ i się z tego cieszycie, to nie zapominajcie, że przy każdych zakupach oddajecie te 500+ z nawiązką. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Lista zmian wprowadzanych w nowelizacji podatku VAT, którą przedkłada rząd, przyprawia o zawrót głowy i uświadamia, jak skomplikowany jest system podatkowy. Odczytam tylko dziewięć z tych zmian, które tutaj wynotowałem. Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych, umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku. Trzecie, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie zastosowania. Czwarte, ułatwienie odliczania VAT na samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej, 100% odliczeń od wydatków poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd. Piąte, umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na bieżąco, rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia poprzez korektę deklaracji. Szóste, dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Siódme, uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny. Ósme, umożliwienie wydania zgody na uwalnianie środków z rachunku VAT, jeśli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty. Dziewiąte, umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS. Nic dziwnego, że ludzie potrzebują doradców podatkowych, żeby prawidłowo płacić podatki. Przypomnijmy, że podatek VAT jest harmonizowany na poziomie Unii Europejskiej, w związku z tym te zasady, które tutaj, w Polsce, mamy, również są przedmiotem uzgodnień międzynarodowych, a to oznacza, że nie tylko kadra podatkowa Ministerstwa Finansów, ale również eurokraci czuwają nad tym, byśmy się w tym nie pogubili. Jednak trzy zmiany, które ministerstwo zapowiadało i które wydawały się korzystne dla przedsiębiorców, zniknęły z tego projektu. O ile te wcześniej wymienione zmiany wydają się pozytywne i korzystne dla przedsiębiorców, to korzystając z obecności przedstawiciela Ministerstwa Finansów siedzącego w ławach rządowych, ministra Sarnowskiego, pragnę zwrócić uwagę na te trzy zmiany, które zniknęły. A więc zapowiadana była likwidacja obowiązku odpowiedniego oznaczenia faktur oraz faktur korygujących. Dziennik Gazeta Prawna” informował, że w lutym na konferencji prasowej właśnie pan wiceminister podkreślał, że takie wymogi są wyłącznie w trzech krajach unijnych: Francji, Holandii i Polsce, i że zasadniczo są niepotrzebne. Ostatecznie państwo od tego odstąpiliście. Druga sprawa. Zrezygnowano również z planowanego zniesienia ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Pierwotnie Ministerstwo Finansów zapowiadało, że podatnicy będą mogli je wystawiać nie tylko w odniesieniu do całych faktur, ale także do konkretnych pozycji, co miało przyspieszyć, uelastycznić proces wystawiania zbiorczych korekt. To też zniknęło. Z projektu zniknęła też zmiana mająca na celu wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawianie faktury jeszcze przed transakcją. Obecnie jest 30 dni, miało być 60 dni, to także z projektu wyparowało. Jako Konfederacja zadajemy pytanie: Dlaczego te, wydaje się (Dzwonek), racjonalne pomysły wyparowały z projektu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kto z pań i panów posłów chce zgłosić się do zadania pytania? Mamy posłów do zadania pytania? Bardzo proszę, 1 minuta na zadanie pytania i zamykam listę. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska.

To tylko świadczy o rozchwianiu i skomplikowaniu naszego systemu podatkowego. Kiedyś były 3 miesiące na wydanie indywidualnej interpretacji. Przepisy COVID poszerzyły to, jeżeli dobrze pamiętam, nawet do 9 miesięcy.

Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mówiliśmy o tym podczas pierwszego czytania, ale dzisiaj, podczas drugiego czytania, chciałbym usłyszeć zapewnienie pana ministra i potwierdzenie tego, że tak rzeczywiście było, że te postulaty wynikały i pochodziły od przedsiębiorców, że bardzo dużą aktywność wykazał tutaj rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To jest ustawa, która idzie w dobrym kierunku, ale to za mało, panie ministrze. Dzisiaj mamy w Polsce taką sytuację, że są setki nowelizacji, setki poprawek, mamy coraz grubsze ustawy, a przedsiębiorcy oczekują zupełnie czegoś innego. Przedsiębiorcy oczekują czytelnych i krótkich przepisów prawnych, żeby mogli rozwijać własne biznesy. Ona jest zbyt dowolna, czasami na tę interpretację trzeba czekać bardzo długo i niestety ona czasami jest skierowana przeciwko przedsiębiorcom. Ta pozycja Polski niestety w ostatnich latach spada. Zatem powinniśmy tworzyć warunki, by polscy przedsiębiorcy chcieli inwestować w Polsce. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Minister Kościński, zapowiadając pakiet Slim VAT 2, stwierdził, że rozwiązania zawarte w ustawie przygotowane zostały jako odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rynek.

Kiedy doszliście do władzy, temat szybko zniknął. VAT nie został obniżony nawet w okresie najlepszej koniunktury. Proszę o odpowiedź na pytanie: Dlaczego z noweli zniknęły zapowiadane wcześniej uproszczenia dotyczące fakturowania?

Co jest powodem tego nagłego pośpiechu? Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Ilość zapisów w ustawie o VAT jest oszałamiająca, ale brakuje tych kluczowych.

Tak usprawniacie pracę przedsiębiorcom. Pytam: Dlaczego wycofaliście się z kluczowych zapisów tak istotnych dla przedsiębiorców?

Ostatnie pytanie, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ponieważ wczoraj podczas posiedzenia komisji pan minister był uprzejmy nie zaszczycić swoją obecnością, to chciałem prosić o odpowiedź na dwa bardzo ważne pytania, które pojawiły się w stanowisku Związku Banków Polskich. Pierwsze dotyczy dostosowania systemów teleinformatycznych.

Związek Banków Polskich informuje i alarmuje, że na dzisiaj nie ma wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób ten problem rozwiązać. W związku z tym pytam, co tutaj proponuje ministerstwo. Pytanie - oczywiście w relacjach wewnątrzwspólnotowych - brzmi: Jakie (Dzwonek) należy zastosować kursy walutowe w ramach tych przeliczeń? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Cieszymy się, że możemy wspólnie realizować te projekty i po prostu wdrażać w życie postulaty, które trafiają do nas z rynku. Rzeczywiście jest to projekt, którego założenia były przygotowane wspólnie na linii Ministerstwo Finansów - rzecznik MŚP, natomiast o ile duża część propozycji wpłynęła bezpośrednio od niego, o tyle były one zgłaszane również przez Konfederację Lewiatan i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji. To są podmioty najaktywniejsze w zgłaszaniu nam możliwych kierunków działania, również kierunków w zakresie uproszczeń systemu podatkowego, za co chciałbym także tutaj, na tej sali, przy państwu posłach najserdeczniej podziękować.

Przeprowadziliśmy spotkania i ze Związkiem Banków Polskich, i z poszczególnymi jego członkami.

Specjalnie po to, żeby ułatwić dostosowanie systemów bankowych do nowych rozwiązań, rozłożyliśmy ich wdrażanie w czasie, tak że od 1 października wejdzie w życie możliwość uwalniania środków z rachunków technicznych, a dopiero 1 stycznia z rachunków VAT-owskich na rzecz KRUS-u, na rzecz płatności w tym kierunku.

Treść tego rozporządzenia już jest widoczna na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Odnośnie do elementów dotyczących oznaczania faktur duplikatami, ewentualnie tego, że faktura jest korektą, odnośnie do zbiorczych faktur korygujących oraz wydłużenia terminu na wystawienie faktury, to biorąc pod uwagę fakt, że jest to projekt dotyczący fakturowania, jest on procedowany przez Ministerstwo Finansów wraz z projektem e-faktury. Oznacza to, że trafi w najbliższych tygodniach pod obrady Rady Ministrów, ale to też oznacza, że ścieżka legislacyjna tego projektu według planu Ministerstwa Finansów zostanie zakończona w perspektywie października tego roku, a przepisy wejdą w życie w styczniu, razem z większością rozwiązań zawartych w tej konkretnej ustawie. Tak że tutaj nie ma żadnego zagrożenia dotyczącego przyjęcia tych założeń, zostaną one zrealizowane tak, jak o tym komunikowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku, w całości. Powodem błyskawicznego przyjęcia przez Radę Ministrów omawianego dzisiaj pakietu jest bardzo dobre przyjęcie jego założeń przez rynek w ramach prekonsultacji, które realizowało Ministerstwo Finansów.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

Ta ustawa, tak jak wspomniałam, kompleksowo określa status zwierzęcia na służbie: od momentu doboru np. psa do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych służbach, aż do momentu wycofania go ze służby. Psy wspomagają funkcjonariuszy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i spokoju. Psy używane przez służby ratują życie i zdrowie w ramach akcji poszukiwawczych, pomagają wyszukiwać narkotyki czy innego rodzaju kontrabandę i są nieocenione, jeżeli chodzi o wyszukiwanie ładunków wybuchowych, a także pomagają w działaniach wykrywczych związanych z poszukiwaniem sprawców przestępstw.

Pierwszy pies, jaki w ogóle pełnił służbę, nazywał się Topper. Pierwsza szkoła dla psów policyjnych została otwarta w Bawarii.

Ustawa określa wymogi dla opiekuna, któremu powierza się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach. Określa też bardzo dokładnie obowiązki tego opiekuna, czyli to, w jaki sposób ma o tego psa dbać, zapewnić mu odpowiednią karmę, odpowiednie wyżywienie, odpowiednią kondycję, odpowiednią pielęgnację.

Zwierzęta zostają wycofane ze służby na skutek trwałej utraty sprawności użytkowej, wystąpienia choroby nierokującej poprawy, wystąpienia narowów u konia, braku postępów w szkoleniu.

Nie zawsze jednak taka osoba będzie mogła wziąć zwierzę pod swoją opiekę, dlatego ustawa dokładnie przewiduje, kto w następnej kolejności może zostać jego opiekunem.

Stworzył on takie miejsce, ale nie ukrywajmy, bardzo trudno jest prowadzić tego rodzaju schronisko bez żadnego wsparcia. Po przyjęciu tego projektu ustawy sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej.

W trakcie prac komisji zostały złożone poprawki.

Panie ministrze, oczywiście, to jest żart. W imieniu moich koleżanek i kolegów z komisji proszę Wysoką Izbę o jak najszybsze uchwalenie tej ustawy. Czworonożni funkcjonariusze i ich opiekunowie na to czekają. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

4 maja pani marszałek skierowała go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pierwsze czytanie odbyło się 14 czerwca. Projekt był szczegółowo omawiany w komisji i z pełną aprobatą przyjęty przez wszystkich członków komisji. Ustawa reguluje status zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa oraz zwierząt, które pracują w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i w Służbie Więziennej. Pomimo znacznego postępu, rozwoju nowych technologii, zwierzęta nadal odgrywają i będą odgrywać znaczną rolę, wspierając funkcjonariuszy w wykonywaniu ich ustawowych zadań. To właśnie zwierzęta stanowią realne wsparcie dla funkcjonariuszy, a w niektórych przypadkach są wręcz niezastąpione. Zatem konieczne i społecznie oczekiwane było uregulowanie statusu zwierząt w służbach. W projekcie ustawy wprowadzono możliwość używania psów służbowych lub koni służbowych w celu realizacji określonych zadań ustawowych: ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia działań kontrterrorystycznych, wykrywania przestępstw i wykroczeń, ścigania ich sprawców, realizacji zadań reprezentacyjnych, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach i wreszcie ochrony obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów.

Rocznie ok. 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę. Zaproponowane w ustawie rozwiązania dotyczą zwierząt od momentu ich doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po czas ich wycofania ze służby i pobyt na emeryturze. W projekcie ustawy określone zostały obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt obejmującego: racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody, dbanie o stan zdrowia i kondycję, pielęgnację, utrzymanie zwierząt w czystości i zapewnienie warunków utrzymania dostosowanych do potrzeb biologicznych. Jednocześnie określony został mechanizm przydzielania przez poszczególne formacje zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera projektowaną ustawę, która zawiera dziesięć artykułów.

Poprawka określa status zwierząt używanych w Siłach Zbrojnych. Dotyczy dbania o zdrowie tych zwierząt i szkolenia. Określa się nadzór nad psami, które pracują w Siłach Zbrojnych. Ustawa, o której rozmawiamy, wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawodawca jednak przewidział możliwość realizacji zapisów tej ustawy już wcześniej, a więc zwierzęta wycofywane ze służby będą mogły być objęte szczególną ochroną jeszcze przed jej wejściem w życie. Przyjęcie projektowanych rozwiązań stanowi realizację oczekiwań społecznych (Dzwonek), w tym oczekiwań samych funkcjonariuszy i żołnierzy, a więc proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy ponad podziałami, z pełną aprobatą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zawartego w druku nr 1132. Podstawowym celem projektu jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Służbie Więziennej poprzez zapewnienie dożywotniego utrzymania i opieki weterynaryjnej psom i koniom, które będą pozostawały na stanie danej jednostki także wtedy, gdy przejdą na tzw. emeryturę. To drugie podejście w trwającej kadencji Sejmu do tego zagadnienia. Wówczas tzw. mały projekt został wniesiony w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przez posłankę Katarzynę Piekarską, która została sprawozdawczynią obecnego projektu. W służbach znajduje się ok. 1 tys. psów oraz kilkadziesiąt koni. Rocznie blisko 10% tych zwierząt jest wycofywanych ze służby. Co jakiś czas w mediach pojawiały się informacje o usypianiu psów z powodu braku chętnych do sprawowania nad nimi opieki.

W projekcie określono wszystkie obowiązki, jakie opiekun zwierzęcia ma wykonać w stosunku do swojego czworonożnego podopiecznego. Ponadto jednoznacznie określony zostanie mechanizm przydzielania przez służby wycofywanych zwierząt opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką zgodę. W przypadku gdy żadna uprawniona osoba nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Zaproponowano ponadto możliwość powierzenia przez jednostkę organizacyjną danej formacji opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W trakcie prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych uzupełniono przepis tak, aby objęto nim również psy służące w Straży Marszałkowskiej. Projekt ustawy nie przewiduje jednak rozwiązań regulujących sytuację zwierząt służących w ochotniczych strażach pożarnych. Dotyczy on tylko psów ratowników stanowiących własność osoby fizycznej będącej członkiem podmiotu włączonego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub podmiotu, z którym zawarto umowę cywilnoprawną. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż przepisami nie objęto zwierząt służących w Krajowej Administracji Skarbowej. Co prawda służba ta uregulowała te sprawy w osobnym rozporządzeniu, niemniej jednak warto by było, żeby zapisy były jednakowe dla wszystkich psów należących do tych służb. Pani Marszałek! Koalicja Obywatelska popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 1132.

Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Szczepański, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1132 i 1258. Od tysięcy lat niektóre zwierzęta służyły ludziom. W niektórych przypadkach zdolności psa nie zastąpi nowoczesna technika. Zadaniem zwierząt służących w służbach mundurowych jest pomoc w wykonywaniu zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Używane są przy zabezpieczeniu porządku publicznego, wykonują zadania patrolowe, tropią ślady ludzkie, wykrywają zapachy, niebezpieczne ładunki, narkotyki, szukają ludzi pod gruzowiskami. Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w marcu br. w Policji służyło 915 psów i 54 konie, w Straży Granicznej - 252 psy i 8 koni, a w Państwowej Straży Pożarnej służyło 25 psów. Utrzymanie tych zwierząt podczas służby regulują akty wewnętrzne. Brak jest uregulowań prawnych w zakresie postępowania w przypadku zwierząt wycofanych ze służby. Tylko w Państwowej Straży Pożarnej istnieje partycypacja w kosztach utrzymania psów. Niestety zdarzały się przypadki, że po zakończeniu służby niektóre zwierzęta były usypiane, a konie - oddawane na rzeź. W marcu Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w ramach swoich prac zapoznała się z sytuacją zwierząt służących w służbach mundurowych podległych resortowi ministerstwa spraw wewnętrznych. Już wówczas ministerstwo zapowiadało ten projekt. Cieszę się, panie ministrze, że po niecałych 3 miesiącach możemy dzisiaj nad nim debatować. Jak wiemy, prace były prowadzone we współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi. Przedłożony projekt ustawy reguluje status zwierząt służących w służbach mundurowych, tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej i Służbie Więziennej, od momentu doboru zwierzęcia do służby do czasu wycofania go z tej służby. W trakcie prac komisji przy aprobacie rządu do ustawy wpisano również psy służące w Straży Marszałkowskiej. Nie było akceptacji, tak jak mówiła moja koleżanka, czego również żałuję po rozmowie zarówno z panią minister Rzeczkowską, jak również z dyrektorem departamentu Ministerstwa Finansów, aby również psy służące w tej formacji objąć zapisami ustawy.

W omawianej dzisiaj ustawie zostały określone wymogi, które powinien spełniać opiekun zwierzęcia oddanego mu na emeryturę. Określone zostały obowiązki opiekunów zwierząt. Ustawa określa również zasady żywienia zwierząt, badań i profilaktyki oraz leczenia tych zwierząt. Doprecyzowuje przypadki, kiedy zwierzęta będą wycofane ze służby. Według ustawy zwierzęta nawet wycofane ze służby będą nadal pozostawały pod opieką formacji. Określony został również nadzór nad opiekunem zwierzęcia wycofanego ze służby. Pierwszeństwo w opiece nad zwierzęciem wycofanym ze służby będzie miał dotychczasowy opiekun, inny funkcjonariusz, pracownik jednostki, a w przypadku braku zainteresowania zajmie się nim stowarzyszenie bądź fundacja zajmująca się opieką nad zwierzętami. Na te zwierzęta opiekunowie będą otrzymywać świadczenia żywieniowe w naturze, organizacje społeczne - ekwiwalent w formie ryczałtu. Zwrot kosztów leczenia będzie następował na podstawie rachunków od weterynarza bądź za kupione leki. Zakazane będzie rozmnażanie zwierząt na emeryturze bądź używanie ich do celów zarobkowych. Kierownik jednostki będzie sprawował nadzór, czy opiekun sprawuje właściwą opiekę nad oddanym mu zwierzęciem, czy też ta opieka nie jest właściwa. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie zaaprobowała przedłożony przez rząd projekt ustawy. Mój klub będzie głosował za jego uchwaleniem. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi honor zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. To są druki nr 1132 i 1258. Podstawowym celem projektu jest kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w Siłach Zbrojnych i Służbie Więziennej. Kierunek zmian wytyczonych w przedstawionym projekcie jest bez wątpienia słuszny. W zasadzie muszę powiedzieć, że jest to jeden z bardzo nielicznych przypadków, gdy możemy stwierdzić, że przedłożenie rządowe jest przez nas w pełni akceptowalne. Psy i konie policyjne, niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji ustawowych zadań przez służby, są widoczne wtedy, gdy znajdują się na pierwszej linii. Potem, gdy wiek lub stan zdrowia nie pozwala już na ich wykorzystywanie, nagle nikną z pola widzenia rządzących. Nie oznacza to oczywiście, że nie można mieć do zaproponowanych rozwiązań szeregu uwag. Zasadniczo można uznać, że zasady pozyskiwania i wykorzystywania w służbie zwierząt - w praktyce odnosi się to do psów i koni - zostały określone w projekcie wystarczająco precyzyjnie. Wzięto pod uwagę opinie specjalistów, którzy z tym zagadnieniem mają do czynienia praktycznie od początku funkcjonowania formacji wykorzystujących zwierzęta w swoich działaniach. Ewentualne propozycje zmian są zatem nieznaczne.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Kilka lat temu Internet obiegło wzruszające zdjęcie pochodzące z Indii.

Słyszymy wiele historii o zwierzętach, które w bohaterski sposób pomagały w takich sytuacjach. Dla wielu z nich to codzienna praca wymagająca wyszkolenia, uwagi, panowania nad instynktami. Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie ok. 1200 psów i ponad 60 koni, a rocznie ok. 10% tych zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę.

Nieczęsto zdarza się, żeby w tak twardych obszarach jak obszary działania Sił Zbrojnych, Policji czy innych formacji uwzględniano aspekt emocji.

Można będzie również przekazać psa lub konia organizacji społecznej, ale tylko takiej, która statutowo zajmuje się ochroną praw zwierząt. Projekt zapewnia też dobre warunki emerytowanym czworonogom: wyżywienie, zabiegi profilaktyczne, leczenie, podstawowy standard, jaki w cywilizowanym państwie powinny otrzymać. A przecież te 9 lat dla psa i 15 lat dla konia, bo taki wiek emerytalny określają przepisy, to czasem dopiero połowa ich życia. Kiedy projekt ustawy był jeszcze w trakcie konsultacji rządowych, zapytaliśmy o zdanie zaprzyjaźnione organizacje. Ich reakcja była jednoznacznie pozytywna, a uwagi, jak np. dotyczące corocznej kontroli u weterynarza, finalnie znalazły miejsce w rozporządzeniu wykonawczym załączonym do projektu. Dobrym pomysłem było też poszerzenie zakresu formacji o Siły Zbrojne i Służbę Więzienną jeszcze na etapie prac rządowych. Polska 2050 przyjmuje projekt przedkładanej ustawy z dużym zadowoleniem. Może on liczyć na nasze poparcie. Chcielibyśmy jednak, aby również inne zwierzęta w Polsce, nie tylko te pracujące w służbach mundurowych, były traktowane w godny i jak najlepszy sposób. Wciąż czekamy na przepisy uwalniające je zza ciasnych klatek, zza małych kojców, zza krótkich łańcuchów. Procedowany projekt poprawi byt tysięcy psów i koni, które co roku będą odchodzić ze służby, ale pamiętajmy, że 10 mln zwierząt w Polsce jest każdego roku bezsensownie zabijanych na futra, a jeszcze więcej wciąż czeka na przepisy lepiej chroniące je przed okrucieństwem i złym losem. Ta ustawa to krok w dobrą stronę. Mało takich ustaw pozostawimy po sobie w tej kadencji. Ale ciągle jest szansa, że jeszcze ten Sejm zrobi więcej w kwestii praw zwierząt i że z tego zostaniemy wszyscy zapamiętani. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W tej ustawie mówimy o zwierzętach szczególnych, ponieważ to one bardzo często ratowały ludzkie życie, okazywały się nie do przecenienia podczas poszukiwań osób zaginionych, miały bezpośrednio wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Wątpię, że teraz te zwierzęta oglądają tę debatę. Myślę, że nie mają też aż takiej świadomości, jak ogromną rolę odegrały w naszym życiu. Natomiast my tę świadomość mamy. I myślę, że pojawienie się tej ustawy w Sejmie, jak również głosowanie za nią będzie najlepszym dowodem naszego szacunku i wdzięczności dla nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W rozdziale 8 art. 136 procedowanego projektu zostały wymienione osoby, instytucje, organizacje, które mogą sprawować opiekę nad wycofanym z użycia psem służbowym lub koniem służbowym. W dalszej części wymieniono, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zapewnić prawidłowe utrzymanie zwierzęcia po odbytej służbie. To bardzo dobry projekt, ale mam pytanie do ministerstwa. Czy nie warto byłoby rozszerzyć katalogu instytucji, którym można by było przekazać służbowe konie na tzw. zasłużoną emeryturę, o szkoły rolnicze? Oczywiście te, które spełniają warunki właściwego utrzymania zwierząt i mają odpowiednią bazę.

A przede wszystkim (Dzwonek) bezpośredni kontakt z żywą istotą z pewnością zaprocentowałby na przyszłość. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście ustawa dotycząca tzw. emerytur dla psów wykorzystywanych do celów specjalnych to odpowiedni krok, który wspieramy.

Czy rząd pracuje nad kwestiami związanymi z zakazem wykorzystywania zwierząt w cyrkach? Czy rząd pracuje nad kwestiami związanymi z obowiązkiem identyfikacji, czipowania psów oraz utworzenia centralnego rejestru, który by zapewniał to, że zwierzę zagubione będzie mogło być łatwo odnalezione przez właściciela? Obszar ochrony zwierząt jest bardzo ważny. Dzisiaj zajmujemy się tymi zwierzętami (Dzwonek), które były wykorzystywane, które służyły społeczeństwu, natomiast jeszcze jest kwestia tak naprawdę doprecyzowania wielu zapisów, które pozwolą powiedzieć, że mamy w Polsce dobrostan zwierząt. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący komitetu do spraw bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nareszcie pies, który przez lata pomaga ludziom, tropi przestępców, wykrywa narkotyki, ratuje z katastrof będzie miał prawo do emerytury i zasłużonego odpoczynku. To długo oczekiwana i bez wątpienia potrzebna zmiana. Ale skoro już poruszamy temat dobrostanu zwierząt, to gdzie reszta od dawna zapowiadanych przez prezesa partii rządzącej zmian? Wiem, że za ludźmi nie przepada, ale podobno kocha zwierzęta, więc: Co z zakazem hodowli na futra, z zakazem występowania zwierząt w cyrkach, z końcem rytualnego męczenia i zabijania zwierząt na mięso, z odejściem od męczenia psów i trzymania ich na łańcuchu? Pan poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewica. Panie Ministrze! Odmiennie niż pani posłanka Klaudia Jachira zakładam optymistyczny rozwój zdarzeń i zakładam, że jest to pierwszy z wielu, wielu projektów, które będą indywidualnie przedkładane jako piątka dla zwierząt. Tego życzę wszystkim nam.

Mam na myśli psy, które służą na terenie lotnisk, pomagają służbom celnym. Ale jest ustawa, ona powinna regulować prawa wszystkich psów i koni, które wykonują takie, a nie inne zadania.

Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Muszę powiedzieć, że jak się skończył ten lockdown. W sprawie tej ustawy.

Tak, dowiedzieliśmy się w komisji, że Krajowa Administracja Skarbowa ma swoje własne przepisy dotyczące tych zwierząt.

Państwowa służba powinna być ujęta w jednej ustawie i raczej dążyłbym do tego, żeby te instytucje też tam były. Bo może być coś takiego, że jedne psy będą miały lepiej, drugie gorzej, jak się jedne dowiedzą, to może drugie zaczną strajkować. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby w ramach całego pakietu opieki nad zwierzętami w trakcie pełnienia służby nie zapominać o tym, co dzieje się ze zwierzętami po odbyciu służby - w przypadku psów po 8 latach, w przypadku koni po 14 latach.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że przedmiotowa nowela będzie przyjęta pozytywnie przez wszystkich parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Zwierzęta takie jak psy i konie, które poświęcają całe swoje życie dla służby, są traktowane przez opiekunów i innych funkcjonariuszy formacji mundurowych jak partnerzy, których w wielu działaniach nie zastąpią zaawansowane technologie i które zasługują na godną egzystencję po wycofaniu ze służby.

I ostatnie pytanie: W skali roku ile środków trzeba zabezpieczyć, aby ta ustawa w sposób skuteczny weszła w życie? Pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Bardzo się cieszymy z tego projektu ustawy i z tych zapisów, ale jednocześnie pytamy, kiedy zakaz hodowli zwierząt na futra, kiedy zakaz trzymania zwierząt na stałej uwięzi.

W SOK-u takich psów jest ok. 100, są to głównie wilczury. Jest więc pytanie, czy takie zwierzęta także z taką systemową ochroną się spotkają. I druga kwestia, kwestia pseudohodowli. Chciałam się spytać, czy państwo jakoś zamierzacie kontrolować to, czy psy, które są wykorzystywane w służbie dla państwa, pochodzą z normalnych, zdrowych, pełnowartościowych hodowli. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Natomiast tak jak już mówili moi przedmówcy, mam nadzieję, że jest to początek pewnej drogi, albowiem zwierząt, które służą nie tylko w instytucjach rządowych, ale także samorządowych, chociażby w strażach miejskich, jest bardzo wiele. Wydaje się, że nie powinno być tu rozróżnienia: psy, konie czy inne zwierzęta, które służą chociażby w Policji, i na te, które służą w służbach samorządowych. Natomiast chciałbym zapytać, jaką kwotę rząd zabezpieczył na rok bieżący i na rok przyszły, aby zapewnić skuteczne wykonanie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To jest czas, aby złożyć podziękowania wszystkim osobom z wszystkich ugrupowań politycznych, jak również panu ministrowi za wspólną pracę włożoną w ten projekt. Uchwalenie tej ustawy jest oczywiście naszym ponadpartyjnym obowiązkiem i sądzę, że nikt nie będzie polemizował z tak postawionym pytaniem. Ponadpartyjna debata i wspólna praca posłów z rządem musi budzić uznanie. Mam jednak pytanie do rządu: Czy ustawa nie powinna obejmować wszystkich zwierząt: psów i koni wykonujących prace w polskich służbach?

Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! To ważny projekt, zwłaszcza że budowany w szerokim porozumieniu, ponad podziałami politycznymi, wyznaczający też określone standardy dla innych służb publicznych, które wykorzystują psy i konie na potrzeby służby. Jeśli dzisiaj ten projekt nie obejmuje właśnie m.in. psów i koni, które funkcjonują w służbach, np. w strażach miejskich, to też wyznaczamy określone standardy, z których te jednostki mogą również korzystać.

Ile będzie wynosiło to w całości, jeśli chodzi o zabezpieczenie tejże ustawy? Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Dyduch, klub Lewica. Wysoki Sejmie!

Dzisiaj mamy ogromny postęp w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, i za to chwała i tej Izbie, i sposobowi myślenia w naszym kraju.

Ja chciałbym się dowiedzieć, jak do tej pory były rozwiązywane te problemy, jeżeli chodzi o zwierzęta, które skończyły służbę. W jakiej skali one były usypiane, np. konie po skończeniu tej służby, i w jakiej skali były usypiane psy? Po prostu czy to była praktyka powszechna, czy jednak one podlegały jakiejś ochronie? Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Izbo! Jak powszechnie wiadomo, psy wykorzystywane w służbach, dobrze wyszkolone potrafią zastąpić pracę wielu ludzi i okazują się często szybsze i skuteczniejsze od urządzeń lokalizacyjnych. W przypadku straży pożarnych w Polsce zwierzęta te pełnią służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W uzasadnieniu czytamy, że procedowana ustawa to odpowiedź na poczucie etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom wycofanym z użycia. Dlaczego zatem nie przewiduje się rozwiązań regulujących sytuację wszystkich psów służących w ochotniczych strażach pożarnych, lecz tylko psów w tych jednostkach, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? Z etycznego punktu widzenia byłoby wskazane, żeby wszystkie psy (Dzwonek) służące mogły być traktowane jednakowo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani Marszałek! Chciałabym dopytać może o to, o czym przed chwilą mówiła moja koleżanka, żeby to było dobrze zrozumiane i żeby ci, którzy mają być objęci tą ustawą, tym uregulowaniem, również mogli to jasno wiedzieć. Chodzi o status psów.

Czy należy uważać, że pies kontraktowy to również pies, który służy w OSP? Tu bardzo bym prosiła pana ministra, żeby odpowiedział na to pytanie. No i oczywiście już kilka razy przywoływane były konie. Tutaj też chciałabym zapytać i jak gdyby podkreślić to, co mówili przedmówcy: Czy konie w straży miejskiej nie powinny również zostać objęte tą regulacją? Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O odpowiedź na pytania pań i panów posłów bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Błażeja Pobożego. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim państwu za konstruktywną dyskusję podczas pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także za tę dzisiejszą debatę, za wszystkie pytania, sugestie, wszystkie głosy. Bardzo za to jednoznacznie dziękuję. Bardzo również chciałbym podziękować za to - jednoznacznie pozytywnie oceniam ten fakt - że tą najważniejszą, kluczową i chyba jedyną w pełni merytoryczną poprawką była inicjatywa objęcia naszą regulacją również psów służbowych Straży Marszałkowskiej. Przy tym od razu powiem: my czekaliśmy po prostu na taką poprawkę i dobrze, że ona się pojawiła. Proszę pamiętać, że pierwotnie projekt dotyczył tylko zwierząt odbywających służbę w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, zresztą będę o tym za chwilę mówił. I przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że podczas pierwszego czytania nasz projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został przyjęty jednogłośnie. Rzeczywiście jest tak, że rzadko przedstawiciel rządu ma przyjemność usłyszeć tyle dobrych słów o rządowym przedłożeniu, bo wszyscy tak naprawdę ten projekt poparli i wyrazili to nie tylko w swoich wystąpieniach, ale także w głosowaniu, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo! Zadaniem zwierząt znajdujących się w służbach jest wspomaganie funkcjonariuszy w realizacji ustawowych zadań. I rzeczywiście jest tak, że pomimo znacznego postępu oraz rozwoju nowych technologii zwierzęta nadal odgrywają istotną, kluczową rolę, stanowiąc realne wsparcie funkcjonariuszy, a w niektórych przypadkach są wręcz niezastąpione. Wspomagają realizację zadań związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego w ramach akcji poszukiwawczych, prowadzą działania wykrywcze związane z poszukiwaniem sprawców przestępstw lub ofiar tych przestępstw, prowadzą działania zapobiegawcze dotyczące wykrywania niebezpiecznych substancji. Wreszcie, o czym też powinniśmy pamiętać, odgrywają istotną rolę ceremonialną podczas rozmaitych oficjalnych uroczystości państwowych. W ocenie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczasowe rozwiązania dotyczące sytuacji zwierząt w formacjach mundurowych były i nadal są niewystarczające. Właśnie dlatego kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac nad kompleksowym uregulowaniem statusu zwierząt wykorzystywanych w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarówno w odniesieniu do zwierząt używanych do wsparcia realizacji zadań ustawowych, jak i tych - bo od początku ta idea nam przyświecała - wycofanych ze służby.

Przypomnę, pierwsza wersja dotyczyła tylko i wyłącznie uregulowania statusu zwierząt w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mówiono we wszystkich niemal wystąpieniach, że psy i konie służą w Policji, Straży Granicznej, w Siłach Zbrojnych, a psy w Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej i w Straży Marszałkowskiej. Szanowni Państwo! Chciałbym wyraźnie podkreślić - bo ten wątek się tutaj nie pojawił, ale wydaje mi się, że dobrze, aby wybrzmiał z tej mównicy - że niniejszy projekt nie wyłączy stosowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt. On stanowi jej dopełnienie, odnosząc się do zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych. Zgodnie z art. 4 pkt 20 wspomnianej ustawy o ochronie zwierząt poprzez zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych rozumie się zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe zasady działania służb oraz zasady szkolenia i wykorzystywania psów. Natomiast do tej pory brakowało odrębnych przepisów - one tą ustawą są wprowadzane.

W naszym projekcie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu doboru ich do służby, poprzez cały okres trwania tej służby, aż po wycofanie z użycia w formacjach. Natomiast w dalszym ciągu zastosowanie będzie miał przykładowo art. 15 ustawy o ochronie zwierząt, określający zasady postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych. Szanowni Państwo! Przechodząc do krótkiego omówienia głównych założeń projektu, należy wskazać, że w określono w nim warunki, jakie powinien spełniać opiekun, któremu przydziela się zwierzę w poszczególnych formacjach; obowiązki opiekunów zwierząt; zasady żywienia zwierząt; zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu oraz sposób ich finansowania; zasady postępowania w sytuacjach nagłych, w których zagrożone jest zdrowie lub życie zwierząt; wreszcie przypadki wycofania zwierząt z użycia w poszczególnych formacjach; bardzo szczegółowo rozpisany mechanizm powierzania opiekunom zwierząt wycofanych z użycia przez służby - przy założeniu, i to jest zmiana kluczowa, że na zawsze pozostaną one na stanie i pod opieką formacji, w której dotąd służyły. Ma to znaczenie dlatego, że jeden z podstawowych deficytów wcześniejszych, tych ledwie szczątkowych regulacji wewnętrznych w poszczególnych służbach dotyczył sprawowania nadzoru. Teraz ta ustawa określa również zasady sprawowania nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad tym, jak ta opieka nad powierzonymi zwierzętami wycofanymi ze służby jest sprawowana. A zatem, w kontekście wspomnianego nadzoru i innych kwestii, które wymieniłem, należy wskazać, że ten projekt ma charakter uzupełniający względem rozwiązań przyjętych w ustawie o ochronie zwierząt.

Pierwsze czytanie miało zgodny i koncyliacyjny charakter, bo my te poprawki - w cudzysłowie poprawki - uwzględnialiśmy już na tamtym etapie. Właśnie zdecydowaliśmy o tym, że w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt na wniosek opiekuna komendanci określonych służb i formacji będą mogli objąć tymi przepisami także zwierzęta, które zostały wycofane ze służby przed wejściem w życie tej ustawy. To jest kluczowa sprawa, zwłaszcza dla takich instytucji i organizacji społecznych, których celem jest ochrona zwierząt, jak wspomniana przez m.in. panią poseł sprawozdawcę ta organizacja, to schronisko, ten azyl, o którym mówiliśmy.

Po pierwsze, bardzo dziękuję za głosy jednoznacznie wspierające i deklarujące poparcie dla tej ustawy.

Po pierwsze, chcę jeszcze raz przypomnieć, że wyjściowo był to projekt dotyczący zwierząt wykorzystywanych w służbach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z art. 64 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który określa sytuację zwierząt służbowych używanych w ramach kontroli celno-skarbowej, w drodze rozporządzenia uregulowano ich status oraz warunki, w których pozostają one pod opieką opiekunów.

Zgodnie z art. 2 ustawy o strażach gminnych straż gminną może utworzyć rada gminy i ten sam organ może ją rozwiązać.

Jest to jednostka organizacyjna gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy, mówi o tym art. 5 ustawy o strażach gminnych. W związku z tym trudno byłoby nam nakładać na władze gminne obowiązki o charakterze stałym.

Myślę, że mamy dziś możliwość dać dobry przykład i jeśli poszczególne samorządy będą chciały pójść za tymi rozwiązaniami, to będzie bardzo dobrze.

Finansowanie będzie w ramach obowiązujących limitów w poszczególnych formacjach.

Wtedy, gdy ktoś decyduje się na włączenie dodatkowego zwierzęcia, bierze na siebie ten koszt. Wysoka Izbo! Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że ten projekt wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom, oczekiwaniom samych funkcjonariuszy, ale nie tylko ich. Wszystkie te oczekiwania, myślę, mają swoje źródło w poczuciu naszego wspólnego etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom w służbie i tym wycofywanym ze służby.

Wierzę, tak jak wspomniałem podczas pierwszego czytania projektu w czasie prac komisji, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami politycznymi i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Dziękuję. Domyślam się, że i poseł sprawozdawca, czyli pani poseł Katarzyna Piekarska, będzie chciał zabrać głos, odpowiadając na pytania postawione przez panie i panów posłów. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy! W zasadzie pan minister odpowiedział już na wszystkie pytania, które były zadane.

Ja za tę debatę również dziękuję. Bardzo ciekawy wątek poruszyła pani posłanka Rosa, mianowicie chodzi o pozyskiwanie psów. Mam taką prośbę, żeby służby, które będą się tym zajmowały, rzeczywiście dopilnowały tego, aby psy, które trafiają do funkcjonariuszy, były z wzorcowych hodowli, żeby to nie były te tzw. pseudohodowle.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych celem przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1259 i 1296) Uprzejmie proszę panią poseł Annę Kwiecień o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, na którym rozpatrywany był przytoczony projekt.

W związku z tym uprzejmie proszę Wysoką Izbę, Wysoki Sejm o przyjęcie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Katarzyna Czochara. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1259. Proponowane zmiany w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych obejmują zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym, gospodarczym i zdrowotnym COVID-19. Proponowane zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia zakresu działalności agencji o eksperymenty badawcze, wspierania przez agencję oprócz badań klinicznych także nowych eksperymentów badawczych i doprecyzowania regulacji dotyczących funkcjonowania agencji, których dotychczasowe stosowanie powodowało utrudnienia w sprawnej realizacji zadań ustanowionych przez agencję. Rozszerzenie zakresu zadań agencji o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przez możliwość udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych będzie miało istotne znaczenie w pozyskiwaniu nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zwiększających m.in. możliwość zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu można będzie uzyskać wsparcie finansowe z agencji nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze, co może znacząco wpłynąć na pobudzenie tego rodzaju działalności, a tym samym przyczynić się do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę z tego miejsca również podkreślić, iż proponowane zmiany ww. ustawy były wielokrotnie podnoszone przez przedstawicieli środowisk medycznych jako postulat rozszerzenia przedmiotu zadań agencji również o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia w przypadku eksperymentu badawczego. Proponowana zmiana jest także zgodna z kierunkiem realizowanej polityki w zakresie innowacyjności w ochronie zdrowia, dla której strategicznym odniesieniem jest przyjęty przez rząd dokument „Polityka lekowa państwa” Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii albo uzgodnienia projektu. Projektowana ustawa będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój innowacyjnych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje ww. ustawę i rekomenduje jej przyjęcie. Pani Marszałek! Również w imieniu klubu parlamentarnego pragnę przedłożyć sześć poprawek. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Rajmund Miller. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw.

W uzasadnieniu, jeżeli chodzi o to, co przedstawiła moja przedmówczyni, mówi się o wpływie tych badań, które są zakładane, na gospodarkę, na zdrowie, na różne inne dziedziny życia publicznego w naszym kraju. Przede wszystkim, jeżeli państwo przeanalizujecie opinię BAS-u, opinia BAS-u jest krytyczna wobec zapisów tej ustawy. Po pierwsze, nie może być tak, że eksperci będą powoływani nie na zasadzie ustawy o zamówieniach publicznych, tylko tak sobie. Nie trafia do nas wyjaśnienie, że nie ma ekspertów na rynku. Dlaczego ten sam ekspert, który będzie opiniował celowość danych badań, będzie również kontrolował te badania? O pozostałych powie pani poseł Elżbieta Gelert, która uzupełni moją wypowiedź, dlatego że mamy również wiele innych wątpliwości co do zapisów tej ustawy. Proszę państwa, mam zaszczyt przedłożyć pani marszałek dwie poprawki do tej ustawy. Dobrze, dziękuję bardzo.

Dziękuję, panie pośle. Wysoka Izbo! Pani Minister! Nasze wątpliwości budzi również zapis o eksperymentach medycznych.

Prosilibyśmy o odpowiedź na to pytanie.

Finansowo wszystko pasuje. Owszem, proszę państwa, finansowo w każdym zakładzie będzie pasowało, jeżeli się bada plan po korektach. Jeżeli korekty są zrobione w odpowiednim czasie, to nie ma problemów, wtedy wszystko jest zgodnie z planem. Natomiast chciałabym zauważyć, mówił o tym poprzedni kolega, że są to pieniądze, które pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, proszę państwa. I zamrożenie teraz niewydanych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo niekorzystne dla pacjentów, przede wszystkim dla pacjentów. Są to nasze składki, więc bardzo byśmy prosili, żeby tu powiedzieć, dlaczego te pieniądze mają być zamrożone.

Podejście do naszych poprawek będzie warunkowało nasze stanowisko co do projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Marek Rutka w imieniu klubu parlamentarnego Lewica.

Wysoka Izbo! Zdrowie nie powinno mieć ceny. Batalia o powrót do zdrowia całego społeczeństwa powinna być prowadzona w sposób przemyślany, w sposób systemowy. Niestety należy przyznać, że tej systemowości, gdy mówimy o kwestiach zdrowotnych, często brakuje. Działania rozrzucone są po wielu ministerstwach, instytucjach, agencjach. Ich działania bardzo często są nieskoordynowane. To wszystko obniża z jednej strony skuteczność podejmowanych działań, a z drugiej zwiększa koszty tychże działań. Agencja Badań Medycznych jest instytucją pożyteczną i na pewno warta jest rozwijania. Pytanie jednak: Czy wszystkie proponowane w przedłożeniu zmiany zmierzają w kierunku właściwym? Zapis ten przyznaje prezesowi agencji prawo do jednoosobowego, arbitralnego rozpatrywania odwołań i protestów. Stąd też klub Lewicy podczas pierwszego czytania złożył poprawkę, która obliguje prezesa agencji do tego, aby decyzja w przypadku protestu została podjęta po zasięgnięciu opinii rady. Poprawka miała na celu zwiększenie demokratyzacji całego procesu, a na pewno zwiększenie transparentności podejmowanych decyzji.

W grę wchodzą przecież znaczne pieniądze, znaczne kwoty publicznych środków, a doświadczenie uczy, że jednoosobowe podejmowanie decyzji w kwestiach finansowych może nasuwać szereg zastrzeżeń, a przynajmniej wątpliwości, żeby nie powiedzieć: podejrzeń.

Prace badawczo-rozwojowe dotyczą m.in. opracowania, jak czytamy w ogłoszeniu, skutecznej szczepionki na COVID-19. Można byłoby dodać: narodowej szczepionki.

Ten budżet został rozdysponowany na 87 projektów. Mówimy: jednostkowo to nie jest dużo. I teraz odniosę to do kosztów, jakie poniesiono czy jakie rządy krajów poniosły na opracowanie skutecznych, działających już i wdrożonych do produkcji szczepionek przeciw COVID-19.

Przypomnę: całkowity budżet agencji to 1 mld. Natomiast jeśli podliczymy wszystkie wydatki, jakie poniosły rządy Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a więc tych krajów, które opracowały i zarejestrowały skuteczne szczepionki, mówimy o kwocie 22 mld zł. Te kwoty wyglądają zdecydowanie inaczej, oczywiście bardziej imponująco, niż cały budżet agencji. Tutaj warto skupić się na tym, aby te środki publiczne, nie tak duże, ale jednak znaczne, były wydatkowane w sposób właściwy. Mamy doświadczenia chociażby z projektem budowy polskich samochodów elektrycznych, których miało już po naszych drogach jeździć ok. 1 mln. Okazało się, że spółka ElectroMobility Poland, która tak dumnie ogłaszała, że będziemy mieli polski samochód elektryczny. Polski - to jest tylko nazwa, ponieważ jest to wspólne dzieło inżynierów z Niemiec, z Włoch, natomiast jeśli chodzi o Polskę, zostały pieniądze i marka. No i pytanie: Czy w przypadku tej szczepionki z Polski to nie będzie tylko fiolka? Tak wygląda sytuacja z wydatkowaniem środków, co zresztą też zawarte jest w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska pan poseł Dariusz Klimczak. Wysoka Izbo! Agencja Badań Medycznych jest stosunkowo nową instytucją, ale generalnie opinię ma dobrą, dobrze jest oceniana. Dzisiaj są proponowane zmiany, nowelizacja ustawy.

Uważam, że możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, w tym niekomercyjne, ale także na eksperymenty badawcze jest posunięciem dobrym.

Nie podoba mi się wprowadzanie dobrowolności przy wyborze ekspertów, generalnie to, co państwo proponujecie, ta dobrowolność, wskazywanie tych, których uważacie za słusznych, którzy będą współpracować z agencją. W ogóle taki wybór ekspertów przypomina mi dobór ekspertów z komisji pana Macierewicza. Nie chciałbym, żeby w tak poważnej instytucji tego typu zjawiska miały miejsce, tym bardziej że znamy bardzo wiele różnych innych instytucji, w tym samorządowych, gdzie dobiera się ekspertów i nie ma żadnego problemu w oficjalnym ogłaszaniu naborów i przeprowadzaniu procedury konkursowej w trybie zamówień publicznych, tym bardziej że Prawo zamówień publicznych jest naprawdę bardzo elastyczne i można z tego skorzystać, a wtedy jesteśmy transparentni. Tym bardziej przy instytucji tak specjalistycznej i tak specyficznej, która wymaga ogromnego bezpieczeństwa, i tym bardziej że z dużym trudem przeznaczamy pieniądze na jej działalność i wszyscy chcielibyśmy, nie tylko w tej Izbie, ale w całym społeczeństwie, żeby była właściwa kontrola nad wydatkowaniem tych pieniędzy.

Jeżeli chodzi o tzw. niewygasy, uprawnione jest stwierdzenie, że w tak specjalistycznej instytucji, gdzie wszystko powinno być precyzyjnie zaplanowane, trudno jest o wprowadzanie przepisów o wykorzystaniu środków z odpisu niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym. Tym bardziej że tych pieniędzy naprawdę nie ma zbyt wiele, więc ich wydatkowanie powinno być planowane bardzo precyzyjnie i szczegółowo. Osobnym wątkiem jest cała druga część ustawy, po co jest to w tym momencie wprowadzane. Pani minister próbowała bronić swojej tezy i podawać argumenty, że w tym momencie jest to bardzo potrzebne, natomiast uważam, że powinniśmy podnosić standardy legislacji w parlamencie. Jeżeli jest potrzeba standaryzacji prawa wykonywania zawodów i innych przepisów, które dotyczą pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów itd., itd., to powinniśmy to po prostu robić. To żadna różnica, gdybyśmy to zrobili w innym akcie legislacyjnym. To są nasze uwagi i od przyjętych poprawek, odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości zależy nasza decyzja klubowa. Uważamy, że od samego początku można było inaczej poprawić nowelizację tej ustawy, niepotrzebnymi sprawami państwo naruszacie wizerunek tej nowej, dosyć dobrze ocenianej instytucji. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Wysoka Izbo! Mówimy o Agencji Badań Medycznych, która może i powinna pełnić bardzo ważne funkcje, bo badania są bardzo ważne. Badania muszą być oparte na naukowych wzorach, prowadzone zgodnie z naukową metodą, to nie ma być, rozumiem, transmisja od decyzji polityków i potem tłumaczenie ludziom, dlaczego politycy mieli rację albo nie mieli racji, tylko po prostu mają być badania.

Najważniejsze, żeby to były badania naukowe, a więc żeby były obiektywne, dlatego też np. nie wyobrażam sobie, żeby w naukowej instytucji połowa badaczy to nie byli, załóżmy, proszczepionkowcy, a połowa antyszczepionkowcy.

To mają być badania, powtarzam jeszcze raz, z których to badań ma wynikać pewna prawda obiektywna.

Ale, Wysoka Izbo, w badaniach naukowych istotne jest to, na co wydajemy pieniądze, a cenzura roczna jest bez żadnego znaczenia.

Te pieniądze trzeba zostawić agencji, żeby wydała w roku przyszłym, i być może na ten projekt, a być może będzie jakaś ważniejsza sprawa, np. zamiast szczepionek na COVID pojawi się lekarstwo na COVID i trzeba będzie badać, co jest znacznie ważniejsze, np. lekarstwo na COVID.

Co robiono? Więc ten rok powinien mieć wyłącznie znaczenie sprawozdawcze, natomiast nie powinien być żadną barierą do zmiany decyzji, przesuwania decyzji, przedłużania decyzji, rok nie powinien być żadną, powtarzam, żadną cezurą w tego typu pracach naukowych. Proszę państwa, badania, powtarzam, naukowe.

Proszę państwa, najwięksi cwaniacy spełniają kryteria obiektywne, załatwiają sobie specjalnie, co trzeba, żeby mieć spełnione te kryteria, a potem mogą nic nie wiedzieć, mogą umieć tylko jedno: spełniać obiektywne kryteria.

Żeby tylko pod tym płaszczykiem nie kryło się właśnie tworzenie jakichś specjalnych programów, przy których miałaby się pożywić rządząca aktualnie partia polityczna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie tworzymy nigdy idealnych przepisów mimo najwyższych chęci. W związku z tym każda ustawa wymaga co pewien czas weryfikacji z powodu rozsądku. Również ta o Agencji Badań Medycznych, jak widać z przedłożenia rządowego, wymaga poprawy, uzupełnienia.

One oczywiście były dyskutowane, wymagają na pewno rozwagi. Uważam akurat, że generalnie zmierzają one ku rozszerzeniu możliwości dobrego funkcjonowania agencji. Są oczywiście takie kwestie, które budziłyby z naszego doświadczenia wątpliwości dotyczące właśnie procedowania w trybie przetargowym, np. powoływania kogoś, kogo w ogóle rzeczywiście nie tak łatwo pozyskać. To było argumentowane. Są więc pewne rzeczy, które może też będą dalej niedoskonałe, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam eksperyment badawczy, jest to rzecz oczywiście zupełnie zrozumiała, regulowana w polskim prawodawstwie w ustawie o zawodzie lekarza, opisana, zdefiniowana. Jeżeli chodzi o troskę o to, żeby nie było gorzej niż w Europie, to właśnie o to chodzi, żeby nie było gorzej w ogóle niż w świecie, żebyśmy tutaj mogli otworzyć się na to. Natomiast rzeczą, która budzi najwięcej wątpliwości, jest to, że ni stąd, ni zowąd w ustawie o Agencji Badań Medycznych pojawiło się kilka artykułów - w sumie na dziewięć artykułów. siedem artykułów niedotyczących w żadnym wypadku Agencji Badań Medycznych. Szczęśliwie dotyczy to w ogóle zagadnień związanych z opieką zdrowotną, a nie z jakimiś zupełnie innymi sprawami, ale dotyczy to też sprawy trudnej, o tyle trudnej, tzn. już nie trudnej. Po prostu dotyczy to uprawnień samorządów zawodowych zawodów medycznych. Wydawanie prawa wykonywania zawodów medycznych jest jednym z podstawowych zadań samorządów zawodów medycznych opisanych ustawowo wcześniej.

Najgorsze jest to, że w żadnym wypadku nie uzyskano opinii żadnego z samorządów zawodów medycznych, które zostały pozbawione pewnych uprawnień.

W tej chwili jest to nic innego jak pomieszanie nieudolności z arogancją wobec setek tysięcy polskich lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych. Naprawdę nie powinno to mieć miejsca. Szkoda, że tak się dzieje, bo rzeczywiście była okazja, żeby kolejny raz to uszanować. Natomiast w związku z tym, że uważamy, że nie powinno to mieć miejsca, chciałem przedłożyć pani marszałek poprawkę koła dotyczącą właśnie skreślenia tych artykułów, co zresztą proponowałem też na posiedzeniu komisji. Myślę, że również dla wnioskodawców, pomysłodawców lepiej by było, żeby to przepracować i w zupełnie innym trybie procedować nad uzgodnieniem tego z samorządami, bez niepotrzebnego rzeczywiście odsunięcia ich od wpływu na swoje zadania. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ramach dyskusji o ustawie o Agencji Badań Medycznych chciałem się odnieść do bardziej ogólnej sprawy.

Agencja Badań Medycznych finansowana jest przede wszystkim z pieniędzy, które ubezpieczeni zbierają na swoje leczenie, na świadczenia medyczne.

Co jakiś czas odzywają się głosy, że brakuje na leczenie tego lub innego pacjenta. Jeżeli te lub inne świadczenia nie są finansowane, to miejmy świadomość, że kilkaset milionów złotych przeznaczonych na leczenie pacjentów bez ich zgodny - oczywiście Sejm jako reprezentant tych pacjentów to zalegalizował - przeznaczanych jest nie na ich leczenie, tylko na badania i eksperymenty medyczne. To jest grzech pierworodny.

W związku z tym będziemy przeciwni jakimkolwiek działaniom związanym z Agencją Badań Medycznych, dopóki nie zostanie rozwiązany problem jej finansowania.

Przechodzimy do pytań. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Temat jest niezwykle ważny, ponieważ chodzi o 213 mln zł rocznie. To są środki z naszych składek zdrowotnych.

Czym są badania medyczne? Mówi się, że Agencja Badań Medycznych to dziecko pana ministra Szumowskiego.

Ta nowelizacja ma przede wszystkim uczynić wydawanie tych środków jeszcze bardziej nietransparentnym. Chcecie wyłączyć z zamówień publicznych wybór (Dzwonek) ekspertów zewnętrznych do oceniania wniosków. Chcecie również ograniczyć możliwość złożenia protestu od wyników konkursów. Wreszcie, chcecie rozszerzyć eksperymenty badawcze na eksperymenty medyczne przeprowadzane na ludziach.

Bardzo proszę.

Bardzo proszę o wskazanie, o jakie inwestycje chodzi.

Brakuje nam pieniędzy na leczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Pani Marszałek!

Kiedy z panem posłem Szczerbą zapukaliśmy do drzwi tej agencji w 2020 r., okazało się, że brat pana ministra Szumowskiego, który zainwestował w jedną spółkę, został udziałowcem kolejnej.

Teraz do ustawy o Agencji Badań Medycznych jest dopisywane, że wyłącza się stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie. Czy to jest prywatna firma pana ministra Szumowskiego i PiS-u, która będzie rozdawała miliardy złotych na prawo i lewo? Co to w ogóle jest?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Typowa sytuacja. Sam pomysł, żeby zwiększyć uprawnienia Agencji Badań Medycznych, jest jak najbardziej dobry. Czekamy na technologie innowacyjne, na postęp.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu tej ustawy czytamy: Dzięki proponowanemu rozwiązaniu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego z agencji nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze, co może znacząco wpłynąć na pobudzenie tego rodzaju działalności, a tym samym przyczynić się do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Czy ewentualne nakładanie na Agencję Badań Medycznych zadań związanych z tworzeniem szczepionki oraz leków na COVID-19 nie będzie aby działaniem spóźnionym o 2 lata, przejawem megalomanii władzy, przykładem propagandy sukcesu za wszelką cenę, bez uwzględnienia czynników ekonomicznych? Jeżeli Polska ma ambicję bycia producentem szczepionek, to istnieje dużo prostsza metoda niż zaczynanie badań od zera. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Wysoka Izbo! Projekt ustawy rozszerza zakres działalności Agencji Badań Medycznych. Cel jest słuszny, ale przedstawione zapisy ustawy są bardzo złe, wręcz korupcjogenne. To po prostu dzielenie łupów.

Po prostu żyć nie umierać.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!

Mam pytanie.

Jakie osiągnięcia ma ta agencja?

Dziękuję bardzo. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu zadań Agencji Badań Medycznych o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia. Pragnę przypomnieć, że w lutym br. wspólnie z grupą posłów zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy zamierza refundować możliwość terapii za granicą w przypadku chorób onkologicznych i rzadkich, gdy terapie dostępne w Polsce nie uratują zdrowia lub życia pacjenta. Resort zdrowia poinformował nas wówczas, że nie widzi możliwości takiej refundacji, chce za to rozwijać i szerzyć wiedzę na ten temat. Pragnę podkreślić, że ulotkami finansowanymi z budżetu państwa, audycjami radiowymi rząd nie pomoże pacjentom. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie, kiedy Polki i Polacy uzyskają dostęp do refundowanego, innowacyjnego, nowoczesnego, ratującego ludzkie życie leczenia dostępnego za granicą. Dziękuję bardzo.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że te wszystkie ustawy to gmeranie w systemie, który nie ma szans dobrze działać. Szpitale już te pieniądze mają i nie muszą konkurować o pieniądze, które szłyby za pacjentem, jakością usług i efektywnością wykorzystania tych środków.

Jak komuna była w żywności, to były wielkie kolejki, tak jak dzisiaj w ochronie zdrowia, i mały, delikatnie mówiąc, wybór asortymentu - tak jak dzisiaj w ochronie zdrowia. Trzeba pozbyć się komuny w ochronie zdrowia i wtedy będziemy mieli szansę na normalny system ochrony zdrowia. W tym momencie to jest tak, jakby mieć chorobliwie grubego (Dzwonek) grubasa i przypudrować mu nosek, zamiast go odchudzać, żeby ratować mu zdrowie i życie.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Ile będzie wówczas wynosił ten odpis i na co w agencji zostanie przeznaczony? Druga rzecz to pomoc osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji, a walczącym chociażby, jeśli chodzi o małe dzieci, z taką chorobą jak SMA. Tutaj rodzice robią wszystko (Dzwonek), zbierają za pomocą fundacji środki finansowe. Państwo stoi z boku. Pani poseł Anna Kwiecień, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystać w Polsce potencjał rozwoju badań medycznych i naukowych dotyczących zdrowia, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, które przed powstaniem agencji stanowiły 2% wszystkich zarejestrowanych badań. To naprawdę znikomy procent w porównaniu z innymi państwami. Dla porównania w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi ok. 40%. Celem agencji jest zwiększenie odsetka niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu co najmniej 30%.

Dlatego bardzo proszę panią minister o ponowne przedstawienie argumentów, które przemawiają za tym, aby pozostały tzw. niewygasy, czyli środki, które w danym roku nie zostały wykorzystane, a które można wykorzystać w roku następnym. Wysoka Izbo! Dla pieniędzy wydatkowanych na naukę mówimy: tak, dla pieniędzy wydatkowanych na badania naukowe mówimy: tak, ale dla pieniędzy, które mają być wydatkowane przez Agencję Badań Medycznych, pieniędzy pochodzących z NFZ, które agencja chce wydawać bez żadnej procedury, bez żadnego przetargu, bez żadnego nadzoru, mówimy stanowczo: nie.

Bardzo proszę o informację, czy zapisy, które znajdują się w projektowanej ustawie, dotyczące właśnie eksperymentów są zgodne z ustawodawstwem unijnym, z prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 kluczowe znaczenie mają wszelkie działania stymulujące konkurencyjność i innowacyjność przemysłu farmaceutycznego. Polskie firmy są potentatem w skali europejskiej w dziedzinie produkcji substancji czynnych. Warto podkreślić, że w pierwszej fazie epidemii koronawirusa wiosną ub.r. najwięksi wytwórcy substancji czynnych na świecie, a więc Chiny i Indie, wstrzymali eksport komponentów do produkcji leków i tylko dzięki polskim firmom farmaceutycznym nie doszło do załamania się dostaw leków stosowanych m.in. w terapii respiratorowej. Dziękuję. Pan poseł Paweł Szramka, Polskie Sprawy. Wysoka Izbo! Mój kolega z Koła Poselskiego Polskie Sprawy poseł Andrzej Sośnierz mówił o tym, że środki na działanie agencji pochodzą z naszych składek zdrowotnych. Nie jestem przekonany co do tego, czy Polacy zgadzają się z takim stanem rzeczy. Dlatego bardzo proszę stronę rządową o odpowiedź na pytanie: Czy istnieje sposób na zmianę finansowania tej agencji, aby środki na jej działalność nie pochodziły z budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia? Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania postawione przez panie i panów posłów odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani minister Anna Goławska. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy ma na celu usprawnienie i uelastycznienie pracy Agencji Badań Medycznych, która - jak tutaj wielokrotnie padło - jest bardzo ważną instytucją, jeśli chodzi o rozwój nauk o zdrowiu, rozwój firm farmaceutycznych czy rozwój nowoczesnych terapii leczenia chorób, które są bardzo skomplikowane, rzadkie i na które niejednokrotnie dotychczas nie wynaleziono sposobu leczenia. Podnoszone uwagi dotyczące wyboru ekspertów są nie do końca słuszne z uwagi na to, że ta procedura jest już opisana na stronach internetowych. To nie jest tak, że brak zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych powoduje, że eksperci są wybierani w sposób niejawny, niejasny czy nieklarowny. Otóż są określone zasady, kryteria naboru ekspertów. Każdy, kto spełnia wymogi określone przez Agencję Badań Medycznych, może się zgłosić i brać udział w pracach związanych z wyborem, oceną, rozliczaniem projektów czy dokonywaniem analiz. Takie zasady stosowane są nie tylko w przypadku ekspertów wybieranych w Agencji Badań Medycznych, lecz również np. w przypadku środków europejskich, w odniesieniu do których nie jest stosowana

Już dzisiaj są przepisy, które mówią, w jaki sposób należy prowadzić badania kliniczne czy eksperymenty medyczne. Mają one służyć przede wszystkim leczeniu, zastosowaniu nowoczesnego leczenia u osób, które cierpią na bardzo skomplikowane choroby, choroby rzadkie.

Jest to niejednokrotnie szansa na uratowanie życia osobom, dla których dotychczas nie wynaleziono odpowiedniego leczenia.

Jedyną zmianą odnośnie do środków finansowych jest uelastycznienie wydatkowania środków przez Agencję Badań Medycznych.

Dodam jeszcze, co bardzo istotne, że te środki muszą być wydatkowane na ten konkretny cel, na który zostały przeznaczone pierwotnie. Agencja nie będzie miała możliwości zmiany celu wydatkowania środków, a więc zostają zachowane pierwotne założenia, pierwotne cele. Tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy beneficjenci nie zdążą zrealizować zadania, środki zostaną przesunięte na kolejny rok. Środki na inwestycje w Agencji Badań Medycznych będą przeznaczane z dotacji celowej, czyli będzie ściśle określony cel wydatkowania tych środków. Środki te pochodzą z budżetu państwa, a nie z odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby Agencja Badań Medycznych sprawnie funkcjonowała, musi posiadać chociażby systemy informatyczne czy sprzęt komputerowy.

Jeżeli chodzi o pozostałe przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu, podkreślam, że wszystkie samorządy zawodowe są z nami w stałym kontakcie i mają świadomość wprowadzanych zmian.

Dotychczas emitentem były samorządy, które decydują o nadaniu prawa wykonywania zawodu, jak również wydają prawo wykonywania zawodu. Zawsze było to ich zadanie własne.

Jest to o tyle istotne, że dokumenty te będą wydawane już od 1 stycznia i muszą spełniać wymogi określone w ustawie, przede wszystkim związane z brakiem możliwości ich sfałszowania czy wykorzystywania przez niewłaściwe osoby.

Otóż protesty będą składane w przypadku negatywnej oceny wniosku o finansowanie badania. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy ktoś odwołuje się np. od tego, że otrzymał zbyt mało środków.

Podkreślając ponownie rolę Agencji Badań Medycznych w rozwoju terapii lekowych, innowacyjnych leków oraz innowacyjnych terapii leczenia, należy jak najbardziej wspierać agencję, zwłaszcza że jest ona bardzo dobrze oceniana. Raport NIK nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Raport NIK nie weryfikuje jedynie analizy finansowej, ale weryfikuje także wszystkie procedury, które są stosowane w agencji. Tak więc należy podkreślić, że projekty są wybierane w sposób rzetelny, transparentny, obiektywny, zgodnie z przyjętymi procedurami, które są opisane na stronie internetowej, w dokumentacji konkursowej przez osoby, które są bezstronne w procesie, nie mają żadnych powiązań z wnioskodawcami.

Jest również niezbędna opinia komisji bioetycznej, więc wszystko jest realizowane zgodnie z zasadami i przepisami. Ale przepraszam bardzo, pani minister nie wymieniała żadnego nazwiska, więc nie widzę trybu. w jakim trybie? To proszę podać, bo nie znam takiego. Szanowni państwo, projekt jeszcze będzie procedowany w komisji. i zawsze będzie szansa na dopytanie. Zamykam dyskusję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem przedstawić sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, druk nr 1231.

Komisja wnosi o to, ażeby projekt ten został uchwalony.

W związku z powyższym wnosimy, ażeby Wysoka Izba uchwaliła przedłożony projekt nowelizacji po poprawkach. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Kazimierz Smoliński. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość wobec poselskiego projektu zmiany ustawy o partiach politycznych, druk nr 1231. Wysoki Sejmie! Ustawa o partiach politycznych jest z 1997 r. i w niektórych aspektach nie przystaje do aktualnego stanu prawnego. Dlatego posłowie wnioskodawcy stwierdzili, że należy dokonać zmiany art. 18 tej ustawy, który zakłada jawność ewidencji partii politycznej, co jest ze wszech miar potrzebne, natomiast elementy tej jawności idą za daleko. Ta ewidencja jest jawna w zakresie adresów zamieszkania osób, które wchodzą w skład władz partii oraz osób, które są uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu partii, a także adresów na listach osób, które są założycielami, popierają założenie partii. Dlatego projekt ingeruje w tę ustawę i wykreśla możliwość ujawniania tych danych.

To jest właśnie ta zmiana, która mówi o tym, że ewidencja wraz z tekstami statutów partii jest jawna, z wyłączeniem informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, i to zarówno tych osób, które wchodzą w skład organów uprawnionych, jak również osób zgłaszających partię do ewidencji. Zmieniono również zapis, który jednoznacznie stwierdza, że jawne informacje zawarte w ewidencji podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej sądu, w przypadku czego zdaniem prawników rzeczywiście wcześniej nie było podstaw prawnych wprost, dlatego uzupełniono projekt w tym zakresie. On zdaniem klubu Prawo i Sprawiedliwość zasługuje na poparcie i będziemy go popierać, ponieważ te zmiany są naszym zdaniem konieczne, aby chronić te dane osobowe, które nie powinny podlegać ujawnieniu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak jak przedstawił to pan poseł Mularczyk, projekt ustawy nie wzbudza kontrowersji o tyle, że wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom, bo nie dość, że zostaje uregulowana kwestia jawności adresów zamieszkania osób, które są uprawnione do reprezentowania partii politycznych i zaciągania zobowiązań, a pamiętajmy, że to są też osoby, które nie muszą być jednocześnie osobami publicznymi, które nie muszą być aktywnymi politykami, więc jest to zmiana, której kierunek jest dobry, to jeszcze zostają też jednocześnie wprowadzone pewne takie kwestie porządkowe dotyczące jawności, dotyczące publikacji chociażby dokumentów dotyczących partii politycznych. A więc Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego projektu ustawy. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jawności i uczciwości w życiu publicznym potrzeba nam jak przysłowiowego dżdżu. Poziom zaufania społecznego jest w Polsce dramatycznie niski, niższy od średniej europejskiej. Obserwujemy już negatywny kapitał społeczny, negatywne zaufanie objawiające się w nasilającej się korupcji i klientelizmie. Statystyczny Polak zakłada brak dobrej woli po stronie instytucji państwa i po stronie jego przedstawicieli. Nie ufamy ani państwu, ani parlamentowi, ani partiom. Nie wiem, czy państwo czytacie Fukuyamę czy Rothsteina, może chociaż Sztompkę, nie wiem, czy w postępującym braku zaufania, zgeneralizowanego, instytucjonalnego, dostrzegacie kryzys podstaw demokracji, ale na pewno przeglądacie wyniki badań opinii publicznej i oglądacie relacje z polskich ulic, gdzie okrzyki kierowane wobec polityków, zwłaszcza wobec polityków partii rządzącej, wskazują na niski kapitał społecznego zaufania, a od frustracji tylko krok do eskalacji przemocy. Ubiegłoroczne badanie CBOS na temat zaufania społecznego pokazało, że 3/4 społeczeństwa wyznaje pogląd, że w relacjach z innymi ludźmi należy być bardzo ostrożnym. Co ciekawe, najbardziej nieufny wobec innych jest wasz elektorat, a największe zaufanie do innych mają ludzie o lewicowym światopoglądzie. Wiem, że żerujecie na nieufności waszego elektoratu, ale Polska jest częścią Europy i tęskni za tym, co tak pięknie opisał kiedyś Kapuściński - za Europą, czyli światem pozbawionym cwaniactwa, opryskliwości, chamstwa i właśnie wrogiej nieufności. Także wasz prawicowy elektorat tęskni za tą europejską normą. To było widoczne tu, na tej sali dzisiaj, kiedy przegraliście głosowanie, bo posłowie chcieli pełnej informacji o interesach pana Obajtka. Dostrzegacie zbliżającą się klęskę wyborczą, bo Polacy mają dość kumoterstwa i obsadzania rodzinami i znajomymi królika spółek Skarbu Państwa i wszelakich rad nadzorczych. Ponieśliście klęskę propagandową, bo ani ordynarne tyrady na sali plenarnej, ani wszystkie media tzw. publiczne nie dały rady poszczuć jeszcze bardziej obywateli na znienawidzone przez was instytucje. Ponad dwa razy więcej Polaków ufa Unii Europejskiej niż polskiemu parlamentowi.

Ludzie śmieją się z tych żałosnych wpadek typu pana Bielana, który za siedzibę własnej partii obrał biuro poselskie lewicowej posłanki. Paradoksalnie więc dobrze, że chcecie, by niejawne stały się adresy kluczowych członków partii politycznych, bo to zakończy ten lumpiarski zwyczaj szukania słupów, ale likwidowanie zapisów generujących nadużycia i kombinatorstwo nie wystarczy, bo dostęp do informacji o państwie, partiach i sposobie zarządzania mieniem wspólnym trzeba poszerzać, a nie ograniczać. Złożyłam w imieniu Lewicy stosowny projekt ustawy. Kolejne projekty przyniesione przez stronę społeczną czekają w sejmowych zamrażarkach. Ustawę o partiach politycznych trzeba zmieniać w wielu aspektach. Partie nie mogą być trampolinami do żerowania na majątku publicznym. Partie nie mogą być bytami mafijnymi. Tu przypominam wam przegrany proces z prof. Sadurskim, który zdiagnozował PiS-owski styl uprawiania partyjnej polityki. Lewica chce dalszego procedowania nad tym projektem i chce jego poszerzenia o zapisy gwarantujące, że Polacy będą mogli na powrót zaufać swojemu państwu, swojemu parlamentowi, drugiemu człowiekowi, a do tego jest potrzebna jawność i uczciwość, bo bez tego kolejne miliony wyjadą z kraju, a ostatni zgasi światło na tym padole frustracji, nienawiści i traktowania drugiego człowieka jako potencjalnego źródła zła i zarazy. Panie Pośle Mularczyk! Do dzieła. Teraz czas, by przyjął pan uwagi opozycji czy Lewicy, także wnioski mniejszości. Niech zostanie po was coś dobrego, choć jedna rzecz zrobiona dla dobra kraju i jawności, a nie dla dobra partyjnych kolegów i koleżanek. Pani poseł, czasami warto przeczytać projekt ustawy i do niego się odnosić. Pan poseł Dariusz Kurzawa w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści zaprezentować nasze stanowisko w sprawie zmiany ustawy o partiach politycznych, druki nr 1231 i 1256. Chodzi m.in. o nazwę partii, datę założenia, symbole, nazwiska i adresy założycieli oraz reprezentantów i inne istotne informacje. Zmiana polega przede wszystkim na wpisaniu do art. 18 ust. 1 zapisu o jawności wspomnianej ewidencji, z wyłączeniem informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych. Proponowane zmiany w ustawie są naszym zdaniem uzasadnione. Wrażliwe dane osobowe, do jakich należy bez wątpienia adres zamieszkania, są chronione w wielu postępowaniach i dokumentach. Ta sama zasada powinna również mieć zastosowanie w ustawie o partiach politycznych. Powszechne udostępnienie danych adresowych w Internecie jest niebezpieczne i stwarza duże zagrożenie dla sfery prywatnej polityka i jego najbliższych. Posłowie i senatorowie są chronieni w tej sferze w ustawie o wykonywaniu mandatu, a w drugiej, tj. o partiach politycznych, tej ochrony już nie ma. Przytaczany, również w uzasadnieniu, argument o brutalizacji życia publicznego jest trafny, ale chciałbym nieśmiało przypomnieć, że do tej brutalizacji doszło zwłaszcza w ostatnich 5 latach za sprawą mediów publicznych i niektórych najważniejszych osób w naszej polityce. Tym niemniej proponowane zmiany w tej ustawie są konieczne i pożyteczne oraz wspierane przez wielu legislatorów. Dlatego mój klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści popiera wspomniane zmiany i będzie głosować za. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Wysoka Izbo! Zanim przejdę do omówienia tego projektu, projektu zawartego w druku nr 1231, pozwolę sobie na parę słów wstępu. Byłabym wdzięczna, pani marszałek, gdyby pani nie cenzurowała mojej wypowiedzi, bo mam prawo do tego, żeby sformułować ją w dowolny sposób.

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Otóż mamy dzisiaj w Polsce wiele problemów, np. suszę. Dzisiaj rolnicy mówią o tym, że za chwilę będzie tragedia. Służby mówią o tym, że chwilę zaczną płonąć lasy. Dla pana prezesa Glapińskiego nie jest to ważne, co za każdym razem podkreśla w swoim wystąpieniu. Mamy problem przemocy. Mamy problem braku usług publicznych na poziomie odpowiadającym naszemu rozwojowi i naszym aspiracjom. Kolejki do lekarza zagrażają życiu ludzkiemu. Można byłoby długo mnożyć tematy, którymi powinien zajmować się polski Sejm. Mogłabym wymieniać przez 5 minut listę tylko tych tematów, którymi się polski Sejm powinien zajmować.

Tymczasem my się zajmujemy adresami polityków.

Załóżmy, że potraktowalibyśmy ten temat poważnie, że chcielibyśmy coś w tych partiach politycznych poprawić. W związku z tym zgłosiliśmy poprawki. Pierwsza poprawka mówi o tym, żeby poza sprawozdaniami finansowymi składać też sprawozdania merytoryczne z działalności partii politycznych.

Ale pan poseł Mularczyk prowadzący prace nad tą ustawą uznał najwyraźniej, że jeśli coś jest wymyślone poza PiS-em, to jest to po prostu myślozbrodnia. Proponuję, żeby pan sobie odświeżył lekturę Orwella, bo naprawdę zbliżacie się państwo już nie tylko do tych postaci, ale do ich karykatur. Zagłosujemy za tą ustawą, ale uważamy, że skandaliczne jest to, że Sejm zajmuje się tak nieważnymi dla ludzi tematami, kiedy ważne tematy nie są zaadresowane.

Wysoka Izbo! Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na pewne kuriozum.

Jest to jakaś absurdalna sytuacja i uważam, że powinniśmy zdecydowanie przemyśleć tryb procedowania, tryb dyskusji nad takimi rzeczami i ustalić, jakie mamy priorytety. Do rzeczy, do rzeczy. Od samego początku zmierzam do rzeczy. Ten poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych jest niekontrowersyjny, bo co miałoby być kontrowersyjnego. I pewnie w takiej formie zostanie uchwalony. Jednak tym, czego naprawdę potrzebujemy, są zmiany systemowe, a tych Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi przygotować, ponieważ nasz skostniały system polityczny trzeba zmienić. My nie mamy, tak jak często to państwo określają, jakiejś demokracji, tylko mamy oligarchię partyjną, gdzie prezesi poszczególnych partii wyznaczają, kto dostanie jedynkę i w związku z tym, kto ma zostać posłem. Trzeba zmienić nasze prawo wyborcze, tak aby realnie posłowie, którzy pracują w swoich okręgach, którzy są znani, mogli mieć możliwość, że zostaną wybrani, bez tego, że będą musieli podlizywać się prezesowi swojej partii. Zdecydowanie ułatwiłoby to życie nam wszystkim.

I na to są potrzebne pieniądze. Jeśli państwo nie wiedzą, z czego to finansować, to bardzo proste, obetnijmy subwencje i dajmy te pieniądze właśnie na ekspertyzy i ekspertów. Bo Polacy od nas oczekują nie wyrażania swoich emocji, tylko merytorycznej pracy dla nich. Takich zmian oczekują wyborcy i takie zmiany przygotuje Konfederacja, a jeśli zostanie wybrana, to również je wprowadzi. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Pani Marszałek! Mój przedmówca, poseł Krystian Kamiński, słusznie zwrócił uwagę na to, że mamy w polskiej polityce deficyt środków na pracę ekspercką. Jest to w ustawie o partiach politycznych zdefiniowane, ale myślę, że można dość łatwo zrozumieć, dlaczego tak jest. Otóż odpowiedź tkwi w niechęci do projektu, który przedstawiliśmy już 5 lat temu, i solidarnie wszystkie partie polityczne przestraszyły się, nabrały wody w usta. To był projekt o finansowaniu polskiej polityki i działalności w debacie publicznej z zagranicy. Dziś mainstreamowe partie polityczne od PiS-u przez Platformę po Lewicę, PSL pracują za pieniądze niemieckich fundacji politycznych, robią wspólne projekty, a to tzw. prawica z Fundacją Konrada Adenauera, lewica ma odpowiednie fundacje lewicowe, liberałowie - liberalne, tak zwani centrowcy. W żaden sposób wam to nie przeszkadza. Dlaczego? Bo nie zdecydowaliście się nigdy zmienić prawa w ten sposób, żeby ktoś działalności wywrotowej w Polsce nie mógł finansować. Działalność szpiegowska, jak ktoś przywiezie pieniądze w walizce, jest zakazana, ale jak ktoś przeleje prosto na konto fundacji pani Kozłowskiej, jest całkowicie legalna. Dlatego nie zależy wam na tym, żeby była finansowana działalność ekspercka z funduszy politycznych na partie polityczne, bo macie je skądinąd. A jeżeli chodzi o te kwestie, o których dzisiaj rozmawiamy, wykreślenie publikacji prywatnych adresów, polityków, jest to oczywista sprawa. To pokazuje tylko, jak anachroniczna jest ustawa o partiach politycznych. Ustawy o partiach politycznych nikt nie ruszył. Ta ustawa jest w wielu punktach kompletnie niedopasowana do dzisiejszych czasów. Ona jest swego rodzaju prawnym reliktem. Należałoby zrobić okrągły stół partii politycznych, napisać tę ustawę od początku. Zobaczyć, jak partie polityczne powinny działać nowocześnie w XXI w., gdzie w tej chwili cały szereg narzędzi, które stosuje się współcześnie, związanych z Internetem, z finansami jest skrępowany. Ale wam na tym nie zależy, bo sobie wszystko finansujecie jak nie z Polskiej Fundacji Narodowej (Dzwonek), to ze spółek Skarbu Państwa, to z kancelarii premiera. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Pierwsze pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica.

Pytanie jest związane z ustawą o partiach politycznych. Może pan przewodniczący, gdyby był w stanie, choć pytanie nie należy do łatwych. Czy partie polityczne zgodnie z ustawą mogą posiadać majątek? Czy żeby zamontować na budynku partii politycznej fotowoltaiki, partia polityczna może otrzymać dofinansowanie, które otrzymują inne podmioty na zamontowanie fotowoltaiki, na budynkach będących własnością partii politycznej?

Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo! Po wprowadzeniu tej nowelizacji ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych będzie jawna, natomiast adresy przywódców partyjnych jawne nie będą. Rozumiem, że każda grupa polityczna dba o własne interesy, ale posłowie zgromadzeni na tej sali powinni przede wszystkim zadbać o interesy wyborców, a dopiero później o interesy własne. Utajnienie adresów zamieszkania władz partii, których prezesi mogą swoimi decyzjami zniszczyć życie milionów ludzi, moim zdaniem powinno nastąpić w drugiej kolejności, po utajnieniu adresów członków stowarzyszeń, fundacji, a przede wszystkim przedsiębiorców, z których podatków finansuje się działalność partii. Dziękuję. Pan poseł Marek Dyduch, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Możemy to uregulować. Proponuję, żeby 50% dotacji dla tych partii politycznych, które są w Sejmie, mogło iść na wybory, a 50% zostawić na edukację polityków, na dokształcanie ich, jeżeli chodzi o ekspertyzę, ich wiedzę, ich kulturę polityczną, bo dzisiaj tak naprawdę partie polityczne, które są w Sejmie - i to jest różnica, bo różnicują się w ten sposób, mają preferencje - finansują swoje wybory ze środków państwowych. Zainwestujmy w lepszą jakość uprawiania polityki, bo to jest istota.

Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Oczywiście nie mam absolutnie żadnych uwag do tego projektu ustawy, natomiast mam takie ogólne pytanie dotyczące techniki prawotwórczej, dlatego że już dzisiaj słyszymy na tej sali, że są inne propozycje dotyczące zmian w ustawie o partiach politycznych. Rzeczywiście dość kuriozalne jest to, że prowadzimy tutaj półgodzinną dyskusję i dyskusje na posiedzeniach komisji, żeby zmienić jeden artykuł. Jeżeli są już w przestrzeni publicznej czy parlamentarnej jakieś pomysły dotyczące innych zmian w ramach tej samej ustawy, to wydaje się rozsądne, żeby wstrzymać się z tą ustawą i przyjąć jedną. Nie nowelizować jednej ustawy na każdym posiedzeniu Sejmu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Domyślam się, że na pytania chętnie odpowie pan poseł Arkadiusz Mularczyk jako sprawozdawca komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. Wysoka Izbo! Jestem przedstawicielem wnioskodawców.

To był projekt poselski, nie był to projekt rządowy.

Każdy z klubów ma taką możliwość. Co do tych poprawek, o których wcześniej rozmawialiśmy, pani poseł Muchy, to niestety te poprawki zostały zgłoszone do przedłożenia, które dotyczyło zupełnie innego, incydentalnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o większe, szersze nowelizacje, jesteśmy otwarci.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

Uprzejmie proszę pana posła Grzegorza Lorka o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!

W toku prac komisji odbyła się dyskusja oraz wniesiono poprawki. Przypomnę, że w projekcie przewidziano dodanie w Kodeksie cywilnym zapisów, zgodnie z którymi najbliższej rodzinie poszkodowanego, który np. wskutek wypadku doznał trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie odszkodowanie za naruszenie więzi rodzinnej. Na przestrzeni ostatnich lat w orzecznictwie sądów powszechnych ukształtowało się przeważające stanowisko, że tego rodzaju krzywda podlega naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Stanowisko to zostało potwierdzone orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym kierunkiem judykatury sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. W praktyce sądowej można jednak odnotować przypadki prawomocnego oddalenia powództwa najbliższych członków rodziny poszkodowanego o zapłatę zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej.

Ujawniona rozbieżność i zmiana kierunku rozstrzygania o bardzo istotnych społecznie roszczeniach nie są pożądane z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady zaufania do państwa i tworzonego przez niego prawa. Słuszna jest zapłata zadośćuczynienia, gdy najbliższy członek rodziny doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy pan poseł Grzegorz Lorek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, druk nr 1125. Projekt przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym zapisów, zgodnie z którymi najbliższej rodzinie poszkodowanego, który np. wskutek wypadku doznał trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie odszkodowanie za naruszenie więzi rodzinnej. W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Potrzeba zmian, jak zostało to przedstawione w sprawozdaniu, wynika z rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Ujawniona rozbieżność i zmiana kierunku rozstrzygania o bardzo istotnych społecznie roszczeniach nie jest pożądana z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady zaufania do państwa i tworzonego przez niego prawa. Słuszna jest zapłata zadośćuczynienia, gdy najbliższy członek rodziny dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie rekomenduję ww. projekt ustawy. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Z przyzwyczajenia chciałem powiedzieć: marszałek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt ustawy jest konsekwencją luki prawnej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku zadośćuczynienia pieniężnego za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. W praktyce sądowej w wielu przypadkach zarówno sądy powszechne, jak i Sąd Najwyższy uznawały, że mamy do czynienia z dobrem osobistym, o którym mowa w art. 23 Kodeksu cywilnego, i zasądzały, jeżeli uznały ku temu podstawy, zadośćuczynienie pieniężne, właśnie na podstawie art. 23 Kodeksy cywilnego w związku z art. 448 Kodeksu cywilnego. Były jednak orzeczenia zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, w tym ostatnia uchwała Sądu Najwyższego podjęta w składzie siedmiu sędziów, które wskazywały, że nie ma podstawy prawnej do zadośćuczynienia właśnie w takim przypadku, którego dotyczy przedmiotowy projekt ustawy, i kończyło się to oddaleniem powództwa. Taka sytuacja rozbieżności jest dla obywatela nie do zaakceptowania, powoduje bowiem niepewność prawną, sytuację, w której obywatel nie ma pewności, jak sąd rozstrzygnie konkretną sprawę, w której występuje on z roszczeniem pieniężnym, w tym przypadku z pozwem o zadośćuczynienie pieniężne. Na istnienie luki prawnej wskazywała już w 2018 r. pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani prof. Małgorzata Gersdorf w wystąpieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. Tam właśnie mówiła o tym, że kwestia zadośćuczynienia pieniężnego w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia wymaga regulacji prawnej.

Nie, przepis jest jednoznaczny i mówi o ciężkim i trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia skutkującym niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.

Bardzo dziękuję. Głos ma pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewicy.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie prezydenckiego projektu ustawy z druku nr 1125 oraz sprawozdania komisji o pracach nad projektem z druku nr 1218. W dniu wypadku Katarzyna J. miała 17 lat, była licealistką. Kolega, który prowadził Renault Megane, stracił nad nim panowanie i rozbił się na drzewie, a po tygodniu zmarł. We krwi miał morfinę i amfetaminę. Dziewczyny nie przebadano z uwagi na jej ciężki stan. Doznała rozległych obrażeń, a lekarze ocenili jest stan jako wegetatywny. Od tamtego czasu wymaga całodobowej opieki w każdym aspekcie swojego życia, a szanse na poprawę są nikłe. Edyta B. od chwili wypadku drogowego, w wyniku którego doznała ciężkiego urazu mózgu, znajduje się w stanie głębokiego wyłączenia świadomości, w stanie wegetatywnym. Nie ma możliwości nawiązania z nią kontaktu, została ubezwłasnowolniona całkowicie, a przy obecnym stanie wiedzy medycznej nie jest możliwa poprawa jej stanu zdrowia. W dniu wypadku miała 34 lata, była mężatką, matką 6-letniego syna. Pracowała jako lekarka, dermatolożka, pisała pracę doktorską. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców. Młoda matka samotnie wychowująca dzieci w wieku 3 i 4 lat na skutek błędu medycznego doznaje obrzęku mózgu, a następnie pozostaje w utrwalonym stanie wegetatywnym. W świetle opinii biegłych strata matki destrukcyjnie wpływa na rozwój psychiczny dzieci, prowadząc do trudności adaptacyjnych, emocjonalnych, uczuciowych.

Postępowania trwały latami, a rozstrzygnięcia bywały różne. A przecież w takich sytuacjach nie można czekać, nie można i nie trzeba. Nie trzeba czekać na wybudzenie osoby w śpiączce, by stwierdzić, że ona i jej najbliżsi cierpią. Nie trzeba i nie można czekać, by za to cierpienie zadośćuczynić. Członkowie rodziny, których bliscy zapadają w śpiączkę pourazową czy stan wegetatywny, cierpią często nie mniej niż w momencie, gdy bliska im osoba umiera. Dlatego takie zadośćuczynienie musi wprost gwarantować prawo. Przyznanie zadośćuczynienia członkom rodziny poszkodowanego ma być możliwe w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego zerwaniem lub niemożnością nawiązania więzi rodzinnych. Wprowadzenie takiej zmiany przewiduje niniejsze przedłożenie. Proponowana zmiana przepisów ma pomóc w rozstrzygnięciu rozbieżności orzeczniczych, które pojawiły się w ostatnich latach, i to na poziomie zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. Obecnie w Kodeksie cywilnym wprost umożliwia się sądowi przyznanie najbliższym członkom rodziny odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jedynie w przypadku osoby bliskiej zmarłej wskutek czynu niedozwolonego. W praktyce problemy związane z przyznawaniem członkom rodziny zadośćuczynień zaczynają się w momencie, gdy dana osoba doznaje ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Dlatego w projekcie zaproponowano, by podstawa prawna normatywna tego typu rozstrzygnięć została wyrażona wprost w dodanym art. 446 Kodeksu cywilnego. Jak wskazano w uzasadnieniu, przepisy miałyby zastosowanie jedynie do przypadków najcięższych, właśnie takich jak zerwanie więzi rodzinnych w wyniku śpiączki pourazowej, stanu wegetatywnego czy stanów związanych z uszkodzeniem mózgu. Choć nie sposób wycenić czy wartościować cierpienie i krzywdę, to wypłata zadośćuczynienia w takich sytuacjach powinna być możliwa, a możliwość ta powinna być gwarantowana przez prawo. Co ważne, przedmiotowa nowelizacja może mieć zastosowanie nie tylko do zdarzeń, które nastąpiły dopiero po zmianie przepisów.

Ze względu na znaczenie społeczne problemu, z uwagi na fakt, że w toku prac komisji nie zostały wprowadzone zmiany, które zmieniłyby zamysł wnioskodawcy wyrażony w przedłożonym projekcie, klub Lewicy podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w pierwszym czytaniu i uważa, że powyższe rozwiązania zasługują na poparcie. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Krzysztof Paszyk w imieniu Koalicji Polskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści chciałbym przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania komisji o przedstawionym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, druki nr 1125 i 1218. Klub Parlamentarny Koalicja Polska, tak jak i kluby prezentujące swoje stanowiska przed naszym klubem, jest jak najbardziej pozytywnie nastawiony do prezydenckiego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego polegającego na dodaniu art.

Do takich zdarzeń na pewno możemy zaliczyć stan wegetatywny, śpiączkę lub ciężkie uszkodzenie mózgu. Ocena, czy zaszły przesłanki do przyznania zadośćuczynienia, czy nie, w razie sporu będzie leżała w gestii sądów, a można by pokusić się o zamknięty katalog takich sytuacji. Ponadto regulacja powinna być tak skonstruowana, by członkowie rodziny z góry wiedzieli, na jaką wypłatę mogą liczyć w danej sytuacji. Bez takiej regulacji zadośćuczynienia pozostaną w dużym stopniu nieprzewidywalne. W bardzo podobnych przypadkach orzekane zadośćuczynienia różnią się między sobą nawet cztero-, pięciokrotnie. Wątpliwości budzi też sformułowanie: trwały uszczerbek na zdrowiu, które nie ma prawnej definicji. W uzasadnieniu do nowelizacji jest użyte określenie: nieodwracalne upośledzenie funkcji życiowych, a to określenie znacznie lepiej oddaje charakter regulowanej kwestii. Pozostaje również pytanie, który podmiot będzie uprawniony do stwierdzenia, że stan poszkodowanego jest trwały w rozumieniu nieodwracalności upośledzenia funkcji życiowych. Nie wiadomo też, co będzie się działo w przypadku, gdy najbliżsi członkowie rodziny otrzymają zadośćuczynienie z tytułu zerwania więzi rodzinnych, a następnie osoba poszkodowana umrze. Art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przyznaje zadośćuczynienie bliskim z tytułu śmierci. Proponowany przepis nie rozstrzyga relacji między wymienionymi przepisami. Ubezpieczyciele obawiają się, że najbliżsi członkowie rodziny będą mogli dwukrotnie zgłaszać roszczenie. To są wątpliwości, które oczywiście pozostają.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

Po prostu szkoda.

To nie stawia niestety naszego sądownictwa czy powagi państwa polskiego w najlepszym świetle.

Jest jedynie możliwość dialogu czy właśnie to załatwianie spraw dla Polaków.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Wysoki Sejmie! Pani Minister! Koło Parlamentarne Polska 2050 po raz kolejny wyraża poparcie dla projektu tej ustawy. Dobrze, że pojawia się propozycja prawnego rozwiązania zapłaty zadośćuczynienia, kiedy najbliższy członek rodziny dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Ma na myśli szczególnie dramatyczne sytuacje, kiedy w następstwie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest już możliwe występowanie więzi rodzinnej. Istotne będzie jednak określenie, co jest więzią rodzinną i między kim ona rzeczywiście występuje. Koło Polska 2050 proponuje nie rewolucyjną, ale ewolucyjną, nowoczesną zmianę. Upieramy się: postawmy odważnie krok. Nowoczesne demokracje według nas tego wymagają.

Zwracamy uwagę, że Sąd Najwyższy wskazał w wyroku z 21 marca 2013 r., że w każdym przypadku osób wspólnie zamieszkujących ze sobą możliwe jest występowanie takiej więzi emocjonalnej, która uzasadni przypisanie im statusu osób najbliższych. Są i tacy przedstawiciele doktryny - ponownie podkreślamy - którzy uważają, że do rodziny w rozumieniu przepisu art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego należy też zaliczyć wychowanków, narzeczonych, konkubentów, jeżeli ich związek ma charakter dostatecznej trwałości i cechuje się dostatecznie silną wspólnością gospodarczą. Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera projekt. Uważamy za słuszne przyznanie zadośćuczynienia, ale rzeczywiście osobom najbliższym poszkodowanemu, z którym nie występuje już więź. Dlatego składamy tę poprawkę. Pamiętamy słowa pani minister wyrażone tutaj, w Sejmie, o poszanowaniu i równości prawa.

Do pytań zgłosiło się dwoje państwa posłów, właściwie dwóch panów posłów.

Panie Marszałku! Rodzina, więzi rodzinne to podstawa naszego życia.

To nie tylko ta sprawa, to również ustawa o usługach płatniczych. Ale ta konkretna ustawa, mówiąca o więziach rodzinnych, jest niezbędna, jest potrzebna i daje ona sądom jednoznaczne możliwości w zakresie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia. Pytanie zadaje pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Pani Minister! Wysoka Izbo! Zalegalizowana formalnie rodzina jest tylko jednym ze związków, w których ludzie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ustawa zatem powinna jednak szerzej traktować grono osób uprawnionych do wypłat wspomnianej rekompensaty. Powinny być to osoby zaliczone do grona osób najbliższych poszkodowanemu, a nie tylko członkowie jego rodziny. Więzi międzyludzkie stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania każdego związku, w tym również rodziny. Nagłe zerwanie tych więzi powinno być łagodzone przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia, ale ustawa ta powinna jednak szerzej traktować grono osób do tego uprawnionych. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych. Bardzo proszę, pani minister.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Należy podziękować panu prezydentowi za tę inicjatywę ustawodawczą. Nie będę chyba w tej opinii odosobniona, zresztą to już wybrzmiało na tej sali, jak ważny jest to projekt, jak uzupełnia on lukę prawną istniejącą w naszym systemie prawa. W obecnym bowiem stanie prawnym brak jest jasnej, jednoznacznej regulacji, która stanowiłaby podstawę prawną przyznania najbliższym członkom rodziny bezpośrednio poszkodowanego zadośćuczynienia w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego odniósł on ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu, skutkujący niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym. Chciałabym zaznaczyć, że to jest bardzo ważny projekt ustawy, w związku z powyższym nie ma żadnych wątpliwości, że Wysoka Izba powinna go przyjąć. Bardzo dziękuję, pani minister. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani minister.

Wysoka Izbo! Pozwolą państwo, że na początku wyrażę w imieniu pana prezydenta podziękowanie za jednogłośne, jednolite poparcie dla prezydenckiej inicjatywy nowelizacji Kodeksu cywilnego.

Pan poseł Paszyk, deklarując poparcie dla prezydenckiej inicjatywy, zwrócił uwagę na kilka kwestii, m.in. brak katalogu zdarzeń uzasadniających uzyskanie zadośćuczynienia, padały pytania o wysokość zadośćuczynienia, o organ, który miałby oceniać stan poszkodowanego. Te kwestie były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia komisji i króciutko odniosę się do tego. Z pełną świadomością, mając przede wszystkim na uwadze fakt, że są to regulacje Kodeksu cywilnego, a więc systematykę Kodeksu cywilnego, brak definicji legalnych, a także doprecyzowywanie i wykładnie tych przepisów w drodze orzecznictwa sądowego, w tym w szczególności orzecznictwa Sądu Najwyższego, w ocenie urzędu prezydenckiego brak jest możliwości utworzenia zamkniętego katalogu zdarzeń.

Po stronie sądów w ocenie urzędu prezydenckiego powinna być zarówno kwestia wysokości zadośćuczynienia, jak i ocena stanu poszkodowanego, chociażby ze względu na mechanizmy, którymi sam dysponuje, np. możliwością skorzystania z fachowej wiedzy biegłych. Pan poseł Zimoch, ale to również wybrzmiało w pytaniu pana posła Szopińskiego, podnosi kwestie zmiany katalogu osób uprawnionych, czyli wraca propozycja zmiany sformułowania „najbliższy członek rodziny” na „osobę najbliższą” Ta kwestia była dyskutowana zarówno podczas pierwszego czytania, jak również podczas posiedzenia komisji i pragnę państwa zapewnić, że była to kwestia również bardzo dokładnie sprawdzana i analizowana w Kancelarii Prezydenta.

Przede wszystkim ewentualne zastąpienie sformułowania „najbliższy członek rodziny” sformułowaniem „osoba najbliższa” spowodowałoby rozróżnienie katalogu osób uprawnionych do zadośćuczynienia w przypadku stanów wegetatywnych, o których mówimy w tym przepisie, projektowanym i proponowanym przez pana prezydenta, a sytuacją zadośćuczynienia w przypadku śmierci. I to katalog w przypadku tych stanów wegetatywnych byłby w takiej sytuacji szerszy. Po drugie, w tych sprawach mówimy o braku możliwości nawiązania czy kontynuowania więzi rodzinnych i ze względu właśnie na ochronę więzi rodzinnych wydaje się, że to sformułowanie „najbliższy członek rodziny” jest najbardziej odpowiednie, a - proszę pozwolić - tylko na podstawie analizy orzecznictwa, o której wspominałam, ten katalog jest dość szeroko rozumiany przez sądy i wchodzą w to małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, przyrodnie rodzeństwo, w niektórych przypadkach dziadkowie, konkubenci, powinowaci.

Wydaje mi się, że to wszystko. Jeszcze raz, Wysoka Izbo, dziękuję za jednolite poparcie prezydenckiej inicjatywy. Bardzo dziękuję, pani minister. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 1090 i 1210) Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z druku nr 1090. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 25 marca br. jako inicjatywa Komisji Ustawodawczej. W dniu 20 maja na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, a następnie pani marszałek skierowała projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a ta z kolei skierowała projekt do swojej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Podkomisja po kilku godzinach pracy w dniu 8 czerwca przyjęła sprawozdanie zawierające wniosek o przyjęcie projektu w formie tekstu jednolitego projektu z wniesionymi poprawkami, który to projekt został w dniu następnym przyjęty przez komisję, i załączone jest do sprawozdania komisji przedstawionego w druku nr 1210. Wysoka Izbo! Proponowana nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. wydanego w sprawie pod sygnaturą akt P46/13, w którym przesądzono, że art. 156 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowe jest, że przywołany wyżej wyrok jest wyrokiem zakresowym, odnoszącym się do wąskiego zagadnienia przedstawionego trybunałowi. W związku z tym w ramach swoich prac Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach uznała za zasadne zajęcie się szerszym wymiarem przedstawionego przez sąd konstytucyjny problemu, w sposób zapewniający równowagę pomiędzy konstytucyjnymi zasadami legalizmu oraz pewności prawa. Podczas posiedzeń podkomisji i komisji, po rozważeniu szeregu poprawek, zdecydowano o dodaniu sytuacji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2, w której doszło do wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, do dotychczasowego katalogu okoliczności, w których stwierdzenie nieważności jest możliwe w okresie do 10 lat od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, a po upływie którego stwierdza się wyłącznie wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Przyjęto też poprawkę wprowadzającą do projektu nowy, 30-letni termin na rozpatrywanie spraw dotyczących nieważności decyzji, po upływie którego wniosek w tym przedmiocie stanie się niedopuszczalny i zostanie przez organ odrzucony. Na skutek proponowanej regulacji co do decyzji wydanych w okresie pomiędzy 10 a 30 lat wstecz będzie więc możliwe uzyskanie stwierdzenia organu o wydaniu zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa, ale decyzja nie będzie mogła być uchylona. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego wynika wprost, że nieograniczona w czasie wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych nie jest zasadą konstytucyjną, a ograniczenie terminów zaskarżania prawomocnych decyzji administracyjnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa prawnego. Z klauzuli państwa prawnego wynikają bowiem w szczególności zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasada bezpieczeństwa prawnego, które mają dla ustawodawcy charakter wiążący. W związku z powyższym, jak również oceniając wagę zagadnienia, komisja uważa za konieczne wprowadzenie też regulacji międzyczasowych zawartych w treści art. 2. Niewątpliwie bowiem zmiana regulacji objętych projektem odniesie bezpośredni skutek dla szeregu postępowań pozostających na biegu w dniu wejścia w życie ustawy. W tym stanie rzeczy zadaniem ustawodawcy jest przewidzenie rozwiązania gwarantującego uzyskanie merytorycznego rozstrzygnięcia podmiotom, które przed upływem 30 lat od wydania kwestionowanej przez siebie decyzji skorzystały z możliwości jej zaskarżenia, a do wejścia w życie ustawy nie uzyskały jeszcze rozstrzygnięcia - niezależnie od tego, że do tego czasu minie 30 lat od daty wydania kwestionowanego orzeczenia. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie stabilności systemu prawnego poprzez jego zabezpieczenie przed zalewem wniosków wyłącznie dla skorzystania z obwiązującej obecnie regulacji i niezależnie od merytorycznych podstaw do ich złożenia. Stąd też uznano za zasadne, aby wszelkie postępowania wynikające z zaskarżenia decyzji po upływie ponad 30 lat od jej wydania uległy umorzeniu z mocy prawa. Niewątpliwie termin 30 lat pozostaje w polskim systemie prawnym jednym z najdłuższych terminów powodujących określone ustawami skutki prawne, takie jak choćby możliwość nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Znamienne jest, że okres przedawnienia roszczeń cywilnych wywołanych zbrodnią lub występkiem ustalony został na 20 lat. Stąd też zakreślenie 30-letniego terminu dla dochodzenia praw w drodze administracyjnych postępowań nadzwyczajnych przez podmioty zainteresowane będzie realizowało zasady państwa prawnego i praworządności, dając równocześnie podstawę dla trwałości wydanych orzeczeń. Podczas prac komisyjnych wydłużyliśmy też vacatio legis z proponowanych 14 dni do standardowo przyjętych przy nowelizacjach kodeksów 30 dni i proponujemy, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym podziękować wszystkim członkom naszej komisji i ministerstwu, ministerstwom za sprawną oraz merytoryczną pracę. W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wnoszę, aby Wysoki Sejm uchwalił projekt ustawy zawarty w druku nr 1210. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza pani poseł Barbara Bartuś w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypadł mi zaszczyt i przyjemność przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawartym w druku nr 1210. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ramach prac poselskich niejednokrotnie przychodzi nam mierzyć się z zagadnieniami, w których nie ma miejsca na podejście minimalistyczne i konieczne jest szersze spojrzenie na analizowany problem prawny - po to, aby tworzone prawo nie było martwe i aby przede wszystkim skutecznie służyło interesowi publicznemu i interesowi obywatela. Taka sytuacja niewątpliwie wyłoniła się w trakcie prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Reguła trwałości decyzji służy realizacji istotnych wartości, jakimi są ochrona porządku prawnego, stabilności obrotu prawnego, zaufania do organów państwa i samego prawa, a przede wszystkim - ochrona praw nabytych. Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego wszelkich decyzji, zwłaszcza wydanych przed kilkudziesięciu laty, niesie za sobą ogromne ryzyko, zarówno ze względu na rosnące trudności dowodowe, jak i problem dotyczący braku dostępu do akt spraw pierwotnych. Często decyzje o stwierdzeniu nieważności są wydawane uznaniowo, w oparciu o wybrakowany materiał dowodowy i bez możliwości dokonywania pogłębienia analizy faktycznego stanu prawnego. Pamiętajmy, że obowiązują nas przepisy o brakowaniu akt. Nie bez znaczenia pozostają również potencjalne zmiany w wykładni przepisów prawa oraz ocenie zdarzeń ze sfery faktycznej, które stały u podstaw wydawanego rozstrzygnięcia. Sytuacje takie, zamiast doprowadzać do stanu zgodnego z prawem, rodzą faktyczne zagrożenie naruszenia interesu prawnego zarówno podmiotów indywidualnych, jak i społeczności różnego szczebla.

W tym czasie niewątpliwie nie istniały przeszkody w dochodzeniu swoich praw na podstawie obowiązującej obecnie regulacji. Dlatego też proponowany krańcowy czas na podjęcie działań zmierzających do uchylenia skutków prawnych wadliwych orzeczeń administracyjnych ocenić należy jako wystarczający, zwłaszcza wobec obserwowanego rozwoju form komunikacji oraz powszechnego dostępu do informacji, w tym informacji prawnej. Zaznaczam przy tym, że ewentualne odniesienia do instytucji zasiedzenia i przedawnienia nie mają tu wymiaru analogii, a stanowią wyłącznie zwrócenie uwagi na przyjęte przez ustawodawcę okresy wywołujące daleko idące skutki prawne. Skoro po upływie 30 lat możliwa jest ingerencja w prawo własności, które to prawo wskazywane jest jako najsilniejsze prawo majątkowe, to przyjęcie takiego samego terminu do możliwości kwestionowania rozstrzygnięć administracyjnych - nie zawsze wywołujących skutek rzeczowy - musi być uznane za racjonalne i wyważone. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako ustawa zasadnicza ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w naszym państwie. Podstawowym skutkiem wejścia w życie projektowanych regulacji będzie uzupełnienie regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która nie spełnia wymogów konstytucyjnych, o rozwiązanie prawne, które w należytym stopniu będzie odzwierciedlać wnioski płynące z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość deklaruję poparcie dla zaprezentowanej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wobec projektowanej zmiany ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego przedstawionej w drukach nr 1090 oraz nr 1210. Chciałabym przekazać, że merytoryczne rozwiązania przedstawione w tym projekcie nie budzą w zasadzie wątpliwości. Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., który stwierdził niezgodność art. 156 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z konstytucją. Trybunał orzekł, że przywołany artykuł w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W konkluzji wyroku Trybunał podniósł, że stabilizacja stanów faktycznych po upływie określonego czasu leży w interesie porządku publicznego i w tym pozostajemy zgodni.

Pierwsze dotyczy tego, że do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Drugie zastrzeżenie dotyczy krótkiego terminu wejścia w życie ustawy.

Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Wobec niepodjęcia przez ustawodawcę stosownych działań legislacyjnych w reakcji na ww. wyrok orzecznictwo sądowe od blisko 6 lat mierzy się z problemem dopuszczalności i sposobu jego uwzględniania w konkretnych sprawach administracyjnych. Mierzy się ono z jednej strony z problemem braku bezpośredniego skutku prawotwórczego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony - z potrzebą zapewnienia zgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ochrony prawnej dla podmiotów, które znalazły się w sytuacji podobnej, analogicznej do tej, która stanowiła kanwę wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jak podkreślają eksperci, to niezwykle ważna zmiana dla administracji publicznej, dla obywateli zainteresowanych decyzjami chociażby wywłaszczeniowymi. Gdyby zaczął obowiązywać przepis, który został zaproponowany w projekcie, nieważność wydanych decyzji zostałaby wyłączona.

Należy jednak zapytać o ten czas, który upłynął od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Należy również zapytać, co takiego spowodowało tak gruntowne przeformułowanie pierwotnych zapisów projektu na etapie prac komisji, z którym mieliśmy do czynienia.

Bo co np. z tymi sprawami, które są w toku?

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Dobra: że pan naszą poprawkę i nasze działanie w komisji zauważył. Zła, bo myślał pan, że dzisiaj nie złożymy poprawki. Ale by nie powtarzać tego, co już zostało powiedziane, proponujemy skrótowo, czyli: mini, maks - minimum słów, maksimum dobrego prawa.

Przyjęto bowiem bardzo długi, bo aż 30-letni, termin na wzruszenie decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa, które były podstawą nabycia prawa lub stwarzały uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa.

Proponujemy zatem, aby wprowadzić w tym przypadku właśnie termin 10-letni, taki sam jak w przypadku innych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji z art. 156 k.p.a. Wydaje się, że wprowadzenie tak długiego terminu nie wypełnia intencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dążył do kompromisu między zasadami legalizmu a zasadą zaufania obywatela do państwa. Termin 30-letni przyznaje ewidentnie w dalszym ciągu zdecydowany prymat zasadzie legalizmu, skoro pozwala wzruszać decyzje zapadłe pokolenie wcześniej. Podważanie takich decyzji niemal zawsze będzie prowadziło do pogłębiania się chaosu prawnego i konieczności kaskadowego unieważniania kolejnych czynności prawnych podejmowanych już wiele lat temu, często przez osoby fizyczne już nieżyjące lub osoby prawne już nieistniejące. Dlatego na ręce pana marszałka zgłaszamy poprawkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj debatujemy o koniecznym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Co do proponowanych zmian, są one potrzebne, wynikają zresztą z konieczności implementacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do systemu prawa. Ale nie można ich przyjąć w takiej formie. Zaproponowane zmiany wykraczają daleko poza sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa, dotyczących nabycia prawa lub ekspektatywy. W tym projekcie zostały one rozciągnięte również na decyzje wydane bez podstawy prawnej lub wydane z rażącym naruszeniem prawa, niebędące jednocześnie podstawą nabycia prawa bądź jego ekspektatywy. Ponadto w zaproponowanym kształcie ustawa zakłada umorzenie z mocy prawa toczących się już postępowań - wszczętych po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Zapis ten w istocie narusza art. 2 konstytucji, którego naruszenie dotyczyło wydanego przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia. Wątpliwości budzi również stosunkowo krótki, bo 10-letni, termin umożliwiający uzyskanie przez wnioskodawcę nieważności decyzji administracyjnej, co jest istotne w związku z powszechnie występującą przewlekłością postępowań. Mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie, jak również wadliwość zaproponowanych rozwiązań, a także możliwość uznania ich za niekonstytucyjne, jako Konfederacja jesteśmy zdziwieni i mamy nadzieję, że zostaną one naprawione. W tym aspekcie, w aspekcie tej nowelizacji, warto jeszcze powiedzieć o jednym skandalicznym i oburzającym fakcie: przedstawiciel dyplomatyczny nie najwyższej rangi innego państwa strofuje panią marszałek, poucza, jak my w Polsce mamy kształtować naszą legislację. Nie jesteśmy kolonią amerykańską, nie jesteśmy 51. stanem.

Gdyby tak nie było, toby się tym tematem nie zajmował, a przypominam, że obywatelski projekt ustawy jest w komisji i nie chcą państwo nad nim procedować.

I nasza reakcja powinna być bardzo, bardzo stanowcza. Musimy bronić dobrych stosunków polsko-amerykańskich przed wasalizacją, dlatego nie możemy zostawić tak bezczelnego zachowania bez reakcji z naszej strony. Dziękuję. Pani poseł Magdalena Biejat, klub Lewicy. Wysoka Izbo!

Każdy: czy to osoba prywatna, czy też przedsiębiorca, który otrzymuje decyzję urzędową w swojej sprawie, w sprawie swojej własności, musi mieć nie tylko możliwość zaufania temu rozstrzygnięciu. Musi mieć co do niego pewność i móc swobodnie podejmować dalsze działania, decyzje życiowe i inwestycje. Sytuacja przeciwna, która ma miejsce obecnie, gdzie decyzja wydawana z naruszeniem prawa może zostać cofnięta na wniosek strony trzeciej, nawet po upływie kilkudziesięciu lat, jest nie tylko drastycznym naruszeniem autorytetu państwa, podważeniem zaufania do instytucji publicznych i prawa jako takiego, ale jest też po ludzku, po prostu poniżająca dla obywatela. Zaufanie społeczne, prawdomówność, odpowiedzialność za decyzje i kroki, jakie podejmujemy wobec innych, stanowią fundament relacji międzyludzkich.

Chodzi bowiem nie tylko o jej namacalne działanie, o to, czy młoda rodzina może bezpiecznie kupić mieszkanie, czy dostanie na nie kredyt hipoteczny, chodzi nie tylko o lokatorów kamienic i bloków, do których są roszczenia, o firmy, które chcą inwestować, czy o ludzi, którzy wybudują sobie dom i mogą po wielu latach nagle dowiedzieć się, że muszą go rozebrać lub przebudować. Chodzi o elementarne poczucie sprawiedliwości, o pewność otaczającej nas rzeczywistości i swobodę podejmowania życiowych decyzji. Nowela art. 156 k.p.a. to krok w kierunku państwa prawa, któremu możemy zaufać, w którym każdy i każda może bezpiecznie podejmować życiowe decyzje. Warto, by to prawo, które służy naprawieniu dotychczasowych przepisów, było napisane dobrze, dlatego chciałabym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na kwestię trybu, w jakim mają być wygaszane postępowania o unieważnienie wadliwej decyzji. Taka konstrukcja nie występuje nigdzie indziej w postępowaniu administracyjnym. Co za tym idzie, brakuje jednolitej wykładni dotyczącej jej realizacji. W praktyce więc spowoduje to, że część organów będzie wydawać decyzję o umorzeniu postępowania, inne będą zawiadamiać strony o tym, że postępowanie zostało umorzone z mocy prawa, a jeszcze inne nie zrobią nic. Aby uniknąć dalszego chaosu i w pełni zrealizować słuszną intencję projektodawców, należałoby dodać przepis, który wskazywałby, że organ nie wydaje decyzji o umorzeniu postępowania, a jedynie zawiadamia strony o tym, że zostało ono umorzone z mocy prawa. Taką właśnie poprawkę jako klub Lewicy złożymy i bardzo polecam ją uwadze ministerstwa i większości parlamentarnej. Oczywiście jednym z kluczowych aspektów tej zmiany przepisów, o której nie sposób nie wspomnieć, jest kwestia wygaszenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Tego rozwiązania oczekuje od Wysokiej Izby ogół społeczeństwa, dlatego bardzo cieszy fakt, że nowela zyskała tak szerokie poparcie już w pierwszym czytaniu. Mam nadzieję, że to poparcie jednak się utrzyma, dlatego też apeluję do wszystkich klubów i kół parlamentarnych oraz do Senatu o jak najszybsze jej uchwalenie. Nie możemy jednak zapomnieć, że reprywatyzacja jest problemem daleko bardziej złożonym, wykraczającym poza Warszawę i dekret Bieruta czy część gruntów rolnych, których ta nowelizacja może również dotyczyć. Apeluję więc także: nie spoczywajcie na laurach i nie poprzestawajcie na zmianie jednego przepisu k.p.a. Nadal czeka na rozpatrzenie projekt ustawy reprywatyzacyjnej Lewicy, który kompleksowo rozwiązuje wszystkie związane z roszczeniami problemy. Nadal pozostają kwestie dotyczące wyceny reprywatyzowanych nieruchomości, a co za tym idzie - wysokości odszkodowań, weryfikacji prawdziwości roszczeń, uwzględniania ich faktycznego stanu czy obciążenia hipotecznego oraz przede wszystkim handlu roszczeniami. Także te kwestie wymagają pilnej uwagi Sejmu. Rozwiązanie przygotowane przez Lewicę leży i czeka. Liczymy, że krok w dobrym kierunku, jakim jest realizacja wyroku trybunału i zmiana art. 156 k.p.a., nie będzie krokiem ostatnim, a na kolejny obywatele i samorządy nie będą musieli czekać następnych 30 lat.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stanowiący podstawę projektowanej zmiany został wydany 12 maja 2015 r.

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Sejmu, zwróciła się do ministerstwa, że nie ma przekonujących argumentów, by nie można było wydłużyć vacatio legis do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co pozwoli stronom postępowania na przyswojenie nowej regulacji prawa.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie! Wysoka Izbo! Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważna ustawa, tak oczekiwana. Przyszedł moment na jej uchwalenie.

Państwo polskie, Sejm działają w ramach demokracji, podejmują wyzwania i je realizują. W toku dyskusji pojawiają się różne argumenty w przypadku okresu dłuższego, krótszego. Jakie są argumenty za jednym i za drugim? Bo trudno na podstawie tej naszej dyskusji powiedzieć, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Panie Marszałku! Otwarte drzwi do reprywatyzacji przez lata były, oprócz tej nadziei na przywrócenie krzywd, które wyrządzone zostały systemem komunistycznym, niestety drzwiami, przez które przemknęło się dużo niesprawiedliwości, cierpienia, bezduszności i niepewności. Konsekwentnie od kilku lat zamykamy te drzwi, wyrzucamy za nie oszustów, czyścicieli kamienic, zapewniamy spokój i bezpieczeństwo Polakom, którzy przez ten proces i niektóre osoby utracili zaufanie do naszego państwa. Sam proces reprywatyzacji, tak jak powiedziałem na wstępie, niósł nadzieję na naprawienie krzywd. Jednak po 30 latach można powiedzieć, że rachunek nie do końca jest taki, jaki spodziewano się na początku transformacji. Jednocześnie te 30 lat to był okres, w którym to, co się stało, powinno być już zamknięte. Dlatego ten projekt kompleksowo odnosi się zarówno do oczekiwań tych, którzy przez 30 lat oczekiwali naprawienia krzywd, jak i do tych, którzy przez 30 lat ponieśli nowe krzywdy. Dlatego też chciałbym powiedzieć, że ten projekt jest elementem pewnych zmian, które polski parlament przeprowadza w zakresie racjonalnego, odpowiedzialnego zamknięcia m.in. problemu reprywatyzacji, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego do tego się odnosił. Ale problem wzruszania decyzji administracyjnych po wielu latach, w przyszłości, kiedy już żyjemy w pełni demokratycznej Polsce, może przynieść inne niepożądane skutki. Dlatego ta ustawa jest bardzo ważna. Cieszy mnie, że od początku prac nad tym projektem unosił się duch odpowiedzialności za nasze państwo ze strony wszystkich klubów parlamentarnych.

Chciałbym podziękować pani poseł Barbarze Bartuś, która z wielką determinacją od wielu miesięcy przekonuje do prac nad tym projektem. Chciałbym podziękować przedstawicielom innym klubów i kół parlamentarnych, z którymi pracowaliśmy w komisji nad wypracowaniem najbardziej właściwego brzmienia przepisów, żeby w pełni realizowały zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak i te oczekiwania, które wobec klasy politycznej formułuje społeczeństwo. Dlatego też w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości wyrażam pełne poparcie dla tego, co zostało przez komisję wypracowane. Czy pani poseł sprawozdawca chce zabrać głos? Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Trybunał stwierdza: Z uwagi na zakres kontroli konstytucyjności, obejmujący pominięcie ustawodawcze, trybunał nie przesądził o tym, czy właściwym sposobem realizacji tego postulatu jest przewidziany aktualnie w art. 156 § 2 k.p.a. 10-letni termin prekluzyjny, który ogranicza stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych obarczonych niektórymi innymi wadami. Ustawodawca dysponuje swobodą w wyborze instrumentów prawnych służących realizacji wskazanych przez trybunał wartości konstytucyjnych. Ten akapit był takim punktem wyjścia do prac w komisji, w podkomisji nad przedstawionym przez Komisję Ustawodawczą projektem, który był ściśle wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyroku zakresowego. Dlatego też, o czym mówiłam w swoim wystąpieniu, przystąpiliśmy do całościowej nowelizacji tego art. 156 § 2, który był tutaj przedstawiony, a tak naprawdę dotyczyło to przesłanek określonych w paragrafie wcześniejszym, i uznaliśmy, że 10-letni okres to będzie jednak ten okres właściwy, po którym już nie uchyla się decyzji. Przyjęliśmy też dla wszystkich tych wad, o których jest mowa, dla których jest ustanowiony okres 10-letni, żeby jednak po 30 latach już nie prowadzić postępowania. Zrobiliśmy to w duchu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ trybunał wskazywał też na to, że przecież te dokumenty źródłowe też są niepełne.

Pan poseł zwracał się do ministra. To nie minister ustala vacatio legis, tylko ustawodawca. Na posiedzeniu komisji przyjęliśmy właśnie to 30-dniowe vacatio legis, a to z tego powodu, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że brak takiego terminu, takiego ograniczenia możliwości uchylania decyzji jest niekonstytucyjny, jest niezgodny z konstytucją, którą przyjęliśmy w 1997 r.

Ale jeżeli poprawki, które zostały złożone, będą wnosiły do naszego projektu takie zmiany, które mogą jeszcze ulepszyć ten projekt, przyszłą ustawę, na pewno nad tymi poprawkami się pochylimy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pracę. Tak jak pan minister powiedział, dla mnie to jest ważny projekt, bo dotyczy spraw, które znam, dotyczy niesprawiedliwości, która na ten moment się dzieje. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1222 i 1291) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam przyjemność przedstawić sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1222 i 1291. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła rządowy projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 22 czerwca.

Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Marek Ast w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera rządowy projekt. Projekt rzeczywiście ma prokonsumencki charakter, jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak będziemy wnosić do tego projektu jedną poprawkę, ponieważ na etapie prac rządowych zapis, który proponujemy w poprawce, się w nim znajdował.

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt jest realizowany w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłych w czterech sprawach, w tym w sprawie, która dotyczyła również Polski, o sygn. C-545/17.

Warunkiem jest wpisanie przez przedsiębiorcę do rejestru podmiotu zajmującego się doręczaniem jako operatora pocztowego w tym zakresie.

Wprowadzone zostaje również rozwiązanie, które obniża wysokość opłaty od zarzutu do maksymalnej kwoty 750 zł w przypadku, kiedy pozwanym jest konsument.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek doręczenia wraz z pozwem umowy głównej, która była zabezpieczona wekslem. Możliwe również będzie, zostało bowiem doprecyzowane, istnienie po stronie wnioskodawcy uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania. Te rozwiązania, skierowane głównie w stronę konsumenta, mają poprawić sytuację konsumenta właśnie w postępowaniu sądowym i jako takie przyczynić się do poprawy w zakresie tego postępowania. Niestety nie znamy kolejnej poprawki, którą kieruje klub większościowy funkcjonujący w obecnym Sejmie, w związku z tym trudno do niej się odnieść, ale poznamy ją jutro na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej i wtedy będziemy mogli ocenić zasadność treści tej poprawki. Miejmy nadzieję, że wpisze się ona w całokształt tego projektu ustawy (Dzwonek), by nie doszło do momentu, w którym, mimo że projekt jest przyjmowany przez wszystkie kluby poselskie, pojawia się rozwiązanie, które takiej akceptacji nie uzyskuje. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Obowiązkowa kontrola umowy, a nie tylko weksla, dłuższy termin przewidziany na odwołanie oraz niższe opłaty sądowe mające wzmocnić obywateli w sporach z przedsiębiorcami i zwiększyć ochronę konsumentów przed działaniami dużych firm, w tym banków - takie zmiany przewiduje rządowy projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawowy cel zmiany ustawy wynika z obowiązku wdrożenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciw konsumentom.

Wszystko po to, aby wychwycić niedozwolone postanowienia umowne. Należy pamiętać, że wydawany na posiedzeniu niejawnym do wydziału pozwanego, a nawet bez jego pisemnego stanowiska, nieprawomocny nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadania mu klauzuli, a jest to dla osoby pozwanej prawie tak samo dotkliwe jak zajęcie komornicze. Projekt poszerza też zakaz przenoszenia praw z weksla wystawionego przez konsumenta na inne osoby, np. firmy windykacyjne, i obejmuje nie tylko, jak do tej pory, kredyty konsumenckie, ale wszelkie umowy konsumenta z przedsiębiorcą. Taka ochrona ma obejmować nie tylko samego dłużnika, tj. stronę umowy zawartej z przedsiębiorcą, ale i poręczycieli. Występujący z pozwem nakazowym będzie musiał przedłożyć sądowi umowę zabezpieczoną wekslem. Bez tego sąd nie wyda nakazu i skieruje sprawę do zwykłego procesu, więc pozwany konsument uzyska możliwość prezentacji swoich racji przed wydaniem końcowego orzeczenia. W szczególnych przypadkach ma też wystarczyć samo oświadczenie pozwanego przed sądem o tym, że jest konsumentem, choć obarczone grzywną do 300 zł. Przedmiotowa zmiana ujednolica również terminy na odwołanie się od nakazu zapłaty, tzw. zarzuty, do 1 miesiąca, jeśli dłużnik przebywa na terenie Unii Europejskiej, oraz 3 miesiące, gdy doręczenie ma nastąpić poza Unią Europejską. Aby uniknąć komplikacji, terminy mają dotyczyć zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

To znacznie mniej niż obecnie w zwykłym postępowaniu. Projekt dostosowuje polskie przepisy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłych na kanwie spraw wniesionych z Polski oraz Niemiec. Dzięki proponowanym rozwiązaniom zwiększy się ochrona prawna obywateli. Konsumenci i inne strony postępowania cywilnego będą mogli korzystać z porównywalnego w całej Unii Europejskiej poziomu ochrony swoich praw.

Jeśli poprawka zgłoszona teraz w drugim czytaniu nie wpłynie na charakter i zapisy przedłożenia, to klub Lewicy tak jak do tej pory będzie podtrzymywał poparcie dla niniejszego przedłożenia. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze!

Ten projekt wydaje się właśnie takim projektem.

Czy nie warto - tak jak już mówiłem szerzej podczas pierwszego czytania - pomyśleć o odmiejscowieniu? Dzisiaj świat idzie do przodu.

To nie zmienia oczywiście faktu pozytywnej opinii o tym projekcie ze strony naszego klubu. Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera projekt tej ustawy. Cieszy nas dostosowanie wyroków TSUE do polskiego prawa. Cieszy uznanie wyroków TSUE przez polski rząd. Cieszy uznanie przez ministra sprawiedliwości wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I oby tak było zawsze, w każdym innym przypadku z wyrokami TSUE. Ale cieszy też debata przy tym projekcie. Była dyskusja, było spokojne rozwiewanie wątpliwości, a to bardzo rzadki obraz w ostatnich miesiącach w sejmowych pracach, chociaż hasło „gramy razem” dzisiaj dotyczy innej sfery. Bardzo dziękuję.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! I teraz jest Kodeks postępowania cywilnego. Dworczyka temat elektronicznej korespondencji budzi bardzo duże emocje. Tym bardziej warto w kontekście rozpatrywanego przedłożenia wspomnieć o osieroconym art. 165 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, który zawiera normę wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu. Ze sprawozdania komisji sprawiedliwości wynika, że projektodawcy nie dotknęli tego wyzwania, i to mimo już obowiązujących norm w ustawie o doręczeniach elektronicznych, która przygotowuje nas na cyfrową komunikację, m.in. z sądami. Prosta, przyjazna użytkownikowi, a przede wszystkim bezpieczna elektroniczna korespondencja jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju naszej gospodarki.

Panie Marszałku! Analizując proponowane zmiany, a zwłaszcza uzasadnienie, odnoszę wrażenie, że nowelizacja polskiego prawa odbywa się na zasadzie gaszenia pożarów. Gdzie zobaczymy dym, tam kierujemy wozy strażackie, które doraźnie rozwiązują problem. Brakuje tu działań systemowych oraz korelacji z innymi przepisami. Mamy przecież w polskim prawodawstwie jasno określone zasady dotyczące skutków umów zawartych z naruszeniem prawa czy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Pytanie, dlaczego więc tworzymy oddzielne przepisy dla każdego zjawiska gospodarczego, które zostało zakwestionowane, np. przez TSUE, miast stosować do niego istniejące, obowiązujące prawo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewicy. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ochrona ta była i jest jeszcze niewystarczająca w sytuacji, gdy kredyt konsumencki lub inna umowa zabezpieczone były wekslem in blanco. Prezentowane przepisy, które dostosowują nasze prawo do wyroku TSUE, w końcu to zmieniają. Powód będzie miał obowiązek dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument, a sąd będzie musiał tę umowę zbadać. Co więcej, pozew taki będzie można wysłać nie tylko przez Pocztę Polską, ale również w innych uprawnionych jednostkach nadawczych, a także poza granicami Polski. Tutaj, panie ministrze, wracam do mojego pytania z pierwszego czytania. Chciałbym się dowiedzieć, czy udało się panu załatwić, żeby mieszkańcy Bielska-Białej nie musieli jechać ze swoimi przesyłkami za granicę, do Republiki Czeskiej.

Wysoka Izbo! Mam pytanie w związku z poprawką. Pewnie ta poprawka, złożona przez klub Prawo i Sprawiedliwość, została skonsultowana w ministerstwie. Projekt ustawy dotyczył sześciu ustaw. Wśród nich nie ma ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a poprawka składana jest już w drugim czytaniu.

Mam więc pytanie: Jak mamy ocenić to działanie, skoro ustawa, której dotyczy poprawka, nie mieści się w projekcie? Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050.

Pan przewodniczący Marek Ast. Panie Marku, wczoraj wszyscy podawaliśmy sobie rękę, a dzisiaj pan przyszedł tutaj z jakiejś tajnej narady i proponuje pan poprawkę, o której pan nawet nie wspomniał. Pani poseł Barbara Dolniak powiedziała, jak ta poprawka naszym zdaniem powinna być oceniona. Panie ministrze, wczoraj również pan wszystkim dziękował i podawaliśmy sobie rękę. A więc słowa o tym, że tak fajnie było podczas debaty nad projektem tej ustawy, cofam.

Wysoki Sejmie! Ustawa jest bardzo ważna dla konsumentów, wzmacnia ich ochronę na etapie postępowania sądowego wobec przedsiębiorców ich pozywających.

W przypadku pierwszej kwestii, która była poruszona, chciałbym odnieść się do tego, że ten projekt wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

A spory, które toczymy z organami Unii Europejskiej, z moim ubolewaniem bez pełnego poparcia tej Izby, wynikają ze spraw, które w ocenie polskiego rządu nie zostały przyznane Unii Europejskiej. Tego dotyczą ewentualne spory, które między wierszami można było odczytać z pana wystąpienia. Druga kwestia dotyczy operatorów i możliwości mobilnego nadawania przesyłek. Zatem to od nich zależy, w jaki sposób zorganizują tę usługę swoim klientom. Jeśli konkretne firmy, które mogły świadczyć takie usługi, zdecydują się na wprowadzenie konkretnej usługi, o którą pan poseł wnioskuje, w świetle brzmienia tych przepisów będzie to dopuszczalne. O ile oczywiście, zgodnie z tymi zezwoleniami, które aktualnie te firmy posiadają, będzie to realizowane. Kwestia dotycząca składania elektronicznie spraw.

Ta rewolucyjna zmiana w polskim sądownictwie niedługo będzie wdrożona. Jest to bardzo duża, poważna operacja i zachęcam do korzystania z tej usługi.

Niemniej pan poseł ma stosowne instrumentarium wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, by do odpowiednich ministerstw w tym zakresie się zwracać. I pytanie pani poseł Dolniak dotyczące przedłożonej poprawki. Pan poseł Ast wskazał, że to, co jest w poprawce, znajdowało się w pierwotnym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Z uwagi na fakt, że ustawa zwiększa ochronę konsumentów i ochronę uczciwej konkurencji w ramach postępowań sądowych, takie brzmienie było w pierwotnym projekcie, ponieważ ustawa dotyczy właśnie lepszych warunków realizowania ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji. Z tego też powodu uprawnienie wskazane w tej poprawce, ażeby można było realizować uprawnienia wynikające również z prawa unijnego, a nie tylko polskiej ustawy, jest kierunkowo dobre.

To rzeczywiście będzie realizowane, więc mam nadzieję, panie pośle, że będziemy konsekwentnie dzisiaj i jutro grać razem i ta poprawka spotka się również z pana uznaniem - jeśli będzie stosownie przedyskutowana jutro na posiedzeniu komisji. Była przedmiotem prac nad tym projektem, więc dobrze się stało, że ona też finalnie będzie procedowana w komisji. Pan poseł Marek Ast, sprawozdawca komisji. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mogę więc jedynie podziękować za te deklaracje wsparcia dla projektu przez państwa posłów, członków komisji.

Tak że jeszcze raz chciałem podziękować za tę wspólną pracę w komisji. Dziękuję.

Panie ministrze, nie pytałam o pierwotny projekt rządowy. Co tam się znajdowało, to jest zupełnie inna kwestia. Pytałam o projekt, który znalazł się w Sejmie. W związku z tym pytałam o odniesienie do projektu, który znalazł się w Sejmie, a nie do projektu, który państwo gdzieś kiedyś przygotowywaliście i usunęliście z niego tę właśnie ustawę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1307.

Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1276 i 1307) Proszę pana posła Wojciecha Zubowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych na posiedzeniu, które odbyło się dzisiaj, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Były też poprawki merytoryczne, rozszerzające nieco pierwotny zakres ustawy, umożliwiające wytwórcom energii elektrycznej i mocy dostosowanie się do zmieniających się przepisów. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania rekomenduje, wnioskuje o uchwalenie załączonego projektu ustawy wraz z poprawkami. Kilka słów na temat samego projektu. Projektowane zmiany wynikają z dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Przepisy tego rozporządzenia weszły w życie z dniem 4 lipca 2019 r. i bezpośrednio na ich podstawie odbyła się już pierwsza aukcja mocy w roku 2020. Zgodnie z rozporządzeniem rynkowym istniejące już regulacje prawne dotyczące mechanizmów mocowych zdolności wytwórczych, takie jak rynek mocy funkcjonujący w Polsce, powinny być dostosowane do przepisów ww. rozporządzenia, i to niniejszym staramy się czynić. Rozporządzenie rynkowe ustanawia przepisy mające zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz wymogi dotyczące polityki ochrony środowiska, w tym limitów emisji

Szanowni Państwo! Mając na uwadze te zagadnienia, celem i zamierzeniem tych prac legislacyjnych i tej ustawy jest wprowadzenie i osiągnięcie takich rezultatów, jak: dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzenia rynkowego, wyeliminowanie niepewności po stronie uczestników rynku mocy w zakresie jego funkcjonowania po wejściu w życie rozporządzenia rynkowego w kontekście jego bezpośredniego stosowania, określenie rozwiązań w zakresie sposobu uwzględnienia limitu emisji w procesach rynku mocy oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i usprawnienie funkcjonowania procesów rynku mocy. Na koniec, Wysoki Sejmie, panie marszałku, prosiłbym, by parlamentarzyści opozycji, którzy będą próbowali zabierać głos w tejże sprawie, oddzielili kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego od polityki, bo niestety wśród tych głosów merytorycznych na posiedzeniu komisji, jak również po posiedzeniu komisji pojawiały się takie, które nie miały nic wspólnego ze stanem faktycznym. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy pan poseł Jan Warzecha, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS przedstawić stanowisko dotyczące zmiany ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w ustawie rozwiązania mają gwarantować sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymogów w zakresie polityki ochrony środowiska. Wśród najistotniejszych rozwiązań w nowelizacji jest spełnienie unijnych wymogów w zakresie polityki ochrony środowiska.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz podczas pierwszego czytania ustawy posłowie koalicji rządzącej zaproponowali dwie poprawki.

Wysoka Izbo! Pragnę przypomnieć, że w 2018 r. w Polsce wprowadzono rynek mocy, który spowodował przejście z rynku jednotowarowego, tylko energii, na rynek dwutowarowy, energii i mocy. Rozwiązania miały spowodować modernizację znacznej części majątku wytwórczego potrzebnego do prawidłowego bilansowania mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz budowę nowych bloków. Obecne zapisy ustawy o rynku mocy mają zmotywować nowych uczestników rynku, m.in. inwestorów planujących budowę magazynów energii. Mają wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i zmniejszyć ryzyko tzw. blackoutu, bo jak wiemy, najdroższa energia to ta niedostarczona. Jak pokazuje praktyka, koszty rynku mocy są dla biznesu niższe niż potencjalne straty związane z ryzykiem przerw w dostawie energii elektrycznej, które mogą generować milionowe straty wynikające z każdorazowego braku energii. Związana z wprowadzeniem rynku mocy tzw. opłata mocowa, doliczana do rachunków odbiorcy energii od stycznia 2021 r., to inwestycja w budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących jednostek wytwórczych, a także wsparcie dla elektrowni w dostosowaniu się do norm ekologicznych. W projekcie nowelizacji ustawy o rynku mocy zaproponowana została zaakceptowana przez Komisję Europejską nowa formuła naliczania opłaty mocowej. Wysoka Izbo! Procedowane rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, zwłaszcza przez tzw. odbiorców energochłonnych. Co ważne, mają one zastosowanie do wszystkich odbiorców, a zatem nie podlegają zarzutom o nieuprawnione stosowanie pomocy publicznej. Nowa propozycja naliczania opłaty mocowej nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, przyczyni się do zwiększenia stabilności systemu elektroenergetycznego, będzie premiować stabilny pobór energii i jej zużywanie w godzinach pozaszczytowych i pozwoli odbiorcom obniżyć ponoszone przez nich opłaty za energię.

W związku z tym, że zaproponowany mechanizm jest kluczowy dla zachowania konkurencyjności polskiego przemysłu i zachowania miejsc pracy małych i średnich przedsiębiorców, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przyjęcie tej ustawy i przejście do następnych prac nad ustawą. Pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Była to ustawa o rynku mocy. Generalnie system miał nam poprawić bezpieczeństwo, dać środki finansowe na to, żeby energia elektryczna produkowana z węgla mogła jeszcze funkcjonować, żeby kopalnie mogły się rozwijać, dostosowywać.

Czy nam się udało wygenerować nowe źródła, nowe elektrownie? Sami słyszeliśmy, że dalej system energetyczny Polski oparty jest w 2/3 na elektrowniach konwencjonalnych. Cały czas mówiliśmy o tym, że ten węgiel jest taki wspaniały, taki dobry, a nic nie robiliśmy, żadnych kolejnych kroków do przodu, żeby próbować zastąpić elektrownie konwencjonalne nowymi blokami, choćby gazowymi. Dzisiaj stoimy u progu konieczności budowania nowych elektrowni gazowych, a może i elektrowni działających w kogeneracji. I tak się dzieje, ale dzieje się to bardzo powoli. Dzieje się to dlatego, że rząd nie przygotował odpowiedniej reformy, transformacji energetycznej Polski.

Chodzi przede wszystkim o obniżenie opłaty mocowej dla jednostek o tzw. płaskim profilu zużycia energii, czyli zużywających podobne ilości prądu przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Te przedsiębiorstwa od początku domagały się stworzenia takiego mechanizmu, który w jakiś sposób będzie je również promował i chronił. Dzisiaj mam nadzieję, że uda się nam to zrobić i ten mechanizm zafunkcjonuje. Oczywiście jeśli popatrzymy (Dzwonek) na cały mechanizm związany z rynkiem mocy, to zauważymy, że aukcje miały doprowadzić do tego, że ta cena miała być konkurencyjna.

Zobaczymy, jak to się będzie bilansowało i jakie moce energetyczne zostaną zachowane.

Wysoka Izbo! Rzeczywiście dzisiaj odbyło się kilkugodzinne posiedzenie komisji, na którym omawialiśmy ten projekt ustawy.

Nie otrzymaliśmy informacji na temat tego, w jaki sposób dotychczas sprawdzał się rynek mocy, nie mieliśmy żadnych informacji na ten temat. Zabrakło też informacji na temat tego, w jaki sposób gospodarstwa domowe będą reagowały na zwiększoną opłatę mocową. Nie mamy informacji na temat tego, w jaki sposób Unia Europejska ustosunkuje się do tego, że w umowie społecznej mamy wycofanie się z węgla dopiero w 2049 r. To są po prostu nasze życzenia, negocjacje trwają, ale się nie zakończyły, więc tych pytań jest bardzo wiele.

Te pytania ciągle pozostają otwarte, zdajemy sobie sprawę z tego, że transformacja energetyczna, którą już przechodzimy, jest jednym z najbardziej skomplikowanych, trudnych i finansowo obciążających procesów, jakie w Polsce dzisiaj przechodzimy, ale z drugiej strony nie mamy odpowiedniego zaangażowania, wiedzy i merytorycznego podejścia, jeśli chodzi o te kwestie.

Nie można takich rzeczy robić, bo zniechęca się Polaków do włączenia się w cały system przekształceń, bo to ludzie muszą za to zapłacić. Pytanie, ile więcej zapłacą za tę ustawę mocową.

Dzisiaj i tak ta cena jest już dość wysoka.

W czym jest rzecz? Niech on daje szansę stworzenia, tak jak powiedziałem, niezależności energetycznej, a przede wszystkim niech przyspieszy nasze przekształcenia, jeżeli chodzi o przejście z węgla na czystą energię, bo to z kolei ma podwójne znaczenie, bo nasze zdrowie i zanieczyszczenie środowiska jako wtórna rzecz, klimat i te wszystkie rzeczy. Pan poseł to powiedział, pani poseł również. Brak zdecydowania, do końca nie wiadomo, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, bo to są trudne i skomplikowane rzeczy, ale ktoś powinien to zdecydowanie przeprowadzać, a przede wszystkim stworzyć wiarygodność. Mówimy, że nie będzie podwyżek, a podwyżki są; że będziemy ograniczać węgiel, a za tydzień mówimy: nie, jednak będziemy utrzymywać się przy węglu; że będziemy wprowadzać atom, a nic się nie dzieje w tym zakresie. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050.

Ta nowelizacja ustawy o rynku mocy robiona jest głównie po to, żeby dostosować zasady do rozporządzeń Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rynek mocy, bo do tej pory Polska po prostu nie spełniała wszystkich wymogów, np. jeżeli chodzi o limity emisji dla elektrowni, które mogą dostawać wsparcie. Projekt więc wprowadza przede wszystkim właśnie te limity emisyjności określone rozporządzeniem rynkowym, że tak powiem, rychło w czas. Nareszcie. Mamy oczywiście też uwagi, rynek mocy miał z założenia promować powstawanie nowych elektrowni, podczas gdy w zasadzie stał się trochę kroplówką dla węgla i przez to nie stymuluje faktycznie transformacji energetycznej, jak oczekiwano. Dla gospodarstw domowych to jest ok. 10 zł miesięcznie, więc wydaje się, że niewiele, natomiast tak naprawdę głównym płatnikiem są tu przedsiębiorstwa i instytucje, które zużywają 75% prądu w Polsce. I to tam głównie osadzony jest ten koszt, a koszt osadzony w tym miejscu sprawia, że jesteśmy coraz mniej konkurencyjni. Najgorsze jest to, że choć dostosowujemy się do wymagań Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu wciąż nie odpowiedzieli nam na pytanie, jak chcą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne państwa po 2025 r., kiedy już nie będzie można wspierać elektrowni węglowych. Nowelizacja zostawia też ewidentną furtkę - i o to też pytałam na posiedzeniu komisji i nie dostałam odpowiedzi - na dodatkowe wsparcie dla wytwórców poza rynkiem mocy. Pytanie, bo nie wiemy, kogo, w jakiej wysokości i jakie technologie rząd planuje wspierać. Bo jeśli chodzi o to, że energetyka węglowa odchodzi w niebyt wraz z kolejnymi decyzjami spółek o wyłączeniu, chyba już nikt nie ma wątpliwości. Zresztą problemy środowiskowe też to wymuszają, a co za tym idzie, wymogi Unii Europejskiej, ale kosmetyczne zmiany ustawy o rynku mocy tak naprawdę nie rozwiązują problemu z brakiem paliwa do transformacji całego sektora. Więc potrzebujemy jak najszybciej wzmocnić ścieżkę odejścia od węgla i plany zastąpienia mocy wytwórczej tak, żeby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne w kolejnych latach, bo w gruncie rzeczy ten spadek mocy wytwórczej jest już mocno oszacowany. Wiemy, jaki jest. Pytanie, czym go uzupełnimy, bo jeżeli nie uzupełnimy nowymi inwestycjami i pomysłami na wytwarzanie energii w inny sposób niż z węgla, to po prostu będziemy coraz więcej energii importować, a więc też będziemy coraz bardziej podatni na cenę energii importowanej i jej zachwiania.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające konwersję projektów na mniej emisyjne, ograniczając przy tym kary za niewykonywanie obowiązków mocowych. Taki projekt, panie ministrze, mamy jeden, nazywa się Ostrołęka i dobrze by było, żeby pan przyznał, że w ten sposób rozwiązujecie problem wysokich kar. Muszę się przyznać, że zgadzam się z posłem Warzechą właśnie w kontekście zwłaszcza Ostrołęki, że najdroższa energia to ta niedostarczona. Tak, panie pośle, najdroższa energia to ta niedostarczona, bo rodzi ryzyko przestojów, niedostarczania prądu do gospodarstw domowych, do fabryk. Również zgadzam się z ministrem Tchórzewskim, który mówił, że w naszym interesie ogólnokrajowym, wszystkich sił politycznych jest to, by w końcu przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną i by przestać udawać, że nie mamy problemu. Przy okazji zapytam już, panie ministrze, dlaczego ograniczacie inwestycje (Dzwonek), zniechęcając potencjalnych inwestorów nowymi planami legislacyjnymi ograniczającymi uzysk dla indywidualnych klientów z tego typu instalacji.

Panie Ministrze! Rzeczywiście mieszkańców, Polaków nie interesuje, jak się spiera obecny minister z byłym ministrem, który sobie wprowadził tę ustawę o rynku mocy, i tym, który dzisiaj chce ją zmieniać, ale interesuje, panie ministrze, czy wzrośnie po raz kolejny opłata mocowa, bo ona została wprowadzona w tym roku, i czy na rachunkach gospodarstwo domowe dostanie więcej. To jest najważniejsze i to dotyczy Polaków i prosiłbym o taką odpowiedź od pana ministra. W jaki sposób będzie modernizowana? Ta elektrownia też jest w potrzebie. Mówi się o jej likwidacji. Chcielibyśmy usłyszeć, jakie są plany i jak państwo dalej będziecie zmierzać w tym procesie restrukturyzacji czy transformacji elektroenergetyki? Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiono nam bardzo obszerny i naszpikowany specjalistycznymi terminami projekt. Tymczasem statystyczny Polak, który mało, że znajduje się w ogonie Unii Europejskiej pod względem płac, to jeszcze każdego miesiąca po otrzymaniu rachunku za energię elektryczną dostaje palpitacji serca. Rząd natomiast uspokaja Polaków i mówi, że 25 lat będzie lepiej. Dużo rzadziej rząd wspomina o 2 mld wydanych na bloki energetyczne, które teraz za kolejny 1 mld trzeba rozebrać. Nie wspomina o 30-letniej umowie z górnikami, na mocy której będziemy wypłacać im uposażenie, w sytuacji gdy inni Polacy na przebranżowienie dostają rok albo i mniej. Dlaczego z tych pieniędzy nie są też finansowane rekompensaty za podwyżki cen prądu dla wszystkich Polaków? Uprzejmie proszę, panie ministrze, o odpowiedź na piśmie. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ocenie skutków regulacji do tej ustawy, o której mówimy, czytamy: ustanawia przepisy mające zapewnić funkcjonowanie rynku energii oraz wymogi polityki ochrony środowiska, w tym także limitów emisji CO2. Szanowni Państwo!

Kolega zapytał: Czy udało się wygenerować nowe źródła energii?

Jakie państwo z rządu mają plany w tym zakresie?

Panie Ministrze! Panie ministrze, kilka pytań. Prosiłbym tylko o potwierdzenie, bo padły zapytania i pewne chyba wymagające sprostowania informacje dotyczące pierwotnej ustawy o rynku mocy. Po pierwsze: Czy niewprowadzenie tych rozwiązań z roku 2018 mogłoby spowodować, jak szacowano wtedy straty sięgające ok. 10 mld zł rocznie? To jest raz. Po drugie, panie ministrze: Czy wprowadzenie rynku mocy pozwoliło przedsiębiorcom produkującym energię elektryczną na rozpoczęcie inwestycji, na zapewnienie stabilności, jeżeli chodzi o finansowanie? I po trzecie, panie ministrze, proszę również o informację: Czy wprowadzenie rynku mocy, wprowadzenie tzw. opłaty mocowej pozwoliło na spowolnienie wzrostu cen energii przede wszystkim teraz zależnych od kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla?

Wysoka Izbo! Czy będą miały zwiększoną opłatę mocową?

I z drugiej strony: W jaki sposób też wpłynie to, czy macie państwo też takie szczegółowe informacje, na ten rynek gospodarki energochłonnej? Teraz głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Piotr Dziadzio. Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Postaram się odnieść do pytań bardzo kompleksowo, aczkolwiek niektóre pytania trzeba potraktować indywidualnie.

No tak, oczywiście, że wzrośnie. I wiemy, rozmawialiśmy na ten temat i mamy tutaj pewną jasność. Drugie pytanie: Co dalej z Rybnikiem? Więc czekamy, aż te jednostki wszystkie wejdą do rynku mocy tak naprawdę, więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Kolejne pytanie, Łaziska. Mamy plan inwestycji związanej również z umową społeczną w Łaziskach. Myślę, że to jest satysfakcjonujące, bo następuje progres rozwojowy. Dobrze.

Wszystkie te zagadnienia są opisane bardzo dokładnie w polityce energetycznej państwa.

Inwestycje, które były planowane, zostały zrealizowane.

Pytanie Lewicy. Muszę sobie tylko sprawdzić.

Przedsiębiorstwa utrzymają swoją konkurencyjność na rynku. Myślę, że na wszystkie pytania zostały.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Wniosek o odwołanie pana Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Minuta przerwy? Dobrze, ogłaszam minutę przerwy. W takim razie, proszę państwa, ogłaszam 15 minut przerwy.

Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o odwołanie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego była jego wypowiedź polityczna. Sport uczy szacunku do rywala, do przeciwnika. Gloria victis, chwała zwyciężonym, nie biada zwyciężonym, panie marszałku. Chwała zwyciężonym, czyli szacunek dla rywala. Można te słowa przenieść i do świata polityki. Można rywala politycznego nie lubić, nie zgadzać się z nim, ale należy tego politycznego rywala szanować. W Sejmie marszałek Sejmu szacunek powinien okazywać każdemu posłowi, a Ryszard Terlecki dał się w ostatnich latach poznać jako symbol złych standardów zarządzania parlamentem i lekceważenia praw opozycji. Można by wspomnieć wydarzenia z sali kolumnowej z grudnia 2016 r. Przecież pan, panie marszałku, złożył zeznania, w których stwierdził pan wprost, że salę zorganizowano wówczas tak, aby nie dopuścić posłów opozycji do stołu prezydialnego. Pozostańmy jednak przy wydarzeniach z tej kadencji. W listopadzie 2020 r. wicemarszałek Terlecki nie stanął w obronie posłanki Barbary Nowackiej, wobec której policja użyła gazu łzawiącego. Nie stanął także w obronie posłanki Małgorzaty Biejat. Przepraszam, pani poseł. A przecież to było w oczywisty sposób naruszenie nietykalności jednej i drugiej posłanki. W tej kadencji wicemarszałek Terlecki został ukarany przez komisję etyki za słowa: puknij się w czoło skierowane do wybitnego posła Pawła Zalewskiego. A to przecież już w ramach recydywy, bo należy nadmienić, że i w poprzedniej kadencji komisja etyki zwróciła uwagę na niestosowne zachowanie marszałka Terleckiego wobec posła Sławomira Nitrasa, którego nazwał wtedy pajacem. 15 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu Sejmu Ryszard Terlecki przeszkadzał w wypowiedziach, a prośbę posłanki Katarzyny Kretkowskiej, by przywrócił jej należny czas, skomentował słowami: żadna strata. 27 października 2020 r. w sali sejmowej skierował pan, panie marszałku, do posłanek następujące słowa: Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. 15 sierpnia 2020 r. po wystąpieniu posłanki Klaudii Jachiry wicemarszałek Terlecki stwierdził: Na głupotę nie ma rady. A 4 maja 2021 r. świadomie nie dopuścił pan do głosu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w toku dyskusji nad ratyfikacją decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych Unii, pomimo wyrażanej przez niego woli zabrania głosu. Jedna z sejmowych sal otrzymywała imię wybitnej posłanki Olgi Krzyżanowskiej. Powyższe przypadki wskazują na to, że wicemarszałek Ryszard Terlecki nie sprawuje godnie swojej funkcji. Jego wypowiedzi godzą w rację stanu, są obraźliwe wobec posłów, zaś sposób wykonywania przez niego obowiązków narusza prawa zarówno opozycji, jak i członków Rady Ministrów. Drogie Panie Posłanki! Pani marszałek Gosiewskiej, która ciągle tutaj komentuje, przypomnę, że zgodnie z art. 10 ust. 3 regulaminu Sejmu. wicemarszałkowie Sejmu zastępują marszałka w zakresie przez niego ustalonym. Do obowiązków marszałka należy zgodnie z art. 10 stanie na straży godności, powagi i praw Sejmu oraz reprezentowanie Sejmu, godne reprezentowanie. W świetle powyższych faktów nie ma wątpliwości, że Ryszard Terlecki nie daje rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków, choćby dlatego, panie marszałku, że tak cenione w świecie sportu słowa gloria victis, chwała zwyciężonym, są panu niestety obce tu, w parlamencie. Dziękuję, panie pośle. Obecnie proszę pana posła Krzysztofa Śmiszka o przedstawienie również uzasadnienia wniosku z druku nr 1305. Proszę. Wysoka Izbo! Klub Lewicy wraz z kołem Polska 2050 zdecydował się na złożenie wniosku o odwołanie pana Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka polskiego Sejmu z wielu powodów. Pan poseł Tomasz Zimoch wymienił kilka z nich. Postaram się powiedzieć o tym, który jest bezpośrednią przyczyną naszego wniosku. Pan Ryszard Terlecki już od dawna przyzwyczajał nas do swoich aroganckich wypowiedzi. Pół biedy, że obrażał w ten sposób posłów i posłanki opozycji. Mówi się: psy szczekają, karawana idzie dalej. Dokładnie w ten sam sposób pan Terlecki obraża obywateli, sejmowych dziennikarzy czy ostatnio przedstawicieli białoruskiej opozycji prześladowanych przez autorytarny reżim, na którego czele stoi arogancki i butny satrapa, który myśli, że wszystko mu wolno, arogancki i butny satrapa, który chciałby koncesjonować opozycję i mówić ludziom, co im wolno, a czego nie wolno. Brzmi znajomo? Zresztą to nie jest tylko przypadłość pana Ryszarda Terleckiego. Pan jest tylko twarzą pewnej choroby, która dotknęła Prawo i Sprawiedliwość, choroby, która toczy całą waszą formację. Zamieniliście je na: arogancja, nepotyzm i rozpasanie. PiS, rząd, posłanki, posłowie i wasze pociotki w spółkach Skarbu Państwa. Wy już nie znacie granic. Skoro możecie wszystko, to myślicie, że faktycznie wszystko wam wolno, ale to nieprawda. Pan, panie marszałku, zapomniał, że jako jednej z najważniejszych osób w państwie wolno panu mniej, a nie więcej, bo pana głos, o zgrozo, może być postrzegany jako głos polskiego państwa, a pana twarz jako twarz tego rządu formacji rządzącej. I bardzo często to państwo i ten rząd pan kompromituje na arenie wewnętrznej i międzynarodowej. W innej sytuacji można byłoby komuś takiemu poradzić, żeby zanim się odezwie na głos, dwa razy się zastanowił, czy warto, albo żeby nie pisał szybciej, niż myśli - widocznie w przypadku pana marszałka Terleckiego ręce są zdecydowanie szybsze niż głowa - ale pan Ryszard Terlecki w kwestii arogancji jest recydywistą, i to niereformowalnym. Ktoś, kto po prostu nie potrafi zachować się inaczej niż arogancko, nie powinien pełnić funkcji marszałka polskiego Sejmu. Ktoś, kto nie rozumie, że interes białoruskiej opozycji jest zbieżny z polską racją stanu, że powinniśmy ją wspierać ponad podziałami, powinien zniknąć z polskiej polityki i sam poszukać pomocy w Moskwie, bo ktoś, kto dezawuuje dramatyczną walkę białoruskiej opozycji, podważa szczere intencje odważnych działaczy, a zwłaszcza działaczek, jest tylko pożytecznym pomagierem Putina. To, co powiedział i napisał pan Terlecki, po prostu podcięło skrzydła tym, którzy walczą z reżimem, tym, którzy płacą za swoją walkę pobiciami, gwałtami, bezprawnym pozbawianiem wolności czy torturami, niekiedy życiem. Kilka tygodni temu miałem okazję spotkać się we Wrocławiu z rodzicami Ramana Pratasiewicza. Widziałem ich łzy, widziałem ich rozpacz, ich rodzicielską troskę o życie i los ukochanego syna. Widziałem także wdzięczność za to, co Polska robi na rzecz ich kraju, a także ich syna. Widziałem także nadzieję, że ten koszmar kiedyś się skończy, bo kraje Zachodu stoją po stronie demokracji, wolności i praw człowieka, bo na Polskę można liczyć, bo stoi po stronie tego wszystkiego, o co walczy ich syn. A potem jedną wypowiedzią jednej z najważniejszych osób w państwie ta nadzieja znika, bo wicemarszałek Sejmu wplątuje Swiatłanę Cichanouską, działaczkę opozycji demokratycznej, w polskie piekiełko, w partyjny jazgot, który nie bierze jeńców, który nie zważa na to, że tuż za polską granicą mamy do czynienia z Koreą Północną Europy, bo najważniejsze dla niego jest to, czy Cichanouska spotka się z polską opozycją, czy też nie. Swiatłana Cichanouska jeździ po świecie, nie poddaje się w walce o swój kraj, włącza w tę walkę kolejne państwa i kolejne rządy, kolejne międzynarodowe instytucje i organizacje. Nieustannie mobilizuje instytucje Unii Europejskiej, w tym jakże aktywny Parlament Europejski. W każdym demokratycznym kraju przyjmowana jest jak prezydentka elektka, z należnym jej szacunkiem, tylko u nas spotyka ją despekt, tylko u nas spotyka się z brakiem szacunku, tylko u nas wplątuje się ją w polityczne i partyjne piekiełko. Tylko u nas wicemarszałek polskiego Sejmu odsyła ją do Putina, tego samego, który ręka w rękę z Łukaszenką gotuje piekło Białorusinom. Wstydzę się, kiedy spotykam Białorusinów, kiedy prowadzę z nimi rozmowę o tym, co jeszcze możemy dla nich zrobić. Bo zamiast planów wsparcia muszę się tłumaczyć, czy Polska jest z demokratyczną opozycją białoruską, czy też zamyka oczy na tragedie i na nieprawości dziejące się na Wschodzie. Muszę ich uspokajać, że marszałek Terlecki to nie cała Polska, bo Polki i Polacy wiedzą doskonale, gdzie leży dobro i prawda, a te są tam, gdzie są wolni i odważni Białorusini, którzy są wspierani przez odważnych i prawych Polaków. Słowa marszałka Terleckiego godzą w polską rację stanu, w coś, co do tej pory było uważane za ponadpolityczne i ponadpartyjne, w coś, co wymykało się z podziału na opozycję i koalicję rządzącą. A taką racją stanu była demokratyczna, stabilna i wolna Białoruś. Pan marszałek Terlecki wplątał swoją wypowiedzią kwestię białoruską w bieżącą polską politykę i tym samym odbiera nadzieję tysiącom działaczek i działaczy białoruskiej opozycji. Te słowa dziwią tym bardziej, że pan marszałek Terlecki sam kiedyś był opozycjonistą. W latach 70., 80. sam poszukiwał wsparcia u tych, którzy wtedy mieszkali po demokratycznej stronie świata. Zatem tą wypowiedzią przekreśla także swój życiorys. Bo historyczne zasługi i bycie kombatantem nie zwalniają od tego, żeby być przyzwoitym, aby rozumieć procesy polityczne i demokratyczne, które dziś zachodzą u naszych wschodnich sąsiadów. Pan marszałek po międzynarodowej burzy spotkał się z panią Cichanouską. Zapewnił ją, że Polska wspiera dążenia demokratyczne - to dobrze. Ale niestety mam głębokie wrażenie, które podzielane jest przez wielu Polaków, a także Białorusinów i opinię międzynarodową, że odbyło się to za późno i niestety w złym stylu. Dzisiaj to Litwa przejmuje stery, jeśli chodzi o wspieranie Białorusinów. I być może pani Cichanouska zapewniała pana marszałka Terleckiego podczas spotkania, że nie chowa urazy, że wszystko jest okej, ale zaufanie zostało nadszarpnięte. Pytanie, do kogo zwróci się demokratyczna opozycja w kolejnych dniach, miesiącach i latach. Do Litwy czy do Polski? Ale nie tylko działaczka opozycji białoruskiej padła ofiarą mądrości pana Terleckiego. Były też inne grupy. Pamiętacie państwo słowa: a co, oni są normalni? Patrząc na poranne sceny w Sejmie, można śmiało powiedzieć, że niestety, ale standardami nie odbiega pan od naczelnego homofoba Polski, Przemysława Czarnka. Za słowami powinna iść odpowiedzialność, dlatego zwracam się do posłów Zjednoczonej Prawicy, do was, bo z wami wielokrotnie rozmawiam na korytarzach sejmowych i w kuluarach. Ile razy jeszcze chcecie świecić oczami za pana Ryszarda Terleckiego? Czy nie warto chociaż raz postawić interes Polski ponad interesem partyjnym? Przecież i tak część z was - o czym już powiedziałem - przyznaje w duchu, że ktoś taki jak pan Ryszard Terlecki bardziej wam szkodzi, niż pomaga. Tylko powiem tyle: Lewica z przyjemnością zagłosuje za wnioskiem o odwołanie pana Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka polskiego Sejmu. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę, o przedstawienie uzasadnienia wniosku z druku nr 1306. Proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Już sam sposób wyznaczenia tej debaty pokazuje, jak traktujecie polski parlament, jak traktujecie podejście do obowiązków, jak traktujecie obywateli. Pan wicemarszałek Terlecki stał się symbolem, symbolem waszej pogardy dla każdego, kto ma inne zdanie, dla każdego, kto śmie myśleć, czuć inaczej, niż chce tego obecna władza. Ale pan marszałek Terlecki nie jest odosobniony. Pan marszałek jest szefem waszego klubu. Pan marszałek jest jednym z najważniejszych funkcjonariuszy tego obozu władzy. Kiedy zabiera głos, wiemy doskonale, że to nie jest odosobniony głos. To jest linia waszej partii wyznaczana przez prezesa Kaczyńskiego. Gdybyście chociaż raz odcięli się od tych słów, gdybyście choć raz posypali głowę popiołem i powiedzieli: tak, przesadził. Przesadził, kiedy obrażał działaczkę białoruskiej opozycji. Przesadził, kiedy z pogardą, butą i arogancją zwracał się do parlamentarzystek i parlamentarzystów z innych frakcji politycznych. Ale nie. Wy zawsze brniecie w zaparte. Wy zawsze bronicie rzeczy nie do obrony. Dlaczego? Dlatego że pycha, arogancja i buta stały się sposobem na rządzenie. Stały się waszą legitymacją, stały się symbolem tej władzy. Dzisiaj, kiedy bronicie pana posła wicemarszałka Terleckiego, krzyczycie z tych ław, dogadujecie. Bo to jest wasz jedyny sposób na prowadzenie dialogu politycznego. Dzisiaj nie odważycie się wypowiedzieć bardzo prostego słowa. Słowa: przepraszamy.

Kiedy pan wicemarszałek Terlecki w sposób absolutnie niedopuszczalny odniósł się do prezydentki elekta, Swiatłany Cichanouskiej, to zamiast przeprosić, zamiast poprosić o honorową dymisję, brnęliście w to dalej. że na czele białoruskiej opozycji stoi osoba, która wyciągnęła rękę, by ratować waszego marszałka. Zrobiła to dla stosunków polsko-białoruskich. Nie patrzyła na to, że obrażaliście naród białoruski wołający o wolność. Nie patrzyła na to, że odsyłaliście ją do Putina, nie patrzyła na to, że słowa pana wicemarszałka Terleckiego cytowały rosyjskie i białoruskie agencje, tylko wyciągnęła rękę, dlatego że w przeciwieństwie do was jej zależy na jej kraju, jej zależy na dobrych stosunkach z Polską. Jej zależy na czymś, czego wy nie rozumiecie. Nie wiecie, co to jest dialog. Nie wiecie, co to jest parlamentaryzm. Nie będę powtarzał tych słów, które wypowiadał pan wicemarszałek Terlecki, tego, jak zwraca się do posłów, z jaką pogardą, bo ja nie wymagam od was szacunku do siebie. Nie wymagam szacunku do moich koleżanek i kolegów, bo wystawiacie świadectwo sobie, ale jedno, czego żądam na tej sali, to szacunek do wszystkich wyborców. Postawa pana marszałka Terleckiego to nie jest obrażanie tylko tej części sali, ale to jest obrażanie każdej Polki i każdego Polaka, którzy mają inne zdanie niż wasz obóz władzy. Tak, o panu senatorze Jackowskim. Pal licho, że to mówi o nas, ale nawet o waszym koledze mówi tak: Jest szkodnikiem.

Otóż wczoraj pokazaliście kwintesencję tego, z jaką hipokryzją podchodzicie nawet do symboli, które zwykle macie na sztandarach. Wczoraj, w 3. rocznicę śmierci marszałek Olgi Krzyżanowskiej była wyjątkowa uroczystość, która połączyła wszystkie frakcje polityczne, połączyła wszystkich na tej sali. Chcieliśmy wspólnie oddać cześć osobie wybitnej.

Co się okazuje?

Ostentacyjnie wychodzi. To jest rzecz bez precedensu. Możemy pominąć wszystkie nasze spory. Możemy zapomnieć wszystkie słowa, którymi zwracał się do posłanek i posłów opozycji, ale tym gestem obraził symbole, które do tej pory były święte dla nas wszystkich. Obraził symbole Armii Krajowej. Obraził symbole Polski Walczącej. Obraził wielkie ofiary, które ponosili nasi rodacy w ciężkich czasach, bo właśnie przez tę bezczelność, panie marszałku.

Dzisiaj pan zatracił możliwość reprezentowania nas wszystkich. Bo pan nie jest na tej sali wicemarszałkiem PiS-u.

Pan, siedząc na tym miejscu, pełni funkcję marszałka Sejmu, marszałka całego Sejmu. A pan w sposób absolutnie bezczelny odbiera głos, komentuje, obraża. Pan wystawia świadectwo całej klasie politycznej i na to nie ma zgody posłanek i posłów opozycji. Pan nie ma prawa reprezentować osób, którymi pan gardzi. Godność człowieka powinna wyznaczać wartości, w oparciu o które będziemy wspólnie pracować, a pan jest w stanie.

Jeżeli pan nie jest w stanie odciąć się od haniebnych słów ministra Czarnka obrażających Polki i Polaków, jeżeli pan jest w stanie tylko to potwierdzać, to wystawia pan sobie świadectwo. Dzisiaj niestety zajęliście miejsca w tych ławach, żeby bronić rzeczy nie do obronienia. Dogadujecie, przekrzykujecie, tylko potwierdzając, że ten wniosek jest zasadny. Wy odwykliście od debaty parlamentarnej.

Wy myślicie o polemice? Przecież zachowujecie się tak, że tylko potwierdzacie, że przykład idzie z góry. Ale jak możecie nie popierać swojego partyjnego kolegi, jak macie zwykłych ludzi w głębokiej pogardzie?

Obrady prowadzę ja, nie pan. Państwo nie reagujecie. Panie pośle, belkę. Panie pośle, drzazgę widzicie w cudzym oku, ale w swoim belki nie widzicie. Proszę kontynuować, panie pośle. Więc jeśli dzisiaj przed tą debatą ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, czy wniosek opozycji o odwołanie pana wicemarszałka był zasadny, czy też nie, to myślę, że przebieg tej debaty pokazuje, że pan marszałek uosabia wszystkie najgorsze cechy parlamentaryzmu, które wnieśliście do tej Izby. Raz jeszcze chcę podkreślić, że zamieniliście miejsce debaty, miejsce sporu politycznego w arenę jedynej słusznej partii. Wy nie rozumiecie, czym jest dialog, wy nie rozumiecie, czym jest parlamentaryzm.

I dzisiaj, kiedy mówimy o wniosku o odwołanie pana wicemarszałka Terleckiego, [[Oklaski]] miałem nadzieję, pani marszałek, że pani w imieniu waszej większości parlamentarnej przeprosi za to zachowanie, że będziecie w stanie.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Ubolewam nad tym, że życiorys, który kiedyś mógł być dla mojego pokolenia wzorem, pan przekreślił w ostatnich latach właśnie przez tego typu arogancję i butę. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak człowiek z taką przeszłością, jak człowiek, który kiedyś walczył o ideały, jak człowiek, który kiedyś walczył o polską wolność. dzisiaj stał się symbolem właśnie tego, jak można walczyć z własnymi obywatelami. Nie jestem w stanie zrozumieć, że człowiek z takim życiorysem może przez ostatnie lata przekreślić wszystko, co osiągnął. Ale niestety ta debata pokazuje też, że nie ma z waszej strony żadnej refleksji.

I możecie państwo jeszcze wiele krzyczeć, możecie państwo jeszcze nas obrażać, ale nie zmieni to faktu, że wicemarszałek Sejmu pan Ryszard Terlecki stracił moralne prawo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Funkcja wicemarszałka Sejmu to jest niesamowity prestiż. To jest zobowiązanie wobec całej Izby.

Jednym wpisem przekreślił pan 30 lat polskiej polityki wschodniej. Odesłał pan liderkę opozycji do Moskwy, a potem nie powiedział pan nawet słowa „przepraszam” Sejm ustalił, że w dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

Wysoka Izbo! Uspokójmy tę debatę i porozmawiajmy merytorycznie. O Białorusi porozmawiajmy, szanowni państwo. Od ostatnich prezydenckich wyborów na Białorusi. sfałszowanych w taki sposób, że było to widoczne dla całego świata, obserwujemy, jak reżim Łukaszenki nasilił agresywne działania wobec swoich obywateli. Białorusini, którzy mają już dość promoskiewskiego dyktatora, odważyli się dać temu wyraz w masowych demonstracjach i protestach. Reżim odpowiedział represjami i prześladowaniami, bezprawnym zatrzymywaniem, aresztowaniem wielu osób, torturami, doszło też do aktu państwowego terroryzmu, porwania samolotu, aresztowania białoruskiego opozycjonisty pana Protasiewicza. Łukaszenkowskie represje bardzo mocno dotykają też naszych Polaków, naszych rodaków ze Związku Polaków na Białorusi. Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys. Chcę mocno podkreślić, że Polska bardzo poważnie traktuje wydarzenia na Białorusi. Stoimy po stronie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Polska wspierała i wspiera procesy demokratyczne u naszych sąsiadów. I, szanowni państwo, w tak trudnej, dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Białoruś, uaktywniły się w Polsce osoby czy ugrupowania, które chcą na tym skorzystać, zbić kapitał polityczny, wykorzystując do tego białoruską opozycję. Wstyd! Tak właśnie zrobił wasz polityk, Rafał Trzaskowski, który. który za pieniądze niemieckiej Fundacja Konrada Adenauera. organizuje antyrządową inicjatywę. I wszystko po to, szanowni państwo, by wyrąbać swoje miejsce w tonącej Platformie Obywatelskiej. Trzeba to jasno powiedzieć: organizuje działania, które - to nie jest tajemnica - mogą być zaczątkiem nowej partii politycznej. Do swojej indywidualnej, prywatnej kariery świadomie, celowo, bezczelnie i cynicznie, jednym słowem, totalnie wykorzystał Swiatłanę Cichanouską, liderkę białoruskiej opozycji demokratycznej. Wstyd, szanowni państwo! I to jest ten kontekst, na który trzeba zwrócić uwagę w całej tej sprawie. bo, szanowni państwo, każdą ideę można wypaczyć i skrzywić. I to właśnie zrobił wasz polityk Rafał Trzaskowski. Bardzo przykre jest to, że w sposób przedmiotowy. traktuje, a raczej wykorzystuje, osobę, która walczy o wolność swojego kraju, o wolność swoich rodaków. W tym kontekście wpis wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, nacechowany wzburzeniem, odnosił się do tak poważnej sprawy, jak manipulacyjne wykorzystywanie idei wolności obywateli Białorusi przez opozycyjnego, polskiego polityka. Przypomnę: Prawo i Sprawiedliwość wspiera obywateli Białorusi w ich dążeniu do wolności i niepodległości, nie wykorzystując do własnych działań politycznych, szanowni państwo. To rząd Prawa i Sprawiedliwości szybko i sprawnie, od razu, od początku masowych protestów, zorganizował pomoc dla represjonowanych. Przypomnę tylko kilka działań: ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla wydalanych studentów, pomoc niezależnym mediom i organizacjom pozarządowym wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Wartość programu pomocowego dla Białorusi, który przygotował rząd to ile? Pakiet pomocowy „Solidarni z Białorusią” i wsparcie studentów oraz pracowników naukowych. Nie chcecie tego słyszeć. Nie chcecie tego widzieć. Doliczę pani czas. Proszę państwa, to jest klasyczny przykład przeszkadzania, ale jak potem z tej strony są głosy, państwo bardzo protestujecie. Bardzo proszę, żeby zachować spokój i dać możliwość wypowiedzenia się mówcy do końca, dobrze? Mogę?

A co wy robiliście w okresie swoich rządów? Przypomnę, szanowni państwo. Słynna sprawa Alesia Bialackiego. czyli ujawnienie białoruskiemu reżimowi przez polską prokuraturę danych tego opozycjonisty. Jaki był skutek? przez białoruski sąd polski MSZ pod kierownictwem waszego ministra Radosława Sikorskiego. wysłał ok. 30 białoruskim opozycjonistom deklaracje podatkowe PIT z danymi wrażliwy. Korespondencja wysłana listem poleconym z logo ministerstwa. Powiedzmy sobie szczerze: daliście Łukaszence na tacy informacje, które wprost uderzyły w opozycję białoruską. Nie pamiętacie? Kolejna sprawa. Białoruski uchodźca skazany na 3 lata więzienia przez polskie sądy w Białymstoku za waszych rządów na podstawie waszych działań. Boli? Boli? Pani marszałek, proszę zmierzać do końca, dobrze? Proszę. W ostatnim czasie pan marszałek Terlecki. spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską. Sprawa została wyjaśniona, czego nie raczyliście zauważyć. Po tym spotkaniu sama zainteresowana powiedziała: Ryszard Terlecki, Marek Pęk, Włodzimierz Bernacki odwiedzili mnie dzisiaj w Wilnie i wyrazili pełne poparcie dla białoruskiego ruchu demokratycznego. Ogłosili kontynuację programów stypendialnych dla naszych studentów. Zapewnili mnie, że wszystkie partie w Polsce stoją za Białorusią. Ja się tylko zastanawiam, czy rzeczywiście wszystkie? Bo my to robimy, a wy tylko krzyczycie. A więc, szanowni państwo, może wreszcie zróbmy coś razem. Spotkajmy się pod ambasadą Białorusi. w walce właśnie o demokrację na Białorusi. Pamięta pan jak razem to robiliśmy.

Nie przypominam sobie takiej samej reakcji, kiedy podobnych słów używał pan marszałek Terlecki: przecież ja nie wiedziałem, że on wstanie, nie wiedziałem, że on wyjdzie, nie wiedziałem, że nie będzie siedział. i 10 razy wymieniła nazwisko: Trzaskowski. Ani razu nie wymieniła nazwiska: Terlecki. Ani razu. Jak go broniła? Pan Terlecki nie chciał siedzieć, podobnie zresztą jak ja. Pamiętamy to wszystko, pamiętacie państwo - rozmawiamy o tej Izbie - jak zwracał się do parlamentarzystów, jak mówił do parlamentarzystek. A czy pamiętacie państwo, jak wyrywał mikrofon i kabel z kamery dziennikarzowi na korytarzu? Wyrywał. A pamiętacie, jak podjął uchwałę o wyrzuceniu dziennikarzy z Sejmu? Czy dziennikarze pamiętają, kto wyrzucił ich do baraku obok budynku? To nasza determinacja sprawiła, że dziennikarze mogą relacjonować prace Sejmu. Bo wy sprowadzilibyście ten Sejm do Sejmu relacjonowanego przez Orlen media.

Problem polega na tym, że to Polska powinna pomagać Białorusi, a nie białoruska opozycja - polskim ministrom i polskim marszałkom, [[Oklaski]] którzy zachowują się jak Łukaszenka, tak jak Łukaszenka na PGR.

Zacytuję wam taką parafrazę wielkiego dzieła polskiej kultury: Miły panie, po co pytos, przecież Gucwa to nie Witos. Ja mam nadzieję, pani marszałek - również dla pani dobra, żeby panią nie rządził, tak jak rządzi do tej pory - że ten epizod skończy się dzisiaj, bo nawet posłowie Konfederacji mówią, że ten sposób sprawowania władzy jest czymś kompromitującym dla Izby. Kontynuacja.

A jakim prawem państwo próbujecie zamiast mnie prowadzić obrady? Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Opozycja jak zwykle łże.

A pod jego miłą i sympatyczną twarzą kryje się takie monstrum, które, szanowni państwo. które buduje swoją pozycję na radykalizmie (Dzwonek), na obrażaniu innych parlamentarzystów, obrażaniu dziennikarzy, obrażaniu opozycjonistów z innych krajów.

Panie pośle, przekroczył pan tutaj granice. To, co pan przed chwilą zrobił, jest niedopuszczalne. Dziękuję, panie pośle. 33 sekundy miał pan. Absolutnie nie. Proszę bardzo. Panie pośle, koniec pańskiej wypowiedzi.

Bardzo proszę. Pani poseł Magdalena Biejat. Proszę bardzo, pani poseł. Pani poseł, zapraszam. Rezygnuje pani z wypowiedzi, pani poseł?

Ja jednak chciałabym wykorzystać chwilę, którą teraz mam, żeby powiedzieć o kimś znacznie ważniejszym - o Białorusinkach i Białorusinach, którzy nadal dzielnie walczą o swoje prawa. Chcę mówić o działaczce opozycyjnej i polityczce Swiatłanie Cichanouskiej. która mimo całej machiny propagandowej, mimo braku niezależnych mediów i środków docierania do wyborców, mimo strachu przed represjami była w stanie przekonać do siebie ogromną większość społeczeństwa białoruskiego. 9 sierpnia ub.r. wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Białorusi, stała się twarzą wołania o demokrację w Europie Wschodniej i choć została zmuszona do opuszczenia kraju, nie zaprzestała walki. Aleksander Łukaszenka nie zgodził się oddać władzy. Zamiast tego wypowiedział wojnę białoruskiemu społeczeństwu. Kiedy mówię: wojna, nie mam na myśli wojny symbolicznej, walki politycznej, ścierania się idei. Mam na myśli fizyczną przemoc stosowaną przez władzę wobec obywateli, siłowe pacyfikowanie protestów, porwania, bicie i zastraszanie. Do tego momentu wiadomo na pewno o czterech ofiarach śmiertelnych, ale może być ich znacznie więcej. Pierwszą był Alaksandr Tarajkouski, zabity przez milicję na ulicy podczas pierwszych sierpniowych protestów. Alaksandr Wichor, 25-latek, został śmiertelnie pobity przez milicjantów kilka dni później. Jego matka mówi, że nawet nie brał udziału w protestach, po prostu jechał do dziewczyny i przypadkiem znalazł się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Kolejny był Giennadij Szutow, postrzelony w głowę na demonstracji. Wreszcie w listopadzie zeszłego roku na posterunku zakatowano na śmierć Ramana Bandarenkę, artystę, który odnawiał mural przedstawiający i symbolizujący opozycję, walkę opozycji o demokrację przeciwko władzy Łukaszenki. Zaledwie miesiąc temu w więzieniu zmarł Witold Aszurak, więzień polityczny, odsiadujący 5-letni wyrok za organizację zeszłorocznych protestów. Miał 50 lat, był zdrowy. Władze podają, że przyczyną śmierci był atak serca. Nie ma wyników sekcji. To mogą nie być wszystkie ofiary śmiertelne, wieści niełatwo przedostają się przez granicę.

To się teraz dzieje na Białorusi, teraz umierają tam ludzie, nie gdzieś daleko, na drugim końcu świata, ale w Mińsku, 500 km od Warszawy.

chciałabym powiedzieć panu marszałkowi Terleckiemu: Atakowanie w tym momencie białoruskiej opozycji, brak wsparcia dla jej liderek i liderów ze względu na jakieś małe, żenujące wojenki z polską opozycją jest po prostu poniżej standardów, których należałoby oczekiwać od polityków w demokratycznym państwie. Pańska postawa przynosi wstyd nie tylko panu, ale także całemu Sejmowi. Dlatego Lewica wraz z Polską 2050 złożyła wniosek o odwołanie pana z funkcji wicemarszałka i zachęcamy państwa wszystkich do zagłosowania za. Dziękuję. Głos ma poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Od początku tej debaty towarzyszy mi takie przygnębiające wrażenie, że to chyba jest jeden z najsmutniejszych momentów w historii współczesnego parlamentaryzmu polskiego. I wiemy, jaki jest powód tej debaty - słowa wypowiedziane przez pana marszałka Terleckiego do liderki białoruskiej opozycji. żeby pomocy szukała w Moskwie. Nie będę się pastwił nad słowami i działaniami pana marszałka Terleckiego.

Jako profesor historii powinien wiedzieć, że spośród narodów, które tworzyły Rzeczpospolitą Polską Obojga Narodów, Białorusini od początku byli najbardziej przyjaznym nam narodem, język starobiałoruski był językiem kancelarii, oficjalnym, urzędowym, Wielkiego Księstwa Litewskiego, z nimi nasi przodkowie tworzyli jedno wielkie, wspaniałe, europejskie państwo. Jest to naród, z którym napięć na tle etnicznym i religijnym prawie nie znajdziemy. Nie znajdziemy w historii relacji polsko-białoruskich takich momentów, tragicznych momentów, jakie możemy znaleźć na Wołyniu czy w historii Wołynia. Pan prof. Terlecki musi o tym wiedzieć i musi wiedzieć, że dzisiejsi Białorusini - w tym również prawie 0,5 mln Polaków mieszkających na Białorusi, nie imigrantów, nie Polonii, ale Polaków tam urodzonych, [[Oklaski]] którzy nie chcieli nigdy z tamtego kraju wyjechać - marzą o demokratycznym, wolnym, niezależnym państwie, które będzie miało dobre relacje z Rzecząpospolitą Polską. Pan prof. Terlecki musi to wiedzieć i nie jestem w stanie zrozumieć, skąd wzięły się najpierw w jego głowie, a następnie w jego ustach słowa: idźcie po pomoc do Moskwy. Bo Białoruś jako obszar i Białorusini, ich serca, ich umysły, byli zawsze przedmiotem rywalizacji, a nawet, powiedziałbym, walki pomiędzy nami a Rosją, pomiędzy Zachodem i Wschodem. Białorusini dali wyraz temu, gdzie jest im bliżej, podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Bliżej im jest do Zachodu, bliżej im jest do Polaków. I wysyłanie ich do Moskwy to jest wysyłanie ich w łapy, w których nie chcą się znaleźć, bo zbyt długo w tych łapach byli i zbyt długo te łapy ich ciemiężyły. Nie wiem, jak raz powiedziałem, skąd to się u pana wzięło, ale przywołam słowa pana politycznego przyjaciela, partyjnego i politycznego mentora, który cytując Kornela Ujejskiego, mówił: inni szatani byli tam czynni. Tam musieli być jacyś szatani czynni. Niech pan tych szatanów ze swojego serca, ze swojego umysłu, ze swojej działalności przepędzi. Bo ci szatani trują polską politykę, zatruwają relacje polsko-białoruskie i sprawiają, że to, co jest dla naszego narodu, dla naszego państwa kluczowe, czyli poczucie bezpieczeństwa, jest narażone na szwank. Powiem więcej, jest narażone na szwank poczucie nie tylko Polaków i nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej, tej współczesnej, którą z takim trudem, wysiłkiem, my - nasi rodzice i za chwilę nasze dzieci - budujemy. Zagrażają bezpieczeństwu Europy. Pan to musiał wiedzieć, więc niech pan się z tymi szatanami rozprawi. Niech pan mi ich nie zabiera na tę salę, niech pan ich nie sadza obok siebie i niech panu nie podpowiadają. Bo na świecie jest dużo dobra. Jestem przekonany, że ono zwycięży, i chciałbym, żeby pan znalazł się kiedyś po stronie zwycięskiego dobra, a nie przegranego, przeklętego zła. Ale żeby tych szatanów przepędzić, potrzebna jest panu przerwa w wykonywaniu obowiązków marszałka Sejmu.

Dziękuję. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Marszałku Terlecki! Hipisie, opozycjonisto, historyku, naukowcu, profesorze, pośle, marszałku, karząca ręko Jarosława Kaczyńskiego skierowana na odcinek sejmowy, mistrzu bezemocjonalnej impertynencji. Będziemy głosowali za pańskim odwołaniem. Będziemy głosowali za pańskim odwołaniem, ale nie tylko ze względu na ową bezemocjonalną impertynencję, która niestety ma niekiedy tendencję do przeradzania się również na tej sali, również w sprawowaniu tej funkcji w bucowatość. Ale, panie marszałku, będziemy głosowali, ponieważ pańskie sprawowanie tej funkcji jest najlepszą miarą tego, jak fasadowy stał się ten parlament, jak fasadowe stało się obradowanie w tym parlamencie, w którym najważniejsze tematy państwa, najważniejsze tematy, wokół których powinna się koncentrować debata, albo nie są poruszane, albo są przepychane kolanem. Ten parlament, w którym oczywiście standardy, przepraszam za wyrażenie, chamstwa już dawno zostały bardzo wysoko postawione, a ustanowił je.

Przepraszam.

I ten poziom chamstwa będzie ciężko przebić, naprawdę, nawet marszałkowi Terleckiemu.

Bo gdyby był taki namysł i gdyby była taka przestrzeń do debaty, której państwo nie stwarzają - podobnie jak poprzednicy, ale to nie jest żadna zasługa, że nie jest się lepszą jakością - to ten parlament również oceniłby naszą politykę od 30 lat wobec Białorusi, wobec państwa białoruskiego.

To tak samo było krew w piach - i jedno, i drugie. Dlaczego? Dlatego że Polska nie ma rozstrzygających argumentów wobec sytuacji na Białorusi: gospodarczych, politycznych ani militarnych. Prawda jest taka, szanowni państwo, że nadmierne inwestowanie w taką czy inną ekipę na Białorusi przez ostatnie 25 lat po prostu się nie sprawdziło, po prostu poniosło porażkę. Tym bardziej, jeśli słyszymy - w sierpniu ubiegłego roku, w apogeum protestów - z wiarygodnych źródeł bardzo jasny przekaz płynący z Berlina, z Brukseli, z Waszyngtonu, że zależność, w jaką Łukaszenka wpędził Białoruś wobec Rosji, sprawia, że Zachód oczekuje od Moskwy, że to ona będzie rozwiązywała problemy na Białorusi, bo dzisiaj tak wielka jest zależność tego państwa od Moskwy. I jeśli to słyszymy i to wiemy, chodzi o te wszystkie czynniki, i mamy 25 lat doświadczenia w relacjach z tym państwem, to musimy sobie odpowiedzieć jedno: że jedynym możliwym do osiągnięcia priorytetem, który był w zasięgu ręki - pod warunkiem że jest najważniejszym priorytetem w naszych relacjach z tym państwem - jest walka o prawa kulturowe i oświatowe naszej mniejszości na Białorusi. To jest to, co jest w zasięgu i co pod stałą presją całej klasy politycznej, niezależnie od tego, jaki będzie rząd, jest możliwe do uzyskania, ale musi to być priorytetem numer jeden, bo żadnego innego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Taka jest po prostu ponura prawda. Prawda jest też taka, szanowni państwo, że niektórzy z was mówią o tym, że jeśli dzisiaj będziemy inwestować w bardzo dobre relacje z opozycją białoruską, to jak oni kiedyś przejmą władzę (Dzwonek), to będą wobec Polski życzliwi.

Najlepsi przyjaciele będą nas ignorowali, jeśli będziemy słabi, a najwięksi wrogowie będą musieli brać nas pod uwagę, jeśli będziemy silni. I przede wszystkim to - a nie sentymenty takie czy inne - powinno decydować o polityce wobec Białorusi.

Dziękuję również za ten wybuch radości. Panie Marszałku Terlecki! Chciałabym na początek zadać panu pytanie bez agresji.

Jak pan by się poczuł, gdyby ktoś o pana dziecku powiedział: to jakiś świr?

Pan nie obraża tych posłów, pan obraża łącznie ok. 200 tys. ludzi, którzy na nich głosowali. W 1989 r. rozpoczął się w Polsce proces zmian, który można podsumować czterema słowami: demokratyzacja, urynkowienie, samorządność, Europa. To pierwsze słowo: demokratyzacja oznaczało tworzenie nieraz od zera lub przekształcanie instytucji państwa, na których opierają się demokratyczne systemy polityczne - praworządność, trójpodział władzy, pluralizm polityczny. Wśród zadań, które wtedy były przed nami, przed Polakami, w 1989 r., było też odbudowanie znaczenia Sejmu po latach komunizmu, kiedy to ten Sejm odgrywał rolę fasadową. Rozpoczął się demontaż demokracji, demontaż rynku, demontaż samorządności i demontaż polskiej pozycji w Europie i na świecie. Moglibyśmy odwołać pana, panie marszałku Terlecki, za niewłaściwe wpisy na Twitterze, za prostackie, aroganckie, prymitywne czasami, opryskliwe traktowanie posłów i posłanek, ale zasłużył pan na odwołanie, bo jest pan jednym z najbardziej odpowiedzialnych za demontaż instytucji polskiego parlamentaryzmu, [[Oklaski]] a tym samym trójpodziału władzy. I tak zostanie pan zapamiętany przez historię. Sejm przestał być miejscem debaty i poszukiwania najlepszych dla Polaków rozwiązań ustawowych, stał się atrapą. jedną z wielu atrap instytucji polskiego, dumnego państwa, takich jak Trybunał Konstytucyjny - również jest atrapą - KRS i różne inne. Przypominam panu, że demokracja to rządy większości, ale przy poszanowaniu praw mniejszości. Wy cały czas o tym zapominacie, że demokracja jest rządami większości, ale przy poszanowaniu praw mniejszości. To ma swoją nazwę politologiczną, to jest tyrania większości. Wielokrotne łamanie konstytucji przez ten Sejm, głosowanie nad ustawami mającymi wyraźne konstytucyjne wady.

Wielokrotne łamanie konstytucji, głosowanie nad ustawami mającymi wyraźne konstytucyjne wady. łamanie ustaw, łamanie regulaminu Sejmu, procedur, tradycji, dobrych obyczajów wypracowanych przez lata, skracanie czasu wypowiedzi do absurdalnych, liczonych w sekundach wystąpień, odrzucanie choćby najbardziej racjonalnych uwag, nocne obrady, że nie wspomnę o głosowaniu nad budżetem w sali kolumnowej, stosowanie trybu poselskiego, żeby nie przeprowadzać konsultacji społecznych, brak odpowiedzi na pytania, brak odpowiedzi na interpelacje lub traktowanie tych interpelacji (Dzwonek) w sposób lekceważący - to wszystko są wasze zasługi. Powiem tak: Panie marszałku Terlecki, wydaje się, że jest pan dzisiaj Ryszardem wszystko mogę Terleckim. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

Nie będę odpowiadać na to, co tu usłyszeliśmy, bo nie wszyscy z tych, co występowali, powinni mówić to, co mówili. Chcę wyjaśnić dwie kwestie: jedna to taka, o której można dyskutować, druga jest obrzydliwą insynuacją. Jeżeli chodzi o pierwszą, to dotyczy pani Cichanouskiej. Pani Cichanouska spotykała się z różnymi środowiskami opozycji, zarówno z Platformą, jak i z Lewicą. Ja, jak bywałem na Białorusi, spotykałem się zawsze z liderami opozycji. Uważałem to za coś oczywistego i normalnego. Natomiast czym innym było, gdy osoba, która weszła do polityki, jawnie, otwarcie opowiada się po stronie sporu politycznego w Polsce i deklaruje udział w antyrządowym przedsięwzięciu, które organizuje wiceprzewodniczący opozycyjnej partii. Gdy spotkałem się z panią Cichanouską w Wilnie, wyjaśniłem to jeszcze raz. To nie jest odpowiednia rola dla osoby, która pozyskuje poparcie dla swojego narodu, swojego ruchu w walce z dyktaturą. To, że opowiedziała się za tym, zadeklarowała udział w przedsięwzięciu antyrządowym w kraju, w którym rząd wspiera opozycję w sposób, powiedziałbym, zasługujący na uznanie. bo to premier naszego rządu upominał się w Unii Europejskiej o wsparcie dla opozycji białoruskiej, to jest coś niewłaściwego.

Myślę, że to wyjaśnienie zrozumiała.

Prezydium wszyscy opowiedzieliśmy się za tym, że tę salę rzeczywiście należy tak nazwać. Po drugie, wzięliśmy udział w otwarciu, można powiedzieć, oficjalnym nazwaniu tej sali imieniem pani Olgi Krzyżanowskiej. W czasie tego otwarcia miały miejsce dwa wystąpienia: pani marszałek Sejmu, a także bardzo godne uznania wystąpienie pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Te wystąpienia podkreślały znaczenie tej postaci, której poświęcona była sala, i wyjaśniały, dlaczego tak należało tę salę nazwać. Po nich wystąpiła trzecia osoba, która uznała, że jest to dobra okazja, żeby nas obrazić, obrazić mnie. obrazić osoby, które były na tej sali, bo nie byłem jedynym przedstawicielem naszego obozu.

To jest, panie Budka, ordynarna nieprawda. Właściwie na tym mógłbym skończyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć coś, co powinienem powiedzieć, wyrazić moje zaskoczenie, zaskoczenie pozytywne. Bardzo gratuluję pani z Lewicy tego wystąpienia, które tu usłyszałem, bo ono odnosiło się do bardzo ważnych kwestii. A to, że pani przychyla się do wniosku o moje odwołanie, to jest kwestia oczywiście polityczna. Ma pani do tego prawo.

Wysoka Izbo! To właśnie te słowa pana posła Terleckiego pokazują, że nic nie zrozumiał z tej debaty.

Mówiła o tym, w jaki sposób został zamordowany jej ojciec. Ostrzegała i przestrzegała przed wykorzystywaniem prokuratury i sądów do spraw politycznych. Dzisiaj pan poseł Terlecki mówi o tym, że inicjatywa polityczna jest wymierzona w rząd, ma na celu obalenie rządu. Nie rozumiecie państwo, czym jest dyskurs polityczny, czym jest spór polityczny, czym jest coś, co jest normalne w parlamencie.

Proszę państwa, gość nie powinien obrażać gospodarza, który go zaprasza.

To się wydarzyło. Zamykam drzwi i nie wracam do tego.

Jeszcze jedno, jest przerwa.

Podoba się pani takie zachowanie? Podoba się pani? Bo mi nie, proszę państwa. To jest miejsce, gdzie możemy dyskutować. A po drugie, marszałek Sejmu, bez względu na to, czy to jest pani marszałek Kidawa-Błońska, czy pan marszałek Czarzasty, mają przycisk, pilnują czasu i są zobowiązani do tego, żeby przestrzegać regulamin. Państwo są zobowiązani do tego, żeby temu regulaminowi się podporządkować i słuchać poleceń marszałka. Przerwa do godz. 20.15.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Kamińskiego (druki nr 1261 i 1279) Proszę pana posła Marcina Kierwińskiego o przedstawienie uzasadnienia wniosku.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziwna to praktyka zaiste, aby minister nie stawiał się wtedy, gdy ma się odbyć głosowanie nad wotum nieufności wobec niego.

Ale zaiste, pani marszałek, dziwna to praktyka. Podstawą do złożenia tego wniosku był raport na temat wyborów kopertowych, przygotowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. O tym będę mówił za chwilę, ale to, co jest zapisane w tym raporcie, to jest tak naprawdę kolejna odsłona, to są kolejne objawy choroby, którą znamy z przeszłości. Całkowite łamanie prawa, buta i arogancja wobec elementarnej sprawiedliwości i wreszcie traktowanie państwa jak prywatnego folwarku. Należało się tego spodziewać, w końcu takie samo zachowanie pana ministra Mariusza Kamińskiego w latach poprzednich doprowadziło do tego, że został on skazany na 3 lata więzienia i 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych.

Czy pan minister Kamiński przeprosił kiedykolwiek za to, co robił wtedy, gdy za pierwszym razem był ministrem? Nie. Czy wyraził skruchę? Nie, zawsze był tak samo butny, zawsze był tak samo arogancki. A to ułaskawienie spowodowało u niego tylko i wyłącznie jeszcze większe poczucie bezkarności, jeszcze większe poczucie pychy i efekty tego widzimy. Powodów do odwołania pana ministra Kamińskiego jest bardzo, bardzo wiele. Każdy z nich sam w sobie, mógłby stanowić w normalnym demokratycznym państwie prawa powód do dymisji pana Kamińskiego, tylko w każdym normalnym demokratycznym państwie pan Kamiński nigdy nie byłby ministrem, i to jest podstawowy problem. Bo pan minister Kamiński nie ma moralnego mandatu, a zdaniem sądu przez 10 lat nie może sprawować funkcji w administracji centralnej. Szanowni Państwo! Wybory kopertowe, tak jak powiedziałem, to podstawa naszego wniosku. Pan Mariusz Kamiński wraz z panem Jackiem Sasinem, panem ministrem Dworczykiem i wreszcie panem Morawieckim naruszyli prawny i konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej. Wnioski z tego raportu można streścić w czterech bardzo prostych słowach: wielokrotne łamanie prawa i konstytucji. W ten sposób pan minister Kamiński dołączył do niechlubnego panteonu PiS-owskich urzędników, którzy już nie raz złamali i prawo, i konstytucję. Pan minister Kamiński wziął udział w wielkim marnotrawstwie publicznych pieniędzy. Minister, którego rolą, którego obowiązkiem jest dbać o interesy ekonomiczne kraju, uczestniczył w procederze rabowania budżetu państwa.

Taki ktoś w normalnym demokratycznym państwie powinien zasiąść na ławie oskarżonych, to naturalne, i zasiądzie. To z resztą nie jest dla pana ministra Kamińskiego niczym nowym. Działania, które podejmowali ministrowie rządu PiS w związku z wyborami kopertowymi, w tym pan minister Mariusz Kamiński, doprowadziły do gigantycznych strat w budżecie państwa. Ale gdyby nawet ta strata wynosił jedną tylko symboliczną złotówkę, to taki minister powinien być natychmiast odwołany, a wy powinniście się tego domagać, wy jako rządząca większość.

To jest działanie ministra konstytucyjnego państwa polskiego? Nie, to jest działanie, które bardziej przypomina działania zwykłych ordynarnych przestępców. Minister Kamiński doskonale wiedział, że wszystko to, co robił w związku z wyborami kopertowymi, jest nielegalne. Nie podpisał umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, ponieważ bał się. Bał się, że ten podpis, podpis na tej umowie będzie formalnym powodem do tego, aby stawiać mu zarzuty. Dziś będzie odpowiedzialność polityczna, a prędzej czy później będzie odpowiedzialność karna. Pan minister Kamiński zasłynął także tym, że pod jego rządami policja zachowuje się w sposób niebywale brutalny. Chyba nikt na tej sali nie ma żadnych wątpliwości, że wszystko to dzieje się z polecenia, a przynajmniej za aprobatą pana ministra Kamińskiego. Wszyscy pamiętamy te sceny, gdy funkcjonariusze, tzw. tajniacy, funkcjonariusze bez mundurów, używając pałek teleskopowych, bili polskie kobiety. Wszyscy pamiętamy, jak ci sami funkcjonariusze pryskali gazem łzawiącym w kierunku posłanek: posłanki Biejat, mojej koleżanki klubowej Barbary Nowackiej, mojej koleżanki Moniki Wielichowskiej. Za to wszystko. Każdy minister spraw wewnętrznych ma obowiązek przestrzegać, dążyć do tego, aby policja zachowywała się w sposób adekwatny. Zastanówmy się, czy adekwatne jest pryskanie gazem w kierunku posłanki, która pokazuje legitymację poselską. Czy adekwatne jest bicie pałką teleskopową kobiety, która spokojnie stoi na pokojowej demonstracji? Mając wielki szacunek do ciężkiej pracy codziennej policjantów, trzeba bardzo mocno powiedzieć: tę pałkę teleskopową w sposób symboliczny trzymał pan minister Kamiński. Ze służb mundurowych pan minister Kamiński uczynił policję polityczną. Policję, która bardziej dba o jednego obywatela niż o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Przecież wszyscy pamiętamy te obrazki, jak setki policjantów broniły jego szefa politycznego, Jarosława Kaczyńskiego. Nie broniły bezpieczeństwa Polaków, broniły jego szefa politycznego. Te wszystkie kordony naokoło pewnego bunkra na Nowogrodzkiej - to wszystko doprowadza do tego, że etos pracy w Policji spada. Pan minister Kamiński odpowiada za to, że na polskich ulicach pojawiły się obrazki rodem ze stanu wojennego. To jest jego odpowiedzialność. Pan Kamiński przez 3 lata swojego urzędowania postanowił przypomnieć Polakom, jak wyglądała i jak działała Milicja Obywatelska rządzona przez totalitarny reżim. To jest zasługa pana ministra Kamińskiego. I wreszcie chyba rzecz najgorsza, bo uderzająca bezpośrednio w etos pracy policjantów. Ta presja, ta patologiczna presja na policjantów i proste wyznaczanie, kto może awansować, a kto awansować nie może.

Trzeba to nazwać bardzo, bardzo jasno: to jest zbrodnia dokonywana na Policji. To jest zbrodnia na honorze policyjnym i na wizerunku Policji. Policja przez 30 lat odbudowywała swój wizerunek, cieszyła się wielkim zaufaniem społecznym. Do kiedy?

Pan minister Kamiński lubi chwalić się, lubi podkreślać swoją przeszłość opozycyjną.

Dalsze utrzymywanie na stanowisku pana ministra Mariusza Kamińskiego to będzie dalsza degradacja wizerunku polskiej Policji. Ostatnia afera mailingowa, afera, która dotknęła najważniejszych polityków PiS-u: pana premiera Morawieckiego, pana ministra Dworczyka. I jest coś bardzo charakterystycznego w tej aferze. Po raz kolejny służby specjalne zarządzane przez pana ministra Kamińskiego dowiadują się o aferze albo z mediów, albo z rosyjskiego komunikatora, albo z telewizji. Nie są w stanie nigdy działać w interesie bezpieczeństwa państwa. Zawsze coś prześpią, zawsze czegoś nie zauważą.

Tymczasem te służby działają jak trzy anegdotyczne małpki: nic nie widzą, nic nie słyszą i na koniec nic nie mówią, bo nigdy, po żadnej aferze służby specjalne rządzone przez PiS tak naprawdę nic nie powiedziały. Niszczenie polskich służb specjalnych, niszczenie polskiego kontrwywiadu, niszczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - to są fakty. Przecież od tego zaczął urzędowanie pan minister Kamiński. Dziś mówicie, że ABW prowadzi śledztwo w sprawie afery mailingowej.

Cała działalność ministra Kamińskiego to jest jeden wielki proces niszczenia polskich służb specjalnych. Ale jest jedna rzecz, którą pan minister Kamiński zrobił dla służb specjalnych, tylko nie wiem, czy obywatele mogą się z tego cieszyć. Zresztą pan minister Kamiński nie ma odwagi, aby się do tego przyznać. System, który stanowi swoistą broń podwójnego przeznaczenia, bo to system, którego serwery są w innym kraju. Nigdy pan minister Kamiński, nigdy pan minister Wąsik nie potrafili stanąć przed parlamentem i powiedzieć: tak, kupiliśmy ten system. Zawsze kluczyli, zawsze kłamali, zawsze oszukiwali. Więc może teraz panowie ministrowie powiecie: Kupiliście ten system. Panie ministrze Wąsik, ja wiem, że to pana śmieszy. Tylko nie śmieszy tych, którzy są podsłuchiwani. I na sam koniec, szanowni państwo: są pewne bardzo charakterystyczne wyznaczniki sukcesów pana ministra Kamińskiego, wystawione tak naprawdę nie przez polityków opozycji, nie przez media, tylko przez kolegów pana ministra Kamińskiego w tym rządzie. Pierwsza sprawa to kwestia ochrony wicepremiera do spraw bezpieczeństwa pana Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, że pan wicepremier nie chce korzystać z SOP-u, tak heroicznie budowanego i reformowanego przez Mariusza Kamińskiego. Woli płacić za prywatną ochronę, woli wykorzystywać Policję, bo boi się efektów własnych reform, boi się efektów pracy Mariusza Kamińskiego. To Jarosław Kaczyński mówi, że wszystko to, co robi Mariusz Kamiński, jest tak naprawdę do niczego. Posłuchajcie swojego prezesa. Zobaczcie, jak się zachowuje. I jest wreszcie drugi, także bardzo wymierny wyznacznik: kwestie inwigilacji, kwestie tego, że zwykły polski obywatel ma wielkie podejrzenia, czy nie jest w sposób nielegalny podsłuchiwany. Również pan premier Morawiecki z panem ministrem Dworczykiem wolą wysyłać e-maile ze skrzynki prywatnej, żeby tylko się nie archiwizowało, żeby tylko do tych danych archiwizowanych dostępu nie miał pan minister Kamiński (Dzwonek), bo jeszcze będzie ich inwigilował. Jeszcze będzie sprawdzał, co napisali w mailach. To jest poziom, tak naprawdę, braku zaufania, was, waszych ministrów do waszego. Dlatego, szanowni państwo, i zwracam się do posłów prawicy, wiem, że lojalność partyjna, że jesteście do tego często zmuszani, żeby tak głosować, ale zastanówcie się nad tym, czy bronienie człowieka, który codziennie sprowadza niebezpieczeństwo na Polaków, jest dobrą formułą.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Przedstawiam opinię Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 116 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 15 czerwca 2021 r. powyższy wniosek do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu zaopiniowania.

Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Przypominam, że zgodnie z art. 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębne elementy debaty.

Wysoka Izbo! Panie ministrze, pana tu naprawdę nie powinno być. Szkoda, że zabrakło panu tej refleksji, że naprawdę to nie jest miejsce dla pana. Lecz skoro pan już jest, to pan pozwoli, że zwrócę się również do pana kolegów, ale też i do pana. Jest pięć powodów, dla których nie powinno tu pana nadal być, nie powinien pan zasiadać w Wysokiej Izbie. To są wybory kopertowe, gdy łamał pan art. 7 konstytucji, zresztą nie pierwszy raz, mówiący, że władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Ten artykuł nie po raz pierwszy pan złamał. Art. 44 ustawy o finansach publicznych i art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień. Znowu dobrze znany panu artykuł do łamania. Poważne sprawy, bo dotyczą fundamentów demokratycznego państwa prawa, czyli tego, jak zorganizowane są wybory. Pan wiedział. Pan wolał nie zadawać pytań i pan wolał niczego nie podpisać. Zabrakło tej legendarnej odwagi? Gdzie ta siła z opozycji? Pamiętam, jak pan mówił tyle o honorze i godności, ale to były czasy, kiedy nie był pan ministrem od podsłuchiwania i inwigilacji. Jednak prawdziwą winą, którą ponosi pan wobec społeczeństwa polskiego, jest to, co Policja robiła z protestującymi. Z protestującymi przedsiębiorcami i protestującymi kobietami. Panie ministrze, pan był aktywistą - kiedyś. Pan mówił, że trzeba działać i że każdy ma prawo wyrażać opinie tak, jak chce - wtedy, kiedy był pan oskarżany o działania przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu czy ministrowi Wiatrowi. Wtedy rozumiał pan prawa obywatelskie. A co się stało teraz? A teraz wysyłał pan agresywną, źle wyszkoloną policję na protestujące kobiety. Godził się pan, żeby pałkami teleskopowymi były bite dzieciaki. Słyszał pan o panu Maćku, czternastolatku z Krapkowic? Policja przyszła do niego i go zastraszała, bo udostępnił post o proteście. A może słyszał pan o „Moli”, dziewiętnastolatce z Warszawy, której policja złamała rękę w czasie protestu? Czy może słyszał pan o czternastolatce z Olsztyna, którą w czasie protestu policja goniła, wyciągnęła, zastraszała i postawiła pod sądem za rzekomą organizację protestów? Przypomnę, mamy prawo protestować, mamy prawo bronić swoich praw i godności. a pan ma prawo jako minister stać również na straży praw obywatelskich. Parę dni temu słyszałam młodego chłopaka, który wyszedł na demonstrację pod ministerstwem edukacji przeciwko innemu z pana niegodnych kolegów, panu Czarnkowi. Czy to jest Rzeczpospolita, którą chcecie budować? Czy to jest Rzeczpospolita dla młodych? Oni wam tego nie zapomną. Straciliście młode pokolenie właśnie przez takie działania. Kolejna rzecz, w przypadku której nie powinien pan być ministrem, to jest to, co pan zrobił ze służbami i policją. Policjanci zaczęli się wstydzić mundurów, nie chcieli pałować kobiet, nie chcieli brać udziału w demonstracji, często przeciwko ich żonom, matkom i córkom. To jest to, czego minister nigdy nie powinien robić: hańbić munduru i zmuszać innych do jego hańbienia. Raport NIK wyraźnie stwierdza, że pan doskonale wiedział, panie ministrze, że firma związana z handlarzem bronią ma powiązania z czarną listą ONZ-u, a wydał pan rekomendację.

Panie ministrze, jak pan nadzoruje te służby, skoro handlarz bronią miał taką możliwość? Dlaczego tak się dzieje, że przymykaliście oko na przekręty w czasie, kiedy Polki i Polacy umierali i potrzebowali respiratorów? Minister Dworczyk. Przecież pan wie, panie ministrze, dlaczego oni używają prywatnych skrzynek. Bo nie chcą, żeby pan ich podsłuchiwał na służbowych. I to jest kolejna rzecz, którą niszczycie państwo polskie. Państwo Posłowie i Posłanki Prawicy! Dzisiaj pewnie się złamiecie, ale pamiętajcie, że my stoimy również po stronie waszych praw i tego (Dzwonek), żebyście byli bezpieczni w Polsce, tak jak każdy z nas. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wniosek podpisany przez prawie 70 posłów Koalicji Obywatelskiej jest wnioskiem, który opiera się na dwóch założeniach: w pierwszym wysnuwają informację, którą NIK przygotował, a w drugim grillują ministra Kamińskiego z tego powodu, że działa jako minister i nadzoruje policję. Reszta to jest właśnie grillowanie za działania policji. Są tutaj założone czy postawione zarzuty wobec pana ministra Kamińskiego, które kompletnie nie mają odzwierciedlenia w faktach. To jest tylko informacja ogólna, która zwraca uwagę, sugeruje. Ona sugeruje, żeby w państwie polskim przestrzegać prawa. Rewelacyjna informacja, którą NIK w tym raporcie przedstawił. To są wszystko elementy socjotechniczne, które państwo stosujecie od dawna w sposób przemyślany. Powiem tak: wybory, proszę państwa, to święto demokracji. Stawianie zarzutów premierowi i ministrom, w tym ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, że podjęli obowiązkowe działania związane z przeprowadzeniem wyborów, jest niedorzeczne i pozbawione logiki. Informacja NIK-u, na której posłowie oparli swoje zarzuty, jest porażająca swoją stronniczością, albowiem nie uwzględnia podłoża pandemii w tamtym okresie. Wniosek części posłów klubu Koalicji Obywatelskiej to czysta socjotechnika oparta na insynuacjach, sugestiach albo przeinaczeniach.

To jest niepoważne. Według wnioskodawców urzędnik nie może podejmować samodzielnie decyzji, albowiem za niego mają podejmować je inni. Całe szczęście, szanowni państwo, że mamy takiego premiera i takich ministrów jak Mariusz Kamiński, którzy potrafią podejmować takie decyzje, dlatego że te decyzje są dobre i trwałe dla naszego państwa. Wnioski z informacji NIK-u, na które powołują się posłowie wnioskodawcy, są kompletnie miałkie i bezzębne. Niech państwo wskażą w swoim wniosku, że ten raport mówi o naruszeniu prawa i postawieniu komuś jakichś zarzutów. Można więc postawić tezę, że informacja o wynikach kontroli NIK-u jest mięsem armatnim, które podano opozycji do grillowania rządzących, z czego wnioskodawcy z Koalicji Obywatelskiej skwapliwie korzystają. I tu rodzi się pytanie: Jak mocno można rozbujać naszą polską łajbę dla osiągnięcia celu przejęcia władzy w Polsce bez wyborów? To opozycja zachęcała podczas pandemii do wychodzenia na ulicę. To jest wojna. Ulica obali ten rząd. Tak dla przypomnienia, 800 osób pacyfikowanych w akcji „Widelec” [[Dzwonek]] jest państwa udziałem, który w historii zapisał się fatalnie. Stymulowanie akcji prowokacyjnych wobec policji, chęć zastraszenia policjantów, sugerowanie, aby policja nie interweniowała i nie podejmowała stosownych, przewidzianych prawem działań. Dzisiaj zresztą były w przemówieniu pana posła Kierwińskiego właśnie takie sugestie. Apelowanie, aby policja nie była wykorzystywana do celów politycznych i aby policjanci odmawiali wykonywania poleceń służbowych oraz działania zgodnie z prawem, zapewniania Polakom bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Minister Mariusz Kamiński stoi na czele ministerstwa, które zapewnia Polakom i Polkom możliwość pokojowego manifestowania i wyrażania swoich opinii i przekonań, ale w ramach istniejącego prawa. Jestem przekonany, że nie dopuści on do tego, żeby ten porządek był zmieniony, chociaż jest ogromne oczekiwanie, aby tak się stało i żeby ten brak bezpieczeństwa w polskim państwie zafunkcjonował. Szukanie tzw. winnych na siłę. Lansowanie przekazu: będziesz siedział. Panie Premierze! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego jest całkowicie bezzasadny, i będzie głosował za jego odrzuceniem.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! Ja myślę, że to nie jest największy problem. Uważam, że największym problemem jest pana poczucie, że broni pan bezpieczeństwa Polski, a tak naprawdę utożsamił pan bezpieczeństwo państwa z interesem i bezpieczeństwem swojej partii, Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest największy problem. Z tego wynika to, że co kilka miesięcy powracają kryzysy bezpieczeństwa. Przecież już kolejny raz rozmawiamy o naruszeniu bezpieczeństwa, zagrożeniu bezpieczeństwa. Kiedy PiS zadecydował, że chce zorganizować wybory kopertowe, żeby wykorzystać niski poziom zakażeń, jednocześnie obawiając się, że jego zwolennicy nie pójdą do tradycyjnych wyborów, odbyła się rzecz karygodna: przy stole ustalono, że przeznaczone na to zostaną środki spółek publicznych. Przekroczono uprawnienia. Pan premier wszedł w buty Państwowej Komisji Wyborczej. Nastąpiło naruszenie ładu prawnego. Czy w takiej sytuacji, kiedy koledzy przy stole dogadują się co do tak ważnych rzeczy, możemy założyć, że publiczne pieniądze są bezpieczne, gdy pilnuje ich Mariusz Kamiński? Moim zdaniem nie możemy. Na jesieni, kilka miesięcy później, Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem zabrał polskim kobietom wolność. Prawdopodobnie to były największe protesty w historii Polski po II wojnie światowej. Na serio. Taka jest prawda. Na ulicach pojawiła się także policja. Co się działo? Policja wystąpiła w interesie rządzących, uderzając w protestujących.

Czy obywatele, którzy byli zamykani w kotłach, obywatele, którym łamano ręce, obywatele, którzy byli traktowani gazem, mogą czuć się bezpiecznie, kiedy minister Kamiński ich pilnuje? Moim zdaniem nie mogą. Przecież od kilku miesięcy było wiadomo, że konta polityków są przedmiotem ataków. Był atak na konto minister Maląg, były ataki na konta posła Suskiego.

Co się stało po kolejnym ataku? Rząd mówi, że za atak odpowiedzialna jest Rosja, a wszyscy, którzy wskazują na błędy, na niedopatrzenia, są pokazywani jako ci, którzy sprzyjają rosyjskim interesom. Nie można uznać, że to jest poważna odpowiedź na ten kryzys. Natomiast można zapytać, czy bezkarni mogą czuć się ministrowie pilnowani przez Mariusza Kamińskiego. Moim zdaniem mogą się czuć bezpiecznie. I to jest nasz największy problem z ministrem Kamińskim: on jest przekonany, że robi bezpieczne wybory, że broni bezpieczeństwa na ulicach, że broni Polski przed atakami zewnętrznymi. A jakie są efekty? Powracające co kilka miesięcy kryzysy. Obywatele, którzy czują się coraz mniej bezpieczni. Obywatele, którzy nie ufają policji. Zaufanie do policji drastycznie spadło, jak nigdy w historii.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

I całe szczęście, że ta debata trwa, ponieważ jak słyszałem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, to nagle doszedłem do wniosku, że może te wybory się odbyły 10 maja. One się chyba jednak nie odbyły. Czy ktoś poniósł konsekwencje za to, że przeprowadził w ten sposób tę całą procedurę? Nie! Nasze państwo polskie nie jest przygotowane do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. W ogóle nie wiem, kto na ten pomysł mógł wpaść. 40 dni, bo 40 dni dano sobie na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych przy polskiej infrastrukturze. Szwajcarzy robili to 30 lat, Estończycy z małym państwem przygotowywali się ileś lat i to robili w formie elektronicznej. Amerykanie do dzisiaj narzekają na ten cały system. W Polsce, gdzie infrastruktura komunikacyjna funkcjonuje tak jak funkcjonuje, było to nierealne do przeprowadzenia. Z ignorancji, a ta ignorancja wypływa z arogancji. Nie słucha się nikogo. Jest to poważny problem. Musimy też pamiętać, że wyborów prezydenckich nie przelicza się na pieniądze. To nie jest tylko pieniądz.

Dobrze w ministerstwie o tym wiedziano, że tą decyzją się łamie, ponieważ nikt nie chciał się podpisać w wewnętrznej procedurze. Dlaczego? Pan minister też o tym dobrze wiedział, że to wszystko jest trochę na piechotę albo i więcej, że jest to łamanie konstytucji, łamanie prawa. A były inne środki. Może chodziło o to, żeby nie płacić przedsiębiorcom odszkodowania, gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Chcę państwu przytoczyć fragment pewnego reportażu, nie robię tego, ale to chyba warto.

Akcje dezinformacyjne z użyciem zhakowanych kont powtarzają się już regularnie co kilka tygodni, ale wzbudzają jedynie chwilowe zainteresowanie mediów, choć niezidentyfikowanym hakerom udało się przejąć konta pani marszałek Sejmu, kilku członków rządu, grupy posłów, w tym członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych, i samorządowców. Politycy wciąż nie traktują tego zagrożenia poważnie. Tylko, proszę państwa, jest jeden mały problem, zagadka: Kiedy ten artykuł był napisany? Kiedy ten artykuł napisano?

Czy zrezygnowano z korespondencji mailowej? Nie. Wie pani, jakie teraz wypływają informacje? Jakie będą wypływać? Teraz oczywiście to jesteście. Czy pan mnie słyszy?

Wysoka Izbo! Oskarżenie pod adresem ministra spraw wewnętrznych to poważna sprawa i trzeba mieć poważne argumenty.

mam w różnych krajach, oczywiście. Tak samo jest niepoważnym oskarżeniem. Natomiast najważniejsza sprawa jest inna. Oczywiście, że tak.

Gdybyście chcieli naprawdę to zrobić, to złóżcie wniosek o Trybunał Stanu. Ale to jest coś konkretnego, a wy grozicie, że jak dojdziecie do władzy, to wy go tam. Kontynuuje pan poseł Dobromir Sośnierz w imieniu Konfederacji. Po pierwsze, w lipcu 2020 r. w tygodniku „Najwyższy Czas” ukazał się tekst odsłaniający kulisy ataku wywiadowczego na Konfederację ze strony służb kierowanych przez pana ministra Kamińskiego. Chodzi o akcję pod kryptonimem „Sputnik”, która miała służyć wsparciu takiej PiS-owskiej narracji, PiS-owscy politycy często lubią wywoływać taki temat, że Konfederacja ma rzekomo jakieś związki z Rosją. W styczniu 2020 r. pan premier Morawiecki stwierdził np. coś takiego: proszę zauważyć, jak w ostatnich tygodniach zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje, politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki w dużym stopniu z Rosją. To pana wypowiedź, panie premierze.

Pan potem, bezczelnie kłamiąc, mówi, że myśmy dziwnie zamilkli. Pan premier poszedł do pana Mariusza Kamińskiego i powiedział mu, żeby jednak czegoś poszukał. Cytuję tygodnik „Najwyższy Czas!”: w ramach sprawy Sputnik inwigilowano konfederatów, członków ich rodzin, asystentów i związane z nimi osoby. Chodziło o znalezienie czegokolwiek, czym można byłoby uprawdopodobnić powiązania z Rosją. Czyli akcja z góry, na polityczne zlecenie. Nigdy się pan minister nie wytłumaczył z tego, co podsłuchiwał, co tam nagrał i jakim prawem to robił. Po drugie, wybory kopertowe. Mafijne zarządzanie na gębę, zmuszanie kolejnych instytucji do udziału w tej bezprawnej hucpie.

Raport NIK jest miażdżący, nie pozostawia wątpliwości, że rząd - w tym minister Kamiński - z pełną świadomością działał bezprawnie. Po trzecie, Policja dwóch prędkości. Powolna, bierna, nieudolna wobec lewicowych zadym w całym kraju, a prowokacyjna, nadgorliwa, agresywna w stosunku do demonstracji przeciw terrorowi sanitarnemu, wobec marszów niepodległości i tym podobnych demonstracji. Bo to nie są komunikaty z alternatywnej rzeczywistości, jak pan poseł Kierwiński opowiada, że demonstracje były brutalnie pacyfikowane - było dokładnie odwrotnie.

Zwykły obywatel, jak przejdzie w niedozwolonym miejscu przez jezdnię, to dostaje mandat, a ci ludzie blokowali ulice w całym kraju. I Policja pilnowała, żeby kierowcy tam czasem nie podjechali, legalnie mający prawo korzystać z tej drogi. To po czyjej stronie wy jesteście? W Katowicach pod katedrą stał po jednej stronie wyjący z nienawiści tłum żądny krwi nienarodzonych, z drugiej strony garstka ludzi, którzy bronili katedry. Kto jest wzywany na Policję?

Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne powinien być czysty jak łza, absolutnie bez zarzutu. Nie mam najlepszych wieści dla pana ministra - ciężar każdego z tych zarzutów jest tak poważny, że każdy z nich z osobna mógłby stanowić podstawę wniosku o odwołanie. Zacznijmy od wyborów kopertowych. To historia działania poza prawem. Jednym z bohaterów jest właśnie minister Kamiński, jednak korzeni musimy szukać wiele lat wstecz. W 2015 r. Mariusz Kamiński został przez sąd uznany za winnego przekroczenia uprawnień. Wyrok nie był prawomocny, ale wtedy pan prezydent Andrzej Duda uznał, że resocjalizacja nie jest potrzebna i pana ministra Kamińskiego ułaskawił. Dziś widzimy, jak wielki to był błąd. Bo minister Kamiński nie wyciągnął absolutnie żadnych wniosków. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, rząd, próbując obejść Państwową Komisję Wyborczą, działał poza granicami prawa, łamiąc i depcząc konstytucję, która mówi wprost, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Żaden przepis nie upoważnia kogokolwiek do zastąpienia Państwowej Komisji Wyborczej. To istota demokracji i wolnych wyborów, panie ministrze. W Polsce wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza, a nie samozwańcza grupa ministrów. Ale to nie wszystko w tej sprawie. Jak wskazuje ten raport, wszystkie polecenia były wydawane ustnie. Dziś pytamy, które organizacje tak robią, że wszystko jest na gębę, że bez żadnych dowodów. Czy tak postępuje minister konstytucyjny, panie ministrze Kamiński? Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, jak potężna jest ta afera Prawa i Sprawiedliwości - ponad 56 mln zł szkody. Wielka szkoda finansowa wyrządzona Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 56 mln zł, panie premierze, to jest skala tej afery. Panie ministrze Kamiński, był pan członkiem grupy, która do tej afery doprowadziła. Już samo to wystarczy, żeby odwołać pana z tego stanowiska. Ale oczywiście to nie wszystko. Kolejna rzecz to nadzór nad podległymi służbami.

Pan minister nie uznał za stosowne odpowiednio reagować, kiedy dochodziło do nieadekwatnego zachowania służb wobec osób, które wyrażały swoje poglądy, korzystając z praw wyrażonych choćby w art. 54 konstytucji. Wszyscy widzieli agresywne grupy bijące kobiety, młodzież, przedsiębiorców, a po czasie okazywało się, że to są nieoznaczeni funkcjonariusze. Widzieliśmy skandaliczną agresję wobec posłów. Widzieliśmy, kiedy inwigilowano nastolatków i agresywnie nachodzono ich w domach. Upolitycznił pan, panie ministrze Policję, a funkcjonariusze dzisiaj wstydzą się za to, co pan zrobił. Panie Ministrze! Okna pańskich gabinetów zwrócone są za bardzo na wschód, bo to są właśnie tamte wzorce. Tak że to wystarczy, aby zagłosować za pańskim odwołaniem. Wcale nie mniej ważna, ponieważ uderzająca w sedno naszej tożsamości. Kierowany przez pana resort chciał pozbawić strażaków ochotników godności strażaka. I nie ma w sprawie OSP większego grzechu niż uderzyć w te tradycje pielęgnowane od dziesiątek lat. Panie Ministrze! Stara polityka, skompromitowana polityka. Panie ministrze, nie chcemy takiej polityki. My chcemy polityki uczciwej. Chcemy polityki, której historia pisana jest z troską o obywatela, a nie o partyjny układ. Chcemy polityki, w której konstytucja jest dokumentem wyznaczającym zasady postępowania, a nie pustym prawem napisanym, żeby go nie przestrzegać. Niestety, panie ministrze, prawdopodobnie dziś koledzy pana obronią. Obronią, ponieważ jest pan gwarantem, że ta władza będzie trwać. Jedni się pana boją, inni dzięki panu mogą robić to, co uznają za stosowne. Jest pan gwarantem tego, że niewygodne dla rządu fakty zebrane przez podległe służby nie ujrzą światła dziennego. Jednak Polacy zasługują na ministra, dla którego najwyższą wartością jest dobro państwa i dobro obywateli, a nie dobro partii. Przed chwilą wykazałem, panie ministrze, że pan rażąco nie spełnia tego warunku. Nie spełnia pan tego warunku i nie powinien pan piastować funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o zabranie głosu ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Skoncentruję się na sprawach bezpośrednio związanych ze złożeniem wniosku o wotum nieufności. Nie zamierzam odpowiadać na żadne ataki personalne wobec mojej osoby. To jest wasze prawo. To jest kwestia kultury osobistej i kultury politycznej. Jestem również koordynatorem służb specjalnych, ale dzisiaj rozmawiamy o funkcji ministra spraw wewnętrznych w kontekście wyborów, które nazywacie wyborami kopertowymi, a które tak naprawdę były próbą ratowania Polski przed kryzysem, jaki nam groził. Szanowni Państwo! Chcę wyjaśnić pewne mity związane z działaniami ministra spraw wewnętrznych, z działaniami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i z decyzją pana premiera, który powierzył podległej mi spółce pewne zadania. 16 kwietnia 2020 r. pan premier Morawiecki wydał decyzję polecającą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych podjęcie zadania będącego realizacją przygotowań do wyborów korespondencyjnych w naszym kraju. Uważacie państwo, że była to decyzja nielegalna. Na mocy tej decyzji. Premier zobowiązał ministra spraw wewnętrznych do zawarcia umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych dotyczącą refundacji kosztów, jakie spółka miałaby ponieść w związku z realizacją tego polecenia. Istotą czynionego mi zarzutu w tym kontekście z waszej strony - czytałem uzasadnienie tego wniosku - jest to, zacytuję fragment waszego uzasadnienia. że jako minister spraw wewnętrznych nie dopełniłem ciążącego na ministrze spraw wewnętrznych i administracji obowiązku określonego w ww. decyzji premiera, polegającego na podpisaniu umowy i zapewnieniu refundacji kosztów poniesionych przez PWPW w związku z przygotowaniem wyborów prezydenckich, które się nie odbyły. Innymi słowy, żądacie państwo mojej dymisji, bo wedle was nie wykonałem nielegalnej waszym zdaniem decyzji premiera. Sami przyznajcie, że jest to kompletny absurd, że jest to nonsens. A co by było, gdybym podpisał tę umowę? Znając wasze wyrafinowanie polityczne, jestem całkowicie przekonany, że czytałbym w uzasadnieniu zarzut, że przekroczyłem swoje uprawnienia, podpisując umowę będącą nielegalnym poleceniem premiera. Czyli niezależnie od tego, czy podpisałbym umowę, w wypadku gdybym podpisał umowę, stawialibyście mi zarzut przekroczenia uprawień. Gdy tej umowy nie podpisałem, a zaraz wyjaśnię dlaczego, stawiacie mi zarzut niedopełnienia obowiązków. Nie ma żadnej wartości tego typu argumentacja z waszej strony. Ale chcę wam powiedzieć jasno, bardzo jasno, że jestem przekonany, uważam i uważałem, że decyzja, jaką podjął pan premier Morawiecki, była decyzją w pełni legalną. i podjętą w poczuciu głębokiego interesu publicznego. Jeszcze raz chcę podkreślić, że w tamtym czasie groził nam dramatyczny kryzys konstytucyjny związany z niemożnością przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Skala pandemii w tamtym czasie w naszym kraju była duża, a nikt na świecie nie był w stanie przewidzieć, jak rozwinie się epidemia. Nikt. W czarnym scenariuszu groziła nam sytuacja, że nasze państwo pozostanie bez prezydenta: zakończy się kadencja funkcjonującego prezydenta, nie można przeprowadzić wyborów - nie ma w Polsce prezydenta. To była kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności, żeby podjąć działanie w imię demokracji, w imię tego, żeby obywatele wybrali głowę państwa. Taka była intencja premiera, taka była intencja rządu. Wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność. Chcę państwu powiedzieć, że jako minister spraw wewnętrznych, po otrzymaniu tej decyzji pana premiera, zwróciłem się do Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w jaki sposób zamierza zrealizować tę decyzję. Otrzymałem pisemny plan od zarządu, oceniłem go jako poważny i profesjonalny i chcę państwu powiedzieć jasno: Osobiście jako minister spraw wewnętrznych złożyłem podpis zatwierdzający działania planowane przez PWPW. Zamierzałem umowę podpisać.

Żeby wiedzieć, jakie to są koszty, musiałbym wiedzieć, czy będzie druga tura wyborów, bo taka ewentualność zawsze wchodzi w grę. Uważam, że było to działanie racjonalne. Zarząd PWPW miał gwarancję tego i miał promesę w postaci zatwierdzenia przeze mnie planu działania, że taka umowa będzie podpisana. Tu nie ma niczego nadzwyczajnego w tej sytuacji. Nie ma niczego nadzwyczajnego w tej sytuacji. Nie mogłem podpisać tej umowy, ponieważ wybory się nie odbyły, szanowny panie pośle. Nie odbyły się. I Sejm, Wysoka Izba podjęła decyzję, w drodze ustawy, że wszystkie koszty, które poniosły podmioty w związku z koniecznością przygotowań do wyborów korespondencyjnych, będą pokryte z budżetu Krajowego Biura Wyborczego, co też się stało w grudniu ub.r. Chcę zapewnić Wysoką Izbę, że podległa ministrowi spraw wewnętrznych spółka państwowa PWPW nie poniosła żadnych strat w związku z przygotowaniami do tych wyborów. Panie pośle, teraz ma głos pan minister. chcę powiedzieć państwu tak: Oczywiście mógłbym się odnosić do jakichś różnych mniej lub bardziej absurdalnych zarzutów, jak choćby zarzut pana posła Sośnierza, który gdzieś coś przeczytał w swojej gazetce, w swoim biuletynie „Najwyższy Czas”

Tak, taki Sputnik istnieje rzeczywiście. Mógłbym odnosić się do każdego z tych zarzutów, chociaż, tak jak mówię, w części nie dotyczą one ministra spraw wewnętrznych. Ale powiem państwu jedną rzecz: Państwo przytaczacie tutaj różnego typu medialno-polityczne incydenty tak naprawdę sprzed roku. Odwołujecie się do wydarzeń sprzed roku. Za chwilę będzie rocznica tych wydarzeń. Proszę państwa, rozmawialiśmy o tym w Sejmie, w komisji administracji, dostaliście szczegółowe informacje i od ministra, i od komendanta głównego Policji. Jeżeli po roku znowu przytaczacie te same medialno-polityczne incydenty. jako zarzut wobec ministra czy wobec polskiej Policji, to znaczy, że jesteście bezradni, to znaczy, że nie macie żadnych argumentów.

To jest brak elementarnej lojalności państwowej z waszej strony. To, że czasami są takie sytuacje jak chociażby ograniczenia pandemiczne, że Policja musi. egzekwować pewne ograniczenia, które nie są popularne społecznie. To, że Policja musi podejmować takie działania. jest dowodem na jej państwowe działania i państwowy charakter. I ataki na Policję są z waszej strony godne najwyższego pożałowania. Wstydźcie się za to. Chcę powiedzieć z trybuny sejmowej, w kontekście tych różnego typu głupich, niemądrych. i nielojalnych państwowo ataków, do funkcjonariuszy Policji. Za to, że musieliście wykonywać często obowiązki, które nie były popularne społecznie, ale które były niezbędne z punktu widzenia zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego - za to składam wam jako minister spraw wewnętrznych podziękowania. To wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia. I proszę nie komentować mojej odwagi czy mojego honoru.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj opozycja, chyba ze względu na to, że mamy rok olimpijski, postanowiła pobić rekord bezzasadnych wniosków o wotum nieufności. Trzy wnioski, które bardzo szybko można by właściwie zbyć jednym podstawowym argumentem o konieczności przeprowadzenia tamtych wyborów, i za chwilę do tego jeszcze nawiążę. Ale ponieważ padło tutaj bardzo wiele kalumnii, oskarżeń pod adresem pana ministra Kamińskiego, to do kilku zasadniczych kwestii chciałbym się odnieść. Otóż, po pierwsze, służby podległe panu ministrowi Kamińskiemu odegrały fundamentalną i bardzo pozytywną rolę w zabezpieczeniu życia społecznego w czasie największej tragedii ostatnich lat, COVID-19. Policjanci dbali o to, żeby utrzymać porządek publiczny w czasie, kiedy nielegalne demonstracje, podsycane zresztą z tej strony sceny politycznej, doprowadzały - bo to trzeba podkreślać, szanowni państwo - do wielu zgonów kilka tygodni później. Przecież jest rzeczą oczywistą, że wówczas organizowane demonstracje, w szczycie drugiej fali, prowadziły do wzajemnych zakażeń, a w ślad za tym, kilka tygodni później, do zgonów. To jest prawda, która powinna was kłuć w wasze serca.

bo one doprowadzały do zgonów. Ale Policja i służby graniczne także bardzo intensywnie działały nad utrzymaniem porządku w zasadniczych kilku sferach. Po pierwsze, służby graniczne bardzo przyczyniły się do tego, że powstrzymane zostały liczne fale przychodzące do nas z zagranicy, począwszy właśnie od tej marcowo-kwietniowo-majowej z zeszłego roku, poprzez drugą falę. To Straż Graniczna. Później Policja, która prócz utrzymania porządku publicznego weryfikowała to, czy osoby, które powinny być poddane kwarantannie, rzeczywiście się na kwarantannie znajdują. To setki tysięcy weryfikacji, działań dziennie, czasami setki tysięcy, szanowni państwo.

To służby podległe panu ministrowi Kamińskiemu bardzo wydatnie pomagały w opanowaniu tej strasznej zarazy, która nas rzeczywiście dotknęła. Ale, szanowni państwo, mówiliście, tutaj padały takie sformułowania: pałka teleskopowa, jakieś interwencje.

Otóż pamiętacie może akcję „Widelec”, którą „Gazeta Wyborcza” opisała jako skuteczną pacyfikację? na idei solidarności, ma czelność pisać, że to pacyfikacja. Otóż wiecie, co tam było robione podczas tej akcji „Widelec” Poczytajcie sobie zeznania tych ludzi, którzy zostali wtedy bestialsko pobici, bestialsko potraktowani przez, tak, policję i służby specjalne w waszych czasach, czasach waszych polityków. I wy ponosicie za to odpowiedzialność.

Tak było.

kiedy używaliście, rząd Platformy Obywatelskiej używał przeciwko górnikom broni gładkolufowej, armatek wodnych. I, drodzy rodacy, szanowni państwo, tę różnicę, rzeczywiście trzeba powiedzieć, powściągliwość w interwencjach. w porównaniu z tym, co robił rząd Platformy Obywatelskiej, trzeba zaznaczyć i trzeba mieć na uwadze. A może chcecie też przykładów, jak zachowują się policje: niemiecka, francuska, holenderska, belgijska? Podczas protestów żółtych kamizelek zginęło kilkanaście osób, 2 tys. osób było rannych. Skuci, w kajdankach, z rękoma do tyłu, leżący twarzą do ziemi kobiety i mężczyźni. Niemiecka policja. Konno wjeżdżający policjanci holenderscy. To chyba daleko bardziej brutalne interwencje ze strony tamtej policji. W tej trudnej, dramatycznej sytuacji minister Kamiński starał się znaleźć złoty środek, po to żeby zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków. Ale chcę też panu ministrowi Kamińskiemu podziękować z tego miejsca za coś jeszcze. To jest wielka zasługa pana ministra Kamińskiego, [[Oklaski]] pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - w tamtym czasie powołana służba. Wtedy rzeczywiście zaczęliśmy żyć w innym kraju, ponieważ ta zmora III Rzeczypospolitej, jaką była korupcja, przynajmniej w bardzo znacznym stopniu została ograniczona. To jest wielka zasługa tego, co pan minister Kamiński całe życie robił. Pan minister Kamiński jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, przede wszystkim państwowcem. Wiem, że to słowo rzadko pada z waszych ust, nie bardzo jesteście w stanie je zrozumieć, ale, szanowni państwo, pan minister Kamiński dba o jakość instytucji, o to, żeby życie publiczne było jak najbardziej uczciwe. Tego możecie być pewni.

Powinniśmy lepiej się zabezpieczać w sensie prewencji, jeśli chodzi o różnego rodzaju nielegalne demonstracje, potrafić interweniować, ale deficyty, które musimy nadrabiać na skutek tej wielkiej zapaści, jaką było traktowanie państwa jak piątego koła u wozu, jak nocnego stróża co najwyżej w czasach rządów liberałów, neoliberałów, to deficyty, które trzeba nadrabiać latami. Co do wyborów, szanowni państwo, do których jeszcze się odniosę za chwilę podczas dyskusji nad pozostałymi dwoma wnioskami, chcę powiedzieć, że pan minister Kamiński zachował się również jak państwowiec, ponieważ wybory i wybory prezydenckie to jest obowiązek konstytucyjny.

Trzeba mieć odwagę i determinację, aby realizować konstytucję, szanowni państwo. Tak, niech żyje konstytucja. Dlatego, szanowni państwo, bardzo dziękuję panu ministrowi Kamińskiemu za to, że rok temu uczynił to, co trzeba było, to, co do niego wtedy należało, żeby te wybory mogły się odbyć, choć nie odbyły się. Jeszcze do tego nawiążę z innych względów podczas mojego kolejnego wystąpienia, natomiast chcę podziękować z tego miejsca za działania zdecydowane, odważne, ale zarazem rozważne służb podlegających panu ministrowi, a także za jego wspomnianą tutaj drogę życia, którą, owszem, warto w tym miejscu przypomnieć, bo to jest ważna dyskusja nad panem ministrem Kamińskim. To też powinniście mieć na uwadze, kiedy dyskutujecie o jego osiągnięciach, jego determinacji, jego działaniach.

Wiecie doskonale - także ta strona sali sejmowej - że pan minister Kamiński dobrze wypełnia swoje obowiązki. Pan minister Kamiński stara się nadrabiać, redukować te wszystkie deficyty, do których bardzo często wy niestety doprowadziliście. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Aktywów Państwowych - Jacka Sasina (druki nr 1262 i 1302)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiamy dziś akt oskarżenia wobec ministra aktywów państwowych pana Jacka Sasina, który zasiada tutaj obok. Akt oskarżenia powinien być odczytany przed niezawisłym sądem przez niezależnego prokuratora i tak byłoby w każdym demokratycznym państwie.

Jacek Sasin jest ministrem tego rządu, to jest jasne, ale jest też jego symbolem. Wiemy, że cokolwiek powie, jest na opak, dokładnie jak w rządzie Morawieckiego. Jak państwo mówią, że będzie obniżka podatków, to wiemy, że podatki będą podwyższone. Jak mówiliście, że z TVP zrobicie polską BBC, to wiemy, co się z tym stało. Jak mówiliście, że naprawicie Trybunał Konstytucyjny, to wiemy, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie działa. Ten rząd jest symbolem marnotrawstwa, symbolem partactwa, ale jest też symbolem korupcji. Dlatego, że pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, odpowiada za każdego nominata partyjnego, który zasiada w spółkach Skarbu Państwa. I mam dla państwa, drodzy posłowie i panie posłanki z PiS-u, prośbę i zadanie. Proszę, żeby rękę podniósł każdy, kogo rodzina, bliscy nie pracują w spółce Skarbu Państwa. Teraz po kolei. Córka posła Cymańskiego - tam jest pan poseł Cymański - Energa. Syn posła Smolińskiego - Energa. Brat poseł Golińskiej - jest pani poseł Golińska - Energa. Prezes. Szwagierka ministra Sasina - jest pan minister Sasin - lotnisko Lublin. Partnerka Daniela Obajtka - tu idziemy prawie na rekord - cztery rady nadzorcze. Cztery rady nadzorcze. Są lepsi. Żona posła Sobolewskiego - pięć rad nadzorczych. Pięć rad nadzorczych: Pekao, Anwil, lotnisko Goleniów, KGHM, Orlen Paliwa. Rzeczywiście rekord.

Na koniec partnerka europosła Tarczyńskiego - rada nadzorcza spółki zajmującej się produkcją maszyn pneumatycznych. To wszystko z waszej nominacji, to zasługa ministra Jacka Sasina. Szanowni państwo, jak w soczewce widzimy, że nie żyjemy w normalnym kraju. Wy proponowaliście Nowy Ład, ale to na pewno nie jest polski ład. To, co proponujecie, te wszystkie nominacje, minister Czarnek, minister Sasin - to jest wasz nowy ład. W każdym normalnym państwie - w każdym - Jacek Sasin wraz z ministrami zasiadłby na ławie oskarżonych, dlatego że wydał 70 mln na wybory, które się nie odbyły. Panie Ministrze Sasin! Czy pan wie, jak o panu mówią? Mówią o panu odwrócony Midas. Na pewno nie zamienia się w złoto. To jest wasza dewiza. To się stało waszą dewizą i waszym mottem, waszym działaniem każdego dnia. Sprawdźmy na przykładzie Jacka Sasina, jak to wygląda. No to sprawdźmy. Co mówił pan Jacek Sasin o kontroli NIK w sprawie wyborów kopertowych? Szanowni państwo, tu jest wynik kontroli i jest napisane tak: działania ministra Sasina były pozbawione podstawy prawnej.